Wysoka Izbo! Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji: - Infrastruktury - godz. 9.30, Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach - godz. 9.30, - Finansów Publicznych - godz. 10, - Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 10, - Administracji i Spraw Wewnętrznych - godz. 15, - Spraw Zagranicznych - godz. 15, - Zdrowia - godz. 15, - do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - godz. 15.30, - Obrony Narodowej - godz. 16, - Polityki Senioralnej - godz. 16, - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 17. Ponadto w dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Samorządami Gmin, Powiatów i Województw - godz. 14. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Przypominam, że postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 6 minut. Prawo do postawienia pytania dodatkowego przysługuje wyłącznie posłowi zadającemu pytanie. Dodatkowe pytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a uzupełniająca odpowiedź nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Pierwsze pytanie zadają posłowie Jarosław Gonciarz, Wojciech Szarama, Gabriela Masłowska i Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość, w sprawie reformy i reorganizacji parków narodowych - do ministra klimatu i środowiska. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Pani Minister! Rola parków narodowych, których mamy 23, jest w dzisiejszych realiach nie do przecenienia i są one niezastąpione. Parki zajmują wprawdzie niewielką powierzchnię naszego kraju, jednak swoją działalnością wpływają na postrzeganie waloru przyrodniczego całego kraju. Obecnie parki narodowe będące z punktu widzenia organizacyjno-finansowego odrębnymi jednostkami natrafiają na problemy z wykonaniem swoich budżetów z różnych przyczyn losowych. Dodatkowo aktualne rozwiązania prawne dotyczące funkcjonowania parków narodowych nie przewidują najlepszej zachęty dla samorządów w zakresie wyrażania woli co do tworzenia parków na swoim terytorium. W związku z powyższym pragnę zapytać, czy ministerstwo zamierza rozpocząć prace nad rozwiązaniami, które usprawnią organizację i zarządzanie parkami narodowymi, np. poprzez stworzenie jednostki prawnej mającej do dyspozycji dodatkowe środki finansowe na swoją działalność i nowe narzędzia prawne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na pytanie odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pani minister Małgorzata Golińska. Wysoka Izbo! Faktycznie parki narodowe to nasza najwyższa forma ochrony przyrody, ale też miejsce, gdzie poza ochroną różnorodności biologicznej możemy obserwować procesy naturalne. To jest niezwykle ważne dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z intensywnymi zmianami klimatu, bo te nasze parki narodowe mogą być doskonałym miejscem obserwacji, z którego później korzystają m.in. leśnicy.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska już toczą się prace nad projektem zupełnie nowego aktu prawnego, który jeszcze nie funkcjonuje w porządku prawnym naszego kraju, a mianowicie nad ustawą o parkach narodowych. Lasy mają swoją ustawę, leśnicy mają swoją ustawę, a parki narodowe, które chronią polskie dziedzictwo przyrodnicze, dotychczas takiej ustawy nie miały. A warto wskazać, że w tym roku obchodzimy 100-lecie funkcjonowania parków narodowych, bo przecież Białowieski Park Narodowy, który formalnie został powołany do życia w 1932 r., wcześniej zaczął funkcjonować jako rezerwat, specjalna jednostka - właśnie w 1921 r. Więc to jest ten czas - myślę, że najwyższy czas - kiedy powinniśmy pochylić się nad problemami związanymi z funkcjonowaniem parków.

Dzisiaj chcemy poprawić nadzór nad funkcjonowaniem parków, chcemy utworzyć jeden podmiot: polskie parki narodowe, w skład którego będą wchodziły dyrekcja polskich parków narodowych i 23, nazwijmy to, oddziały regionalne.

Warto wskazać, że dzisiaj te 23 odrębne jednostki prawne nie mogą się nawet finansowo wzajemnie wspierać. W ramach jednej instytucji polskich parków narodowych doprowadzimy do sytuacji, w której parki będą mogły się wspierać finansowo. Mało tego, utworzymy fundusz rezerwowy, który będzie przeznaczany właśnie na wspomaganie tych parków narodowych, które są w trudniejszej sytuacji finansowej albo które się znalazły w sytuacjach kryzysowych, jak chociażby Biebrzański Park Narodowy w zeszłym roku w trakcie historycznie dużego pożaru. Będą mogły również wspierać wspólne przedsięwzięcia polskich parków narodowych, bo nawet dzisiaj niestety każdy z parków na własną rękę prowadzi różnego rodzaju działania przyrodnicze, nie wiedząc, że jego kolega działa w podobnym temacie. Na pewno to, o czym pan poseł mówi, jeśli chodzi o samorządy, czyli wsparcie i zrozumienie społeczności lokalnych dla tworzenia i powiększania istniejących parków narodowych, to jest temat, który wywołuje największe zainteresowanie i kontrowersje. Stąd w naszym projekcie będziemy chcieli zmienić sytuację dotyczącą ustalania granic nowego parku narodowego, tak aby w przepisach przewidziano partycypację samorządów lokalnych. Postawimy bowiem również zadania po stronie państwa, co oznacza, że jeśli będziemy chcieli utworzyć park narodowy, to rząd będzie musiał przedstawić strategię rozwoju regionu, w którym będzie nowy park, ze wskazaniem źródeł finansowania. Mamy nadzieję, że zniweluje to obawy samorządów o to, że wraz ze stworzeniem parku narodowego zostanie u nich zahamowany rozwój i że w związku z tym będą tracić finansowo.

Dzisiaj parki narodowe są finansowane w większości ze środków zewnętrznych, bo dotacja z budżetu państwa pokrywa zaledwie 1/3 potrzeb parków narodowych, a w wielu z nich ta dotacja nie wystarcza nawet na podstawowe funkcjonowanie, to znaczy nawet na wynagrodzenia dla pracowników.

To też będziemy chcieli zmienić, zresztą decyzją pana premiera już od kolejnego roku dotacja będzie zwiększona i zamiast 1/3 potrzeb parków (Dzwonek) będziemy pokrywać blisko 50% ich zapotrzebowania. Bardzo proszę pana posła Gonciarza o dodatkowe pytanie. Szanowna Pani Minister!

Czy nowe projektowane przepisy będą wpisywać się w tę unijną strategię? Dziękuję. Bardzo proszę panią minister o odpowiedź na pytanie. Dokument strategia do spraw ochrony różnorodności biologicznej to jest dokument nieformalny, nieobowiązujący jeszcze, przedstawiony jako komunikat Komisji Europejskiej z maja 2020 r. To jest dokument, do którego Polska przygotowała swoje stanowisko, i choć generalnie popieramy cele zapisane w tym dokumencie związane z ochroną różnorodności biologicznej, to w wielu miejscach kwestionujemy drogę, którą przestawia Komisja do osiągnięcia tych celów.

W związku z tym to jest temat, który jest dla nas zupełnie bezpieczny. Mało tego, możemy chwalić się i pokazywać kolegom z innych państw, jak skutecznie chronić przyrodę. Wyzwaniem jest ten zapis dotyczący 10% ochrony ścisłej, po pierwsze dlatego, że nie jest zdefiniowane, w jaki sposób tę ochronę ścisłą rozumieć. W Polsce mamy bardzo radykalne podejście. To oznacza, że nie można podejmować żadnych działań na terenie, który jest objęty tą ochroną. Natomiast jest wiele państw, które ochronę ścisłą postrzegają mniej radykalnie i dopuszczają tam pewne działania, które nie szkodzą. Ta dyskusja wciąż toczy się w trakcie spotkań grup roboczych z Komisją Europejską. Na ile parki narodowe i nasze działania wpisują się w strategię. My oczywiście, tak jak mówiłam, mocny nacisk kładziemy na ochronę różnorodności biologicznej i procesów naturalnych. O ile procesy naturalne możemy obserwować właśnie w trakcie ochrony ścisłej, o tyle nie każdy park narodowy w Polsce ma ochronę ścisłą jako dominującą. Są parki, gdzie wręcz konieczne jest podejmowanie działań, aby zachować przedmioty ochrony.

Wtedy będziemy wiedzieć, z jaką formą i z jak wysoką rangą ochrony mamy do czynienia, a także będzie nam łatwiej dyskutować z innymi państwami (Dzwonek), które chwalą się np. większą powierzchnią objętą parkiem narodowym, a w konsekwencji wyjdzie nam, że nasze parki krajobrazowe i ich parki narodowe to jest ten sam poziom ochrony. Przystępujemy do drugiego pytania. Zadają je posłowie Cezary Grabarczyk, Paweł Olszewski, Małgorzata Chmiel, Dariusz Joński, Maciej Lasek, Czesław Mroczek, Paweł Papke, Grzegorz Rusiecki, Krystyna Sibińska, Franciszek Sterczewski i Krzysztof Truskolaski z Koalicji Obywatelskiej, w sprawie problemów z funkcjonowaniem systemu elektronicznego poboru opłat - do prezesa Rady Ministrów. Pierwsze pytanie zadaje pan poseł Cezary Grabarczyk. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Od 1 grudnia jedynym systemem, który obowiązuje na polskich autostradach, jeśli chodzi o opłaty za przejazd wybranymi odcinkami autostrad płatnych, jest system e-TOLL. To system, co do którego rząd zapewniał, że będzie lepszy, że będzie dźwignią postępu, że spowoduje upłynnienie ruchu na polskich autostradach. Okazuje się, że to były zapowiedzi na wyrost. Mamy coraz więcej sygnałów o problemach z wdrażaniem tego systemu. Aplikacja, którą chwalił się resort finansów, nie działa. To jest bardzo częsty komunikat: nieaktywna obsługa w aplikacji, która została udostępniona kierowcom. Mamy coraz częściej sygnały, że autostrady w miejscach, w których rozpoczyna się płatny odcinek, stają się wielkimi parkingami, co tworzy zagrożenie dla ruchu na drogach szybkiego ruchu. Dlaczego parkingi? Dlatego że aplikacje się zawieszają, nie ma możliwości poniesienia opłaty za przejazd. Czy to jest do wyeliminowania? Czy polscy kierowcy tuż przed świętami będą mieli pewność, że bezpiecznie dotrą na spotkania rodzinne? Czy wpływy z nowego systemu są wyższe niż z systemu via-TOLL? Jaka jest wysokość kar?

Bardzo proszę, na pytanie odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan minister Mariusz Gojny. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Dziękuję za zadanie pytania, panie pośle. Na początek chciałem przedstawić parę uwag ogólnych. Dobrze, dziękuję.

Nowy system został stworzony w oparciu o architekturę umożliwiającą jego modyfikację i rozbudowę, dlatego w trakcie jego wdrażania, jak i obecnie, w trakcie użytkowania, modyfikujemy go i rozwijamy jego funkcjonalności. Wystarczy wymienić chociażby z sukcesem wprowadzoną, nową i bardziej intuicyjną aplikację e-TOLL PL Bilet do zakupu e-biletu bez konieczności logowania, z możliwością płatności różnymi metodami, w tym także blikiem. Biorąc pod uwagę przyrost liczby kilometrów dróg szybkiego ruchu w Polsce, możemy zakładać rozszerzenie sieci płatnych dróg o kolejne 1400 km. To pokazuje skalę oszczędności dla państwa. W poprzednim systemie te pieniądze były wydawane na stawianie bramownic wyposażonych w radiowy system przekazu danych, co było realizowane przez zagraniczną firmę. Dziś te środki przeznaczane są na nowe drogi i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowy system e-TOLL jest odpowiedzią na konieczność wymiany działającego w Polsce od 2011 r. elektronicznego systemu poboru opłat via-TOLL. Poprzednie rozwiązanie bazowało na radiowym przekazie z urządzeń pokładowych OBU/ZSL zamontowanych w pojeździe, z ok. 950 fizycznych bramownic, skąd dane po ich agregacji były przekazywane do systemu informatycznego.

Dlatego wsłuchujemy się w głosy kierowców i dostosowujemy nasze działania do ich potrzeb.

Do tej rewolucji dołączyli chętnie również nasi partnerzy biznesowi. Partnerzy, widząc potencjał biznesowy w obsłudze takiego klienta e-TOLL, wdrożyli nowe rozwiązanie i obecnie oferują usługi wnoszenia odpłatności za drogi. Rozwijamy też sieć partnerską, prowadzimy zaawansowane rozmowy z kolejnymi sieciami stacji paliw.

Istotą systemu jest pobór opłat, a nie nakładanie sankcji.

Jeżeli chodzi o liczbę kontroli wykonanych od 1 października, to takich kontroli było 22 tys., w tym kontroli wynikowych 1325, w tym na autostradach - 13 tys. kontroli, w tym wynikowych - 1039.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie do pana zadaje pan poseł Maciej Lasek.

Pani Marszałek! Panie Ministrze!

Przykładowe opinie: pobrałem aplikację, doładowałem konto, przejechałem odcinek płatny, taki, za który do tej pory płaciłem, i nic, inna: daję 1 gwiazdkę, bo mniej nie można, zawiesza się ona na najnowszym telefonie, kolejna: przechodzę przez cały system wchodzenia w tę aplikację, czyli wstawiania nowych informacji, odpowiadam na mnóstwo pytań, na końcu wszystkiego pojawia się błąd.

Ministerstwo Finansów odpowiada: proszę zakupić bilet. Już wtedy zapewniano nas, pani minister zapewniła nas, że do 1 grudnia wszystkie zgłoszone problemy zostaną usunięte, jednak tak się nie stało. Panie ministrze, ile kosztowało polskiego podatnika opracowanie i wdrożenie tak nieudanego programu? Czy to było robione w Ministerstwie Finansów, czy to jest program, który został przygotowany na zlecenie? Mam również pytanie, do kiedy wszystkie te poważne zastrzeżenia, które możemy znaleźć w sieci, zostaną usunięte.

Bardzo bym prosił o odpowiedź na piśmie. Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie pana ministra Mariusza Gojnego.

Jeżeli chodzi o kwestię systemów informatycznych, to były one budowane przez spółkę celową Aplikacje Krytyczne, czyli spółkę, która pracuje na rzecz Ministerstwa Finansów. Jeżeli chodzi o kwestię jakości tego systemu, to cały czas wsłuchujemy się w głosy kierowców i dostosowujemy te nasze działania do potrzeb kierowców.

Dziękuję bardzo. Przechodzimy do trzeciego pytania, które zadaje grupa posłów: Krzysztof Gawkowski, Wanda Nowicka, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Beata Maciejewska, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Wiesław Buż, Jan Szopiński, Przemysław Koperski, Małgorzata Prokop-Paczkowska, Katarzyna Kotula, Paweł Krutul, Marcelina Zawisza, Rafał Adamczyk, Monika Falej, Robert Obaz, Katarzyna Ueberhan, Maciej Kopiec, Krzysztof Śmiszek, Paulina Matysiak, Wiesław Szczepański, Tadeusz Tomaszewski, Dariusz Wieczorek, Tomasz Trela, Marcin Kulasek, Joanna Scheuring-Wielgus, Anna Maria Żukowska i Anita Sowińska z klubu Lewica.

Pytanie skierowane jest do ministra zdrowia. Bardzo proszę, pani poseł. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 20 grudnia w warszawskim Szpitalu Bielańskim mazowiecka konsultantka ds. ginekologii i położnictwa dr Barbara Pietrzak przeprowadzi kontrolę dotyczącą liczby ciąż oraz przypadków terminacji ciąży. Zamierza skontrolować rejestr zabiegów ginekologicznych, rejestr odmów oraz historie chorób związane z przerwaniem ciąży. Kontrola obejmuje również dane dotyczące porodów, ciąż donoszonych i przedwczesnych oraz liczby ciąż obumarłych. W związku z ogromnym i uzasadnionym niepokojem ze strony lekarzy, którzy czują się zastraszeni - wszyscy pamiętamy śmierć pani Izabeli z Pszczyny - i którzy obawiają się, że kontrola szpitala może wywrzeć na nich presję, by ciąż nie przerywali, a także z uwagi na przerażenie ze strony kobiet, które chciałyby skorzystać z usług szpitala, proszę o odpowiedź na następujące pytania: Dlaczego jest przeprowadzana kontrola w Szpitalu Bielańskim? Czy były jakieś skargi czy sygnały, że w szpitalu są jakieś nieprawidłowości? Jeśli tak, to kto je zgłaszał, pacjentki czy jakieś organizacje, na przykład Ordo Iuris? Jaka jest podstawa prawna tej kontroli? Jaki jest cel kontroli dotyczącej właśnie przerywania ciąży? Lekarze obawiają się, że kontrola ma zniechęcać ich do przerywania ciąż zgodnie z prawem, wzbudzając w nich niepokój i obawy przed represjami. Czy chodzi o to, aby poprawić dostępność świadczeń z zakresu legalnej aborcji, czy aby ograniczyć dostęp do zgodnych z prawem zabiegów? Czego tak bardzo obawiają się pacjentki? Kiedy będzie raport pokontrolny? Proszę o przesłanie raportu pokontrolnego, jak tylko zostanie sporządzony. Szpital Bielański zapewnia szeroki zakres świadczeń medycznych z zakresu ginekologii i położnictwa. Dlaczego kontrola dotyczy wyłącznie kwestii związanych z przerywaniem ciąży? Ministerstwo twierdzi, że jest to rutynowa kontrola, zatem proszę o informację, w których szpitalach w województwie mazowieckim pani konsultantka (Dzwonek) przeprowadziła kontrole w ostatnim roku i jaki zakres świadczeń obejmowały te rutynowe kontrole? Czy rutynowe kontrole przeprowadzone w Szpitalu Bielańskim i innych szpitalach obejmowały wymienione świadczenia medyczne, a jeśli tak, to w których szpitalach? Już kończę, pani marszałkini. leczenie schorzeń z zakresu endokrynologii ginekologicznej, leczenie schorzeń ginekologicznych u pacjentek z chorobą zakrzepowo-zatorową, leczenie nieletnich z problemami ginekologicznymi, onkologia ginekologiczna, terapia wad płodu, np. uropatia zaporowa i inne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Piotra Brombera o odpowiedź na te pytania.

Pani Marszałek! Panie Panowie Posłowie! Szanowna Pani Poseł! Zapowiedziana z dużym wyprzedzeniem kontrola w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, która ma odbyć się, tak jak pani poseł poinformowała, 20 grudnia tego roku, nie jest kontrolą zlecaną przez ministra zdrowia ani przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zgodnie z art. 11 ww. ustawy do zadań konsultantów krajowych i konsultantów wojewódzkich należy m.in. kontrola dostępności świadczeń zdrowotnych. Przepisy ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia umożliwiają zlecenie przez konsultanta krajowego konsultantowi wojewódzkiemu wykonania określonego zadania mieszczącego się w zakresie zadań konsultanta wojewódzkiego. Informację o wydaniu takiego polecenia konsultant krajowy przekazuje ministrowi właściwemu ds. zdrowia oraz właściwemu wojewodzie. W przedmiotowym przypadku możliwe było zlecenie przez konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii wykonania kontroli w ww. podmiocie leczniczym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa mazowieckiego. W przedmiotowym przypadku informacja o zleceniu ww. kontroli została przekazana do wojewody mazowieckiego, natomiast do resortu zdrowia informacja ta została przekazana w trybie roboczym 10 grudnia br. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez konsultanta krajowego 17 listopada tego roku zwrócił się on z prośbą o przeprowadzenie kontroli w oddziale ginekologiczno-położniczym Szpitala Bielańskiego do konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa mazowieckiego, który z kolei zwrócił się z prośbą do Urzędu Wojewódzkiego o zlecenie kontroli obejmującej sprawdzenie jakości realizowanych - co podkreślam - przez rozważany podmiot świadczeń, zarówno dotyczących leczenia ciężarnych, jak i pacjentek z problemami ginekologicznymi, i dostępności, włącznie z poprawnością prowadzenia dokumentacji.

Przedmiotowa kontrola ma charakter standardowy. Zgodnie z wyjaśnieniami konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii kontrole dotyczące prawidłowości działania wybranych oddziałów szpitalnych są prowadzone rokrocznie na terenie wszystkich województw, w tym województwa mazowieckiego.

Celem żadnej kontroli nie jest straszenie kogokolwiek, wręcz przeciwnie, kontrola ma na celu sprawdzenie i poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.

Dlatego proszę o informację, jakie jest uzasadnienie prawne dla żądanego przez panią konsultant (Dzwonek) udostępniania całości dokumentacji medycznej pacjentek z okresu ponad 6 miesięcy. Dziękuję bardzo.

Panie i Panowie Posłowie! Szanowna Pani Poseł! Użyła pani również sformułowania „jakość” Te czynności, o których dzisiaj mówimy, które, podkreślam, są podejmowane z inicjatywy konsultanta krajowego i konsultant wojewódzkiej, wpisują się w kontrolę dostępności i jakości. Celem każdej kontroli jest weryfikacja jakości udzielonych świadczeń.

To doświadczenie, wykształcenie i podstawa formalnoprawna dają podstawę do przeprowadzenia tego typu czynności. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego pytania. Pytanie zadają posłowie Jacek Protasiewicz, Mieczysław Kasprzak i Marek Sawicki, Koalicja Polska, w sprawie negocjacji z Czechami w sprawie kopalni Turów oraz kar nałożonych na Polskę. Bardzo proszę, pierwsze pytanie, pan poseł Jacek Protasiewicz. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Jak niestety wiadomo, Polska jest w dwóch sporach formalnych, formalnoprawnych, w których nałożono na nią kary finansowe w związku z decyzjami czy działaniami podjętymi przez rząd polski.

Na dzisiaj suma kwot wynikających z kar nałożonych na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z tytułu tego sporu wynosi już ponad 40 mln euro. Jest to, z grubsza rzecz biorąc, już ponad 200 mln zł, są to realne straty dla naszego kraju, dla naszych obywateli, dla inwestycji finansowanych z unijnych środków, których jest bez liku w Polsce, albowiem nawet jeśli rząd polski ustami premiera Morawieckiego zapowiedział, że nie będzie tych kar płacił, to są to puste zapowiedzi. To są, że tak powiem, parole, parole, parole, które nic nie znaczą, bo te kwoty zostaną odciągnięte od przyznanych w budżecie 7-letnim Unii Europejskiej funduszy przeznaczonych na realizację inwestycji w Rzeczypospolitej Polskiej z dofinansowaniem środków europejskich. Tych środków zatem w ogóle nie będzie. Mamy więc już do czynienia z 50-dniowym urzędowaniem nowej pani minister, która zapowiedziała, że jej głównym celem, pierwszym celem będzie rozwiązanie sporu z Czechami. Od tej pory efektu nie ma (Dzwonek), a z tych 200 mln strat już dzisiaj realnych 106 mln, ponad 50%, przypada na okres rządzenia, funkcjonowania i negocjowania przez panią minister Moskwę porozumienia z rządem czeskim. Jaki jest stan tych negocjacji i jaka jest przyczyna braku porozumienia, które jest tak kosztowne dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, panie ministrze? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Panie Pośle! Wysoka Izbo! Dziękuję bardzo za pytanie. Odniosę się może najpierw do kwestii prawa unijnego, która została tutaj poruszona, do której odniósł się pan poseł na początku swojej wypowiedzi. Muszę podkreślić, że naruszenie w sprawie dostępu do sprawiedliwości, możliwości odwołania się od decyzji środowiskowych to jest naruszenie, które. Ta sprawa została zamknięta przez Komisję właśnie na początku grudnia dzięki ustawie, którą przygotowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska i która została przyjęta przez Sejm wcześniej w tym roku. Dopiero w tym roku, po 10 latach, udało się w końcu zamknąć sprawę tego naruszenia.

Pan poseł zapytał o przebieg negocjacji. Muszę podkreślić, że z niezwykłą intensywnością prowadziliśmy rozmowy.

Ściśle współpracujemy w gronie tych instytucji.

Czesi po prostu nie chcą się dogadać. Jeżeli nie ma woli po stronie czeskiej, to nic na to nie poradzimy. Mam nadzieję, że z nową panią minister uda się znaleźć dobre rozwiązanie dla rejonu.

Dziękuję bardzo. Drugie pytanie zadaje także pan poseł Jacek Protasiewicz. Z wielką życzliwością chciałbym przyjąć do wiadomości tę pana odpowiedź, ale mam wrażenie, że ona ilustruje stare polskie powiedzenie: złej baletnicy przeszkadza rąbek spódnicy. Najpierw był problem, jak mówiliście, wyborów.

Ostatnio sąd administracyjny orzekł bardzo wyraźnie, że ta koncesja została wydana z naruszeniem prawa, i nakazał konsultacje z organizacją Greenpeace. W związku z powyższym może trzeba zawiesić tę koncesję i poważnie potraktować rozmowy z Czechami, a nie mówić, że umywają ręce. Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź na to pytanie.

Ta kopalnia uzyskała decyzję środowiskową, która była przedmiotem konsultacji transgranicznych ze stroną czeską. I znowu Czesi nie dotrzymują zobowiązań, które podjęli w ramach tego protokołu. My nie możemy ich do tego zmuszać, ale cały proces konsultacji transgranicznych został przeprowadzony.

Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego pytania.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nie tak dawno, jakieś kilkanaście dni temu, została oddana do użytku bardzo ważna obwodnica, obwodnica Niemodlina. Na tę obwodnicę mieszkańcy Niemodlina, Opolszczyzny, ale też kraju czekali ok. 40 lat. Również nie tak dawno została oddana dzięki mocnemu zaangażowaniu, odpowiedniej wizji na to, w jaki sposób ma być realizowana infrastruktura na terenie Opolszczyzny, obwodnica Myśliny czy też obwodnica Nysy. Panie Ministrze! Mam pytanie, ponieważ w ramach „Programu budowy 100 obwodnic” czy też innych realizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury w realizacji są kolejne obwodnice. W sumie tych obwodnic na terenie województwa opolskiego jest dziesięć. Pozwolę sobie je wymienić. Jest to obwodnica Kędzierzyna-Koźla, obwodnica Praszki, obwodnica Olesna, w ramach „Programu budowy 100 obwodnic” są to też obwodnice Prudnika, Brzegu, Sidziny i Lędzin. Moje pytanie brzmi, na jakim etapie prac są wymienione przeze mnie obwodnice.

W ramach rezerwy znalazły się również dwie obwodnice, obwodnica Strzelec Opolskich i Namysłowa. Czy również te dwie obwodnice będą w najbliższych (Dzwonek) latach mogły być realizowane? Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Dziękuję za pytanie, które jest związane ze strategicznymi inwestycjami drogowymi w województwie opolskim. Na wstępie pragnę wskazać, że te inwestycje są realizowane w ramach dwóch programów, bardzo dużych, jeżeli chodzi o zaangażowanie rzeczowe i finansowe.

Zaznaczam przy tym, że „Program budowy dróg krajowych” został przyjęty w roku 2015, a pierwotne środki przeznaczone na jego realizację były dalece niewystarczające. Limit finansowy wydatków tego programu wynosił 107 mld zł, natomiast wartość łączna zadań w nich ujętych sięgała ponad 200 mld zł, czyli po przejęciu odpowiedzialności za inwestycje drogowe minister Andrzej Adamczyk miał do dyspozycji 107 mld zł, a inwestycji wpisanych do realizacji na 200 mld zł, niedobór wynoszący ponad 90 mld zł. Widząc to, podjął bardzo konkretne i skuteczne starania mające na celu podniesienie limitu finansowego. Dzięki przychylności kolejnych rządów Prawa i Sprawiedliwości, pani Beaty Szydło i pana premiera Mateusza Morawieckiego udało się podnieść wartość „Programu budowy dróg krajowych” do obecnej, tj. do 164 mld zł, przez co zadań w ramach tego programu realizowanych jest zdecydowanie więcej. Jedną z inwestycji, która jest realizowana dzięki nowym środkom, jest obwodnica Kędzierzyna-Koźla.

Umowa z wykonawcą, czyli firmą STRABAG, została podpisana 15 października 2018 r. Obecnie prowadzone są prace.

Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe obwodnice wymienione przez panią poseł Katarzynę Czocharę, czyli Prudnik, Sidzina i obwodnica Lędzin, to są one realizowane w ramach drugiego programu, tym razem stworzonego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli „Programu budowy 100 obwodnic” Dostrzegliśmy ogromne zapotrzebowanie na inwestycje dotyczące obejść miast i miejscowości leżących przy drogach krajowych i stąd dedykowany tym inwestycjom program inwestycyjny. Program ten został zapowiedziany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego jesienią 2019 r., a my jako Ministerstwo Infrastruktury od razu przystąpiliśmy do działania, w efekcie czego w tym roku 14 zadań jest w realizacji, jedno - w przetargu, a w przypadku wszystkich pozostałych trwają co najmniej prace przygotowawcze. Wartość tego programu to 28 mld zł. Program ten został stworzony, ponieważ prócz realizacji tak bardzo efektownych inwestycji autostradowych i ekspresowych chcieliśmy położyć duży nacisk na poprawę płynności, a także bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach, które nie znajdują się w ciągu dróg szybkich. Słuszność działań resortu podkreśla fakt, że oprócz konieczności budowy 100 obwodnic, które znalazły się na liście podstawowej i w przypadku których są zabezpieczone środki na realizację, zaistniała konieczność stworzenia dodatkowej listy, listy rezerwowej, obejmującej ponad 50 zadań. Zadania te będą możliwe do realizacji po wygenerowaniu oszczędności w ramach listy podstawowej. Taka sytuacja będzie dotyczyła też obwodnic, które znajdują się na liście rezerwowej, w województwie opolskim. O tych obwodnicach pani poseł też mówiła. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację tych zadań jest związane z decyzjami podejmowanymi w niedalekiej przeszłości przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. O zaawansowaniu budowy obwodnicy Kędzierzyna-Koźla na drodze krajowej nr 40 mówiłem. W przyszłym roku zostanie ona oddana do użytkowania.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Anna Kwiecień zadaje drugie pytanie skierowane do pana ministra. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Bardzo dziękuję za tę pierwszą część, za niezwykle wyczerpującą odpowiedź, ale mam pytanie. Chciałabym spytać, czy to w jakikolwiek sposób opóźnia realizację tych inwestycji.

Czy tutaj są jakieś opóźnienia, zagrożenia?

Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Szanowne Panie Poseł! Szanowni Państwo!

Jeżeli chodzi o obwodnicę Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46, to również w kwietniu br. została podpisana umowa na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

Szacowana długość to ok. 3 km.

Przechodzę do pytania pani poseł Anny Kwiecień o trudną sytuację pandemiczną, która dotknęła nas wszystkich w tych ostatnich kilkunastu miesiącach. Pomimo tej trudnej sytuacji pandemicznej nie mieliśmy do czynienia z zatrzymaniem prac inwestycyjnych w przypadku robót, inwestycji liniowych, zarówno drogowych, jak i kolejowych.

Tak że, co do zasady, nie mieliśmy większych problemów w trakcie pandemii. Mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach również tak będzie. Żeby pokazać determinację rządu w realizacji w tych zadań, powiem, że to właśnie w roku poprzednim, roku 2020, w czerwcu, na wniosek ministra infrastruktury pan premier Mateusz Morawiecki zdecydował o zwiększeniu środków „Programu budowy dróg krajowych” o 22 mld zł właśnie po to, żeby realizować kolejne zadania w tym trudnym pandemicznym czasie.

Posłowie Krzysztof Gadowski, Tomasz Piotr Nowak, Wojciech Saługa, Sławomir Neumann, Mirosława Nykiel, Paweł Poncyljusz i Urszula Zielińska, Koalicja Obywatelska, zadają pytanie w sprawie braku ustawowych zapasów węgla kamiennego dla elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni oraz ograniczenia dostępu dla indywidualnych odbiorców i drastycznego wzrostu cen węgla. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Polskę dotykają mrozy, raz mocniejsze, raz słabsze, a my jesteśmy zasypywani informacjami, że ponad 20 firm, spółek Skarbu Państwa, w dużej części elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, nie ma zabezpieczonych ustawowych zapasów. Po raz pierwszy w tym zestawieniu pojawiła się Elektrownia Kozienice.

Okazuje się, że nawet Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie pisze w tej sprawie do ministra.

Co z tym węglem, panie ministrze? Jakie kary do tej pory zapłaciły prezesowi URE te spółki, które nie zabezpieczyły środków? Gdzie ten węgiel? Już nie mówię o innych, tylko o tych ustawowych, minimalnych, które mają zabezpieczyć bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Dochodzą do nas głosy o reglamentowaniu sprzedaży węgla dla odbiorców indywidualnych. Co jest powodem tej reglamentacji?

Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, panie ministrze. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Panowie Posłowie! Zapasy węgla kamiennego, brunatnego oraz oleju opałowego w przedsiębiorstwach energetycznych gromadzone są na podstawie rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych. Zapasy węgla w przedsiębiorstwach energetycznych są na bieżąco monitorowane, w tym z urzędu przez prezesa URE.

W związku z sygnalizowanymi przez podmioty z sektora elektroenergetycznego problemami związanymi z utrzymaniem zapasów węgla na wymaganym poziomie strona rządowa podjęła działania mające na celu identyfikację przyczyn mniejszych zapasów węgla kamiennego. Teraz przedstawię przyczyny braku węgla energetycznego w dwóch przestrzeniach, tej, o której pan poseł był uprzejmy powiedzieć, tej komunalno-bytowej, a następnie tej zawodowej. Od początku jesieni obserwujemy bardzo wysoki popyt na węgiel energetyczny.

Wpłynęło to na decyzje klientów w zakresie robienia większych zapasów węgla na aktualny sezon grzewczy, 2021/2022.

Najmniejszy import węgla energetycznego można zauważyć w III kwartale br., kiedy to tradycyjnie robione są zapasy na zimę.

Oznacza to, że do Polski wjechało mniej o 1,12 mln t niż rok wcześniej w analogicznym okresie, co jest najbardziej odczuwalne przez podmioty zaopatrujące się do tej pory w importowany węgiel. Są to sytuacje nie do przewidzenia, ponieważ nie są znane plany prywatnych podmiotów chcących importować. Zarzuty podnoszone przez przedsiębiorstwa ciepłownicze i inne podmioty wykorzystujące węgiel energetyczny, miał, dotyczące braku dostępnego węgla pochodzą zasadniczo od podmiotów, które swoje potrzeby surowcowe w części lub w całości zaspokajały poprzez węgiel importowany, co przy jego obecnej niskiej dostępności i wysokich cenach stawia je w bardzo trudnej sytuacji. Polskie spółki górnicze mogą zrealizować ich zapotrzebowanie w drugiej kolejności, po podmiotach, z którymi posiadają zawarte wieloletnie umowy gwarantujące pewność ceny i dostaw.

Ilość węgla, która może zostać skierowana do osób, które opalają swoje domy węglem, jest pochodną całej produkcji węgla. Co do kwestii dotyczących braków na rynku energetyki węglowej, to wśród przyczyn niższych zapasów węgla w stosunku do wolumenu wymaganego rozporządzeniem należy wskazać bardzo wysoki poziom wykorzystania bloków węglowych przez operatorów sieci przesyłowych, a w konsekwencji zwiększenie produkcji energii elektrycznej w stosunku do planowanej produkcji w przeliczeniu rok do roku, zwiększoną produkcję energii elektrycznej ze źródeł węglowych.

Od początku II połowy roku Polska stała się eksporterem energii elektrycznej. Polska zaczęła eksportować energię do krajów sąsiadujących pomimo najwyższych w historii cen energii elektrycznej.

To są dane z przedziału styczeń-październik. Względem 2019 r. nastąpił wzrost o 17%. Bardzo proszę o zadanie drugiego pytania pana posła Tomasza Nowaka. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Ministrze!

Dlaczego w centralnym magazynie węgla w Wielkopolsce nie ma węgla?

Nie ma zabezpieczenia dla elektrowni.

Transformacja to jest coś, co nas czeka, i obawiam się, że niestety jeśli ona będzie robiona w ten sposób, a dzisiaj będziemy obradować nad ustawą, która ogranicza w tej chwili, likwiduje kopalnie, będzie zejście z tymi kopalniami. Bardzo proszę, panie ministrze, o odpowiedź na pytanie. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Ale po kolei. Właściwie drugiego czy trzeciego dnia urzędowania spotkałem się z problemem transportu węgla z kopalń do elektrowni.

Nie ma, tak jak powiedziałem, tragedii.

Bo żeby rozwiązać problem, który mamy dzisiaj, najprościej jest produkować więcej węgla.

Wpłynie to oczywiście na cenę prądu i konsekwencja tego będzie taka, że okej, dostaniemy nadwyżkę jakiegoś prądu od kogoś, nie: dostaniemy, ale kupimy, będziemy mogli kupić, ale za wyższą cenę, i też trzeba się z tym liczyć.

Na tym nam zależy, dlatego że bezpieczeństwo energetyczne ja osobiście rozumiem (Dzwonek) nie tylko jako przestrzeń zabezpieczenia tej energii, ale również zabezpieczenia ceny, która będzie dostępna dla każdego obywatela, i nie dojdzie tu do ubóstwa. Jeśli chodzi o kwestie dodatkowe dotyczące pana regionu, pozwoli pan, że odpowiem pisemnie już po wszystkim. Dziękuję, panie ministrze. Przechodzimy do siódmego pytania. Pytanie zadają posłowie Barbara Dziuk, Grzegorz Wojciechowski, Barbara Bartuś, Witold Czarnecki, Agnieszka Soin i Iwona Arent, klub Prawo i Sprawiedliwość, w sprawie realizacji rządowego programu „Polska cyfrowa” - skierowane do prezesa Rady Ministrów, ministra cyfryzacji. Bardzo proszę, pierwsze pytanie zadaje pani poseł Barbara Dziuk. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Program rządowy „Polska cyfrowa” jest to program bardzo istotny, ponieważ zapewnia budowę szerokopasmowej sieci do punktów adresowych stanowiących białe plamy na mapie dostępu do Internetu. Jest to o tyle istotne, ponieważ widzimy - i wynika to i z rozmów, i ze spotkań - że są oczekiwania zarówno samorządów, jak i osób prywatnych, aby to zadanie było jak najszybciej realizowane. Różne samorządy dają darmowy dostęp do Internetu i tutaj synchronizowanie działań rządowych i samorządowych jest bardzo istotne.

Chciałabym zapytać pana ministra, jak wygląda kwestia organizowania konkursów, na jakich płaszczyznach jest to ustalane, jakie są przewidziane kwoty do uzyskania przez samorządy, ale też przez inne jednostki, przez organizacje pozarządowe. Myślę, że wspólnie powinnyśmy działać, aby wyeliminować białe plamy na mapie, ale też rozszerzyć zasięg telefonii komórkowej w tych miejscach, gdzie jest Polska powiatowa, biedniejsze samorządy.

Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Szanowna Pani Marszałek! Państwo Parlamentarzyści! Na wstępie chciałbym podziękować za to pytanie państwu parlamentarzystom, ja niewątpliwie także się zgadzam z tezą postawioną w tym pytaniu.

Szanowni Państwo! Jeśli chodzi o doposażanie np. jednostek samorządu terytorialnego w sprzęt komputerowy, szkolenia dla pracowników, szkolenia dla pracowników jednostek podległych, zakup sprzętu również dla jednostek podległych, zakup oprogramowania czy też kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, to w tym roku uruchomiliśmy program „Cyfrowa gmina”

Ten audyt pokaże, w jakim zakresie dana jednostka samorządu terytorialnego powinna poprawić swoje bezpieczeństwo w sieci, w zakresie korzystania z serwerów, z rejestrów, oczywiście z e-usług, które także każdy samorząd wprowadza. To w skali naszego państwa, myślę, będzie bardzo dobrym krokiem.

Jeśli chodzi o dostęp do szybkiego, szerokopasmowego Internetu, to nadrobiliśmy także mocno zaległości związane z cyfryzacją szkół w ramach wdrażania ogólnopolskiej sieci edukacyjnej OSE.

Dostęp do szybkiego Internetu, w 90% światłowodowego, otrzyma łącznie ponad 2 mln gospodarstw domowych w całej Polsce, a także 13 tys. szkół oraz ośrodków gminy, kultury czy jednostek ochotniczej straży pożarnej. Do dziś w ramach tych działań zapewniliśmy dodatkowo dostęp dla niemal 1 mln gospodarstw domowych.

Bardzo proszę o zadanie drugiego pytania. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wieś z dostępem do Internetu staje się jakby wsią na wyższym poziomie. Chodzi o wyższy poziom dostępu nie tylko do informacji, ale również do ewentualnych inwestycji, do wymiany tych informacji. Oczywiście pan minister mówił, że jest jeszcze sporo tych białych plam, natomiast chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Dotychczasowe łącza, które były na wsi, mają taką małą przepustowość, że trudno je nazwać łączami zapasowymi. Brak tych łączy czasami uniemożliwia czy utrudnia rozwój. I jeszcze, pani marszałek, jedna rzecz.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź na pytanie. Szanowna Pani Marszałek! Państwo Parlamentarzyści! Oczywiście zgadzam się z tym, co pan poseł powiedział. Będziemy jeszcze uważniej przyglądać się tej kwestii, zwłaszcza na wsi, bo zwłaszcza tutaj jest to dla nas niezwykle ważne.

W całej Polsce, zwłaszcza właśnie w gminach, w mniejszych ośrodkach, mają być specjalnie wyedukowani edukatorzy, których zadaniem będzie bezpłatne świadczenie usług w kontekście likwidacji wykluczenia cyfrowego, także nauki np. seniorów, jeśli chodzi o korzystanie z e-usług, z komputera.

Państwowa akademicka sieć komputerowa NASK jest moim zdaniem najlepszym dowodem na to, że rzeczywiście staramy się łączyć kwestię naukową z cyfryzacją i informatyzacją państwa, ale także zgadzam się, że docelowo ten kierunek musi być wzmacniany, zwłaszcza z tych powodów, o których powiedział pan poseł. Bardzo dziękuję.

Pytanie skierowane jest do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Kolekcja wawelska, która powstała dzięki staraniom wielkich mecenasów w 20-leciu międzywojennym, pieczołowicie zbierana w okresie II Rzeczypospolitej, padła ofiarą wojny. Wciąż poszukujemy zgromadzonych w niej dzieł sztuki, które wojenne losy rzuciły w różne miejsca świata. Wiemy, że odnalezienie kolejnego elementu kolekcji to powód do świętowania. Jednak sukces ten nie byłby możliwy, gdyby nie ciężka praca pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którym udało się odnaleźć obraz na aukcji w jednym z domów aukcyjnych. Proszę pana ministra o informację: Jakie działania zostały podjęte, aby odzyskać obraz, oraz jak do roszczeń polskiego państwa odnosił się dotychczasowy właściciel dzieła? Ponieważ jako kraj padliśmy ofiarą zbrojnej napaści oraz rabunku na niespotykaną skalę podczas II wojny światowej, musimy dysponować sprawnymi mechanizmami mającymi na celu restytucję dzieł zrabowanych przez okupantów. Jaki departament ministerstwa prowadzi aktualnie działania restytucyjne? Ile osób w nim pracuje? Czy ministerstwo planuje dalszy rozwój tego departamentu? Chciałbym zapytać również pana ministra, jak wygląda kwestia odzyskanych już dzieł sztuki. Ile z nich udało się odzyskać, w jakim są stanie oraz jakie działania są podejmowane po odzyskaniu poszczególnych dzieł sztuki? Czy ministerstwo dysponuje środkami, aby przeprowadzić na odzyskanych dziełach najlepsze, najpilniejsze prace konserwatorskie? Bardzo bym prosił pana ministra o udzielenie odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panowie Posłowie! Bardzo dziękuję za to pytanie. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście z perspektywy aktywności, którą mam przyjemność realizować w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, właśnie ta aktywność związana z odzyskiwaniem dzieł sztuki zaginionych w czasie II wojny światowej przynosi szczególnie dużo satysfakcji. Pytał pan konkretnie o ostatnio odzyskane dzieło - pastel Leona Wyczółkowskiego pt. „Góralka”, „Wiejska dziewczyna w żółtej chuście” Szczegółowa weryfikacja obiektu i analiza konserwatorska potwierdziły, że oferowany przez jeden z warszawskich domów aukcyjnych obraz jest zarejestrowany w bazie strat wojennych i stanowił do wybuchu II wojny własność Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Dzieło Wyczółkowskiego wpisane było w inwentarzu Fundacji Wawelskiej im. Na prośbę resortu kultury dom aukcyjny wycofał pastel z aukcji, a dotychczasowy posiadacz podjął decyzję o dobrowolnym zwrocie obrazu na rzecz Skarbu Państwa. Pastel powstał w roku 1900, co potwierdza umieszczona w lewym górnym rogu sygnatura artysty oraz data. Wkrótce potem obraz został zakupiony przez Leona Pinińskiego, profesora prawa rzymskiego, rektora uniwersytetu we Lwowie, polityka znanego, bo był namiestnikiem Galicji na przełomie XIX i XX w. Wśród tych obiektów był właśnie obraz Wyczółkowskiego. To tyle, jeśli chodzi o ten konkretny obraz. Co jakiś czas takie uroczystości na szczęście przeżywamy. Teraz trochę informacji ogólnych na temat zasad działania w ministerstwie związanych z odzyskiwaniem dzieł zaginionych w czasie II wojny światowej. Najpierw informacja, że w wyniku II wojny polskie dziedzictwo kulturowe poniosło ogromne straty, szczególnie w zakresie zagrabionych oraz bezpowrotnie zniszczonych dzieł sztuki. Szacuje się, że Polska w tym czasie utraciła ok. 70% materialnego dorobku kulturowego. W związku z tym nie ustajemy w wysiłkach na rzecz poszukiwania i odzyskiwania polskich strat wojennych. Sprawy grabieży dzieł sztuki, co warto podkreślić, nie ulegają przedawnieniu. Możemy, można powiedzieć, bez końca tych dzieł szukać. Dlatego jednym z kluczowych obszarów działalności ministerstwa jest właśnie restytucja. Ministerstwo gromadzi informacje o utraconych dziełach sztuki, które są podstawą prowadzonych poszukiwań i działań restytucyjnych.

Baza stanowi zbiór otwarty. Do chwili obecnej wpisano do niej ponad 64 tys. rekordów i jest ona stale uzupełniana. Jeżeli je znajdziemy, to po prostu od razu mamy taką grubą teczuszkę udowadniającą, że to jest dzieło utracone w czasie II wojny, które powinno być zwrócone. Ministerstwo prowadzi stały monitoring krajowych i zagranicznych rynków dzieł sztuki. Codziennie weryfikowane są kolejne dzieła sztuki, które stanowić mogą obiekty utracone. Systemy informatyczne, którymi dysponuje ministerstwo, pozwalają na codzienną weryfikację kilkuset dzieł sztuki. W celu poszukiwania polskich strat ministerstwo wykorzystuje nowoczesne narzędzia informatyczne, a wszelkie informacje o obiektach, które mogą być tymi utraconymi, są weryfikowane. Obecnie, w tym momencie, resort kultury prowadzi ponad 80 postępowań restytucyjnych w 11 krajach na świecie, m.in. na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Austrii czy też Tadżykistanu. Jedno takie postępowanie restytucyjne to jest dokumentacja ponad 100-stronicowa, żeby w 100% udowodnić, że to jest nasze dzieło. Kluczem do zakończonego sukcesem procesu restytucji jest łączenie różnych metod negocjacyjnych, wykorzystywanie szeregu narzędzi prawnych i pozaprawnych oraz ciągłe poszukiwanie nowych metod odzyskiwania utraconych dóbr kultury, w tym także współpraca z organami ścigania, np. włoskimi carabinieri, amerykańską FBI czy też amerykańską agencją śledczą Homeland Security Investigations. Warto zauważyć, że podczas polsko-niemieckich konsultacji sprzed 3 lat w Warszawie z inicjatywą wspólnego apelu do obywateli niemieckich o zwrot dóbr kultury zagrabionych podczas II wojny wystąpiła ówczesna minister kultury Monika Grütters. Niestety potem się okazało, że jakaś blokada wewnątrz Niemiec nastąpiła i do takiego apelu nie doszło. Ale do tego tematu wrócimy w związku z pojawieniem się nowego rządu koalicyjnego w Niemczech. I jeszcze istotna informacja: w ostatnich 6 latach dzięki pracy ministerstwa do macierzystych kolekcji w polskich muzeach powróciło łącznie 512 obiektów. Restytucja tych obiektów przebiegała w sposób bezkosztowy, w drodze negocjacji bądź procesów sądowych, całkowicie zgodnych z obowiązującym prawem.

Warto też na koniec powiedzieć, że ministerstwo złożyło 20 wniosków restytucyjnych w stosunku do dóbr, które znajdują się na terenie Rosji. Niestety po dziś dzień strona rosyjska nie uwzględniła polskich roszczeń, pozostawiając je bez odpowiedzi. To jest największy problem: relacje z Rosją w tej sprawie. Rosja przyjęła kilkanaście lat temu ustawę o dziełach, które w czasie II wojny światowej w różny sposób zdobyła właściwie jako łup wojenny (Dzwonek), i nie jest otwarta na rozmowy o zwrocie dóbr kultury. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie zadaje pan poseł Jerzy Paul. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Czy może pan, panie ministrze, przekazać informację, jakie zaginione czy zrabowane dzieła mają dla ministerstwa najwyższą wartość oraz kto odpowiada za opracowanie listy zrabowanych dzieł? Chciałbym jeszcze, panie ministrze, dowiedzieć się, czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego współpracuje w tych sprawach z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jeżeli chodzi o odzyskanie tych dzieł? Dziękuję. Bardzo proszę jeszcze raz pana ministra Jarosława Sellina o odpowiedź na pytanie. Szanowny Panie Pośle! Hierarchia jest oczywista. Najwyżej w hierarchii poszukiwanych dzieł sztuki jest obraz Rafaela „Portret młodzieńca” Jeżelibyśmy ten obraz znaleźli, to. Jest on oczywiście na samym szczycie dzieł, które poszukujemy, bo to jest obraz tej rangi, tej wartości co „Sąd ostateczny” Memlinga w Gdańsku czy też „Dama z łasiczką” Leonarda da Vinci w Krakowie. Wśród tych 64 tys. dzieł są dzieła wielkie, są też dzieła może nie tak cenne, ale wszystkich poszukujemy, bo uważamy, że powinny wrócić do właściwych miejsc. W tym momencie może wykorzystam tę sytuację i powiem o dziełach najcenniejszych, które w ostatnich latach odzyskaliśmy, np. obraz Maksymiliana Gierymskiego „Zima w małym miasteczku”, który wrócił do Muzeum Narodowego w Krakowie, obraz Teodora Axentowicza „Dama w pawich piórach”, który wrócił do Muzeum Narodowego w Warszawie, obraz Michała Gorstkina-Wywiórskiego „Chata w śniegu”, bardzo cenna rzecz pochodząca ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, obraz Abrahama Bloemaerta „Apollo i Dafne”, który wrócił do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, czy też kolekcja 124 obiektów etnograficznych z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Wykorzystam też tę drugą część pytania do poinformowania, jak ta praca w ministerstwie jest zorganizowana. On się tak nazywa. W tym departamencie pracuje ponad 30 osób. Można powiedzieć, że to jest nasz wydział detektywistyczny, który właśnie tropi ślady dzieł, które są gdzieś w świecie, a pochodzą z polskich zbiorów. Ale postanowiliśmy od Nowego Roku, od 1 stycznia przyszłego roku tę sytuację jeszcze bardziej wzmocnić.

Uważam, że mamy ich dużo w ostatnich 6 latach - o tych liczbach mówiłem - ale oczywiście chcemy, żeby tych sukcesów było jeszcze więcej. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Przystępujemy do następnego pytania.

Pytanie jest skierowane do ministra klimatu i środowiska. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze!

Jak wynika z informacji medialnych i informacji wpływających do naszych biur poselskich, Lasy Państwowe prowadzą zorganizowaną akcję działania przeciw lokalnym działaczom społecznym występującym głównie przeciw wycince lasów, zwłaszcza ochronnych.

W związku z tym, że takie działania mogą mieć efekt mrożący i rażąco naruszają te konstytucyjne prawa, które przywołałam, chciałam zapytać: Ile takich spraw w stosunku działaczy organizacji prowadzą poszczególne nadleśnictwa? Jakich kwot żądają od organizacji pozarządowych?

Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pana Edwarda Siarkę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Na wstępie chciałbym zdecydowanie i jednoznacznie powiedzieć, że pytanie, które pani poseł zadała w imieniu kilku posłów na samym początku, zawiera w swej treści nieprawdziwą tezę.

Nieprawdziwa jest teza, którą pani tutaj wygłosiła.

One są czymś naturalnym.

A często tak się zdarza. Chcę powiedzieć, że lasy prowadzą swoją działalność na zasadzie samofinansowania. Pokrywają wszystkie koszty z własnych przychodów.

Nie wyobrażam sobie, żebyśmy takiej obsługi prawnej nie mieli. Dlatego zupełnie nie rozumiem pani zarzutu.

Lasy Państwowe to przede wszystkim 429 nadleśnictw, 17 dyrekcji regionalnych, 26 tys. ludzi.

To wszystko wymaga oprzyrządowania prawnego. Środki, które Lasy wygospodarują, temu wszystkiemu służą. Przypomnę, że cały sektor leśny generuje 500 tys. miejsc pracy w Polsce, więc mówimy o bardzo dużym obszarze działalności.

Bardzo proszę, pani poseł Agnieszka Pomaska, Koalicja Obywatelska, drugie pytanie. Panie i Panowie Posłowie!

Po drugie, proszę się nie dziwić naszemu zaniepokojeniu, dlatego że niejednokrotnie media donosiły o tym, że Lasy Państwowe, niekoniecznie w sposób oficjalny, walczą z organizacjami pozarządowymi, które mają na celu ochronę środowiska.

I związku z tym moje pytanie do pana ministra: Jak pan minister ocenia współpracę Lasów Państwowych, ale też przedstawicieli rządu, z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się kwestiami ochrony środowiska? Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź na pytanie. Pani Poseł! Przede wszystkim na samym początku tej części mojej wypowiedzi chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, że lasy w pojęciu gospodarczym, Lasy Państwowe nie prowadzą, proszę państwa, wycinki.

Chcę powiedzieć, że bardzo dużą wagę przywiązujemy do działań edukacyjnych. Proszę państwa, Lasy Państwowe, jeśli chodzi o funkcję społeczną, na dzień dzisiejszy prowadzą na swoim terenie ok. 6 tys. różnego rodzaju obiektów edukacyjnych.

I na bieżąco te organizacje ekologiczne są dopuszczane czy też biorą udział w uzgadnianiu takich dokumentów jak chociażby plany urządzenia lasu. Tak że nie odbieram tego, co panie mówią, jako braku woli do współpracy, wręcz przeciwnie, lasy są otwarte na taką współpracę i argumenty, które padają ze strony różnych środowisk, na dobrą sprawę w tej działalności są uwzględnione. Dziękuję bardzo. Pytanie zadają posłowie Marek Polak, Grzegorz Lorek, Krzysztof Czarnecki i Kazimierz Gwiazdowski, Prawo i Sprawiedliwość, w sprawie zwiększenia kar za nielegalny import do Polski odpadów niebezpiecznych - do ministra klimatu i środowiska. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Od lat rokrocznie z wielu krajów świata, zwłaszcza z państw członkowskich Unii Europejskiej, do Polski przywożonych jest kilkaset tysięcy ton odpadów, a najwięcej od naszego zachodniego sąsiada, czyli z Niemiec. A powodem takiego stanu rzeczy, jak można się domyślać, jest różnica kosztów przetwarzania odpadów wynikająca m.in. z niższych kosztów pracy, a także opłat i obostrzeń prawnych obowiązujących na terytorium danego państwa. Tak czy inaczej szansę na zysk ma zarówno podmiot przywożący odpady do Polski, jak i przedsiębiorca je przyjmujący. Problem pojawia się dopiero wówczas, gdy polski odbiorca ogranicza się tylko do zdeponowania często toksycznych i niebezpiecznych odpadów bez zamiaru ich przetwarzania i porzuca zgromadzony materiał, który stanowi wówczas nielegalne wysypisko odpadów. Dlatego chciałbym zapytać pana ministra, jaka jest skala powstawania nielegalnych wysypisk odpadów niebezpiecznych, czyli ile w ciągu roku ujawnia się tego rodzaju przestępstw, i jakie są podejmowane działania w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na pytanie odpowie sekretarz stanu w ministerstwie. A, przepraszam, bardzo przepraszam, pytanie było podzielone. Bardzo przepraszam, panie pośle. Dziękuję, pani marszałek. Panie Ministrze!

Osoby, które przyczyniły się do powstania tego składowiska, oczywiście zostały zatrzymane, natomiast problemem jest to, kto ma to teraz posprzątać. Dziękuję. Dziękuję bardzo i przepraszam, panie pośle. Bardzo proszę, pan minister odpowiada na pytanie. Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo!

Ja wolę tę szczerą prawdę niż tuszowanie rzeczywistości. Koszty unieszkodliwienia są gigantyczne, bo ceny unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zdecydowanie wzrosły.

Musimy pamiętać o tym, że na podstawie art. 26a ustawy o odpadach istnieje możliwość dofinansowania unieszkodliwienia takich odpadów dla samorządów, które nie mają odpowiednich środków. Pragnę tutaj przypomnieć, że przez 10 lat przestępcy środowiskowi wpłacili na rzecz narodowego funduszu ochrony środowiska z tytułu orzekanych nawiązek po popełnionym czynie zabronionym z artykułów, które znajdują się w Kodeksie karnym w rozdziale XXII dotyczącym przestępstw środowiskowych, 1 mln zł. Czyli przestępcy, którzy zarabiali gigantyczne kwoty, na rzecz narodowego funduszu wpłacili 1 mln zł. Padło pytanie, co robimy. Podwyższamy dolną i górną granicę właściwie we wszystkich przestępstwach środowiskowych. W zakresie odpadów, które są importowane, w art. 183 podnosimy dolną i górną granicę.

Po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej będzie obowiązek posiadania systemu SENT i kara za nieposiadanie tego systemu.

To daje możliwość zwiększenia wykrywalności.

Karniści mogą się złapać za głowy, ale pamiętajmy, że skala jest bardzo duża.

Ja bym miał prośbę, żeby pani nie rozmawiała przez telefon, bo to trochę dekoncentruje. Poza tym działania związane z Inspekcją Ochrony Środowiska, koordynacja działań z Krajową Administracją Skarbową, Inspekcją Transportu Drogowego. Skoordynowanie powoduje, że ta wykrywalność jest zdecydowanie zwiększona, i daje możliwość, również w zakresie kar, tzw. efektu mrożącego, którego się spodziewamy, bo dzisiaj niestety z przykrością stwierdzam, że odpowiedzialność, a właściwie decyzje sądowe, wyroki są zdecydowanie za niskie.

Ale mogę powiedzieć, że kwoty są bardzo duże. Na przykład Gorlice, koszt unieszkodliwienia to ponad 90 mln, Mysłowice itd., ale to już we współpracy z narodowym funduszem ochrony środowiska, o którym wspominałem, bo tutaj chcemy przekazać źródło finansowania w ramach środków pozyskanych od przestępców.

Chciałam państwa na sali poprosić o ciszę, bo jeszcze mamy parę pytań do zadania i chcielibyśmy to zrobić dobrze. Bardzo proszę pana posła Marka Polaka o zadanie dodatkowego pytania. Dziękuję bardzo. To bardzo dobrze, że rząd dostrzega problem nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych i podejmuje skuteczne działania ograniczające ten proceder, m.in. poprzez podwyższenie kar za tego rodzaju działalność przestępczą, ale w świetle obowiązujących przepisów w przypadku uchylania się właściciela odpadów od likwidacji nielegalnego składowiska obowiązek ten spoczywa wyłącznie na budżetach gmin, a koszty jego realizacji mogą wynosić kilka tysięcy, a nawet miliony złotych. Proszę powiedzieć, co robić, jeśli koszty likwidacji nielegalnego składowiska odpadów przekraczają możliwości finansowe gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę.

Gdy tego nie ma i samorząd nie ma własnych środków, to jest właśnie art. 26a ustawy o odpadach, czyli fundusz, z którego narodowy fundusz ochrony środowiska przeznacza co roku środki finansowe na dofinansowanie tego unieszkodliwienia. My w ramach nowelizacji Kodeksu karnego, tak jak wspominałem, chcemy zwiększenia tego funduszu i odciążenia strony samorządowej na zasadzie koszty plus.

A więc jedyna możliwość to jest znalezienie środków finansowych na dofinansowanie dla strony samorządowej po to, aby te koszty były zdecydowanie mniejsze. Czyli z jednej strony efekt mrożący, zwiększona wykrywalność, a z drugiej to, co zalega, będzie sprzątnięte w dłuższej perspektywie, bo koszty są gigantyczne, za sprawą tych środków, co do których chcemy, aby były wpłacane na rzecz narodowego funduszu ochrony środowiska.

Wiemy, że w kilku przypadkach byłoby to możliwe do zapłacenia przez przestępców, a takie środki mogłyby pozwolić na to, żebyśmy w dłuższej perspektywie przedstawili mapę drogową: wpływy kontra dofinansowanie dla strony samorządowej. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do ostatniego pytania. Pytanie zadają posłowie Waldemar Andzel, Elżbieta Płonka, Jarosław Krajewski i Ryszard Terlecki, Prawo i Sprawiedliwość, w sprawie programu „Rozwój lokalny” - do ministra funduszy i polityki regionalnej. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Polska otrzymała ponad 102 mln zł z funduszy norweskich na rozwój małych i średnich miast. Program „Rozwój lokalny” obejmuje 29 miast. Proszę o wskazanie innych źródeł finansowania tego programu. Na jakie inwestycje zostaną przeznaczone te środki? Jakie są szczegóły tego programu?

Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Nigdy dotychczas nie było takich możliwości w zakresie inwestycji lokalnych jak obecnie. Od roku mamy tę szansę. Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Gminy wiejskie, o które chcę spytać, skorzystają na Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład, dzięki któremu będą mogły prowadzić inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne i gazyfikacyjne. Dziękuję bardzo. I proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pana ministra Waldemara Budę. Wysoka Izbo! Pytanie w zasadzie sprowadza się do dwóch wątków. Rozpoczynając od tego pierwszego poruszonego przez pana posła Waldemara Andzela, przede wszystkim chciałbym wskazać, że program „Rozwój lokalny” to program, który jest finansowany ze środków norweskich oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To jest program innowacyjny, ponieważ po raz pierwszy został zaprojektowany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i samo ministerstwo było instytucją zarządzającą i wdrażającą ten program. Rzeczywiście on się spotkał z bardzo dużym zainteresowaniem, bo na 240 bodajże miast, które były uprawnione do startowania w konkursie o te środki, wystartowało 213 bodajże, a ostatecznie 29 otrzymało pomoc. 54 przeszły do kolejnego etapu, drugiego, a ostatecznie 29 otrzymało pomoc. Dlaczego te środki były tak atrakcyjne i dlaczego ten program był tak ważny? Ano dlatego że, po pierwsze, te inwestycje były finansowane w 100%, czyli nie było wkładu własnego samorządu. Po drugie, wartość tych zadań, które były realizowane, była stosunkowo wysoka, bo 3,5 mln euro na każde z miast.

Czyli to takie strategiczne, horyzontalne podejście do inwestycji lokalnych, taka praca u podstaw, która dała samorządom szansę zbudowania pewnej strategii na przyszłość, na wiele lat.

Przechodzę natomiast do dużego, niewspółmiernie dużego budżetu i programu Polski Ład. Wszyscy wiemy, że to jest program obliczony nawet na ponad 100 mld zł. Jeszcze w grudniu będzie ogłoszony kolejny nabór, też na ok. 20 mld, to będzie już drugi nabór w tym roku.

Na co te środki mają być przeznaczone? Jest 36 zadań, pakietów zadań w ramach czterech priorytetów. Bardzo szeroko zostało to ujęte, tak żeby to samorządowcy decydowali o tym, jakie inwestycje mają być realizowane. Wyjątki stanowią tylko inwestycje z zakresu służby zdrowia, ponieważ tutaj potrzebna jest koordynacja i na to jest osobny fundusz. Natomiast wszystkie inne w zasadzie inwestycje mogły być realizowane z tego funduszu. Pierwsze rozstrzygnięcie, jak państwo wszyscy wiedzą, było bardzo przejrzyste, bardzo transparentne.

Chodzi chociażby o sytuację, w której gmina kilkutysięczna wnioskowała o kilkadziesiąt milionów. Nawet z budżetu wynikało, że nie była w stanie zapewnić wkładu własnego w tym programie, więc oczywiste było, że raczej nie mogła spodziewać się, że te środki otrzyma. W każdym razie w najbliższym czasie, czyli w grudniu, ale też w kolejnym roku 2022, będą co najmniej jeszcze dwa nabory porównywalnej wielkości, więc można się spodziewać, że Polska lokalna w najbliższym czasie będzie wielkim placem budowy. Zachęcam wszystkie samorządy do uczestniczenia w tym konkursie. Rozstrzygnięcie będzie prawdopodobnie - prawdopodobnie, tutaj zastrzegam - do końca lutego, niemniej jeszcze w 2022 r. będą dwa kolejne nabory, myślę, że podobnej wielkości jak ten pierwszy i ten planowany drugi. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Za chwilę ten punkt kończymy. a dokładnie Zagłębia Dąbrowskiego, mam pytanie: Jakie miasta z województwa śląskiego zostaną objęte programem „Rozwój lokalny” Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem pytanie. Rozumiem, że chodzi o listę beneficjentów z regionu śląskiego w ramach „Rozwoju lokalnego” Już wskazuję.

Nie sposób ich wskazać, ale najczęściej to była modernizacja transportu miejskiego, najczęściej były to obiekty kultury, najczęściej były to obiekty użyteczności publicznej. W szczegółach te projekty bardzo się różniły, ale miały jedną cechę wspólną: były bardzo komplementarne, czyli przewidywały inwestycje w wielu sektorach, ale mających cechy skoordynowane, uspójnione, tak żeby stanowiły pewną wartość dodaną po zrealizowaniu tych inwestycji. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Pytanie to kończy rozpatrywanie tego punktu. Ogłaszam przerwę do godz. 11.30.

Wysoka Izbo! Bardzo proszę o powstanie. Wysoka Izbo!

Dziękuję bardzo. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, druk nr 1848. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu, oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął. W związku ze zgłoszonym sprzeciwem sprawę tę rozstrzygniemy w głosowaniu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za wyrażeniem zgody na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu, oraz na wysłuchanie 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół w przypadku poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. U kogo nie działa?

Działa, tak? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm propozycje przyjął.

Wysoka Izbo! Mój wniosek jest dość specyficzny i nietypowy. Mianowicie chciałbym prosić panią marszałek w imieniu chyba nas wszystkich, prawie wszystkich, o wykluczenie z obrad Sejmu piątki posłów Konfederacji, [[Oklaski]] którzy wczoraj przynieśli hańbę tej Izbie, hańbę Polsce, hańbę ofiarom i potomkom ofiar Holocaustu, o wykluczenie ludzi, którzy po prostu zapomnieli, czym jest przyzwoitość, [[Oklaski]] czym jest moralność, czym jest historyczna wierność pamięci, czym jest tak naprawdę służba w Rzeczypospolitej z tego miejsca, z Sejmu, z Senatu, w imieniu narodu.

Natomiast bardzo proszę pana posła Brauna, pana posła Kuleszę i pana posła Bosaka o założenie maseczek. Bardzo proszę panów o założenie maseczek. Proszę pana posła Brauna i pana posła Kuleszę o założenie maseczek. Pan poseł Braun, pan poseł Kulesza. Panowie posłowie, zwracam się. Panie pośle Braun, zwracam uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Bardzo pana proszę o założenie maseczki. Panie pośle, na podstawie art. 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku. i po raz kolejny proszę o założenie maseczki.

Panie pośle, pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad. Na podstawie art. 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę plenarną.

Proszę.

Wiem, że po prawej stronie są też lekarze. Kodeks etyki lekarskiej mówi, że najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego. Co wy w tym czasie robicie? Dlaczego nie wprowadzacie obowiązku szczepień? Dlaczego nie wprowadzacie paszportów sanitarnych? Ludzie umierają, nasi bliscy umierają. Ile jeszcze grobów mamy wykopać, zanim w końcu weźmiecie się do roboty, zanim pozwolicie na to, żebyśmy mogli poczuć się bezpiecznie? My się nie boimy. Pomożemy wam. To jest wasza wina, że ci ludzie umierają.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja z wnioskiem przeciwnym. Proszę państwa, wczoraj umarło 1300 osób na inne choroby. Dlaczego? To też jest wina rządu? Obowiązkiem lekarza jest leczyć, a nie przymusowo leczyć. Proszę państwa, państwo stukający w te pulpity, chcecie, żeby przy waszych wypowiedziach był spokój, ale jak ktoś inny się wypowiada, to tak reagujecie? A gdzie tu demokracja, gdzie tu wolność wypowiedzi? Szanujmy się nawzajem. Proszę bardzo, pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Panie Premierze! Wysoka Izbo! Instytut Pamięci Narodowej szacuje, że w wyniku stanu wojennego zginęło ok. 100 osób. Każda z tych śmierci była tragiczna, każda z tych śmierci była niepotrzebna. Panie pośle, demagogiczne wypowiedzi to nie jest wniosek formalny. Bardzo proszę, pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja, z wnioskiem formalnym. Wysoka Izbo! Prawda jest taka.

Panie Pośle Grupiński! Chciałem panu powiedzieć, że gdyby wykluczano za udział w manifestacjach, w których pojawiły się kontrowersyjne rzeczy, to panie pośle, cały wasz klub, cały klub Lewicy po zeszłym roku musiałby być wykluczony na zawsze z tych obrad. Po 2020 r. was nie powinno być w polskim życiu publicznym.

Szanowni Państwo! Lewica się podzieliła, ale w tej Izbie będzie wiadomo, kto jest na prawicy, kto jest na lewicy.

Proszę nie uskuteczniać takich zachowań, bo to jest niepoważne i niegodne polskiego Sejmu. Panie pośle, radzę ostudzić emocje. Proszę państwa. Nie, trzeba patrzeć, panie przewodniczący, na to, kto zaczął, a nie na to, kto kończy, naprawdę. Powracamy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1821. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1821, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy byli za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Powracamy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1837. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1837, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Powracamy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1836-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Piotra Króla o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1835. Sejm na 44. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2021 r. zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1836 do Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2021 r. wnosi, by Wysoki Sejm sześć poprawek odrzucił, a niniejszy projekt ustawy był łaskaw przyjąć. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz poprawki. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych propozycji. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Z poprawką tą łączy się poprawka 2. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 4. poprawce wnioskodawcy proponują zmiany w załącznikach nr 1, 3 i 4. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Poprawki 5. i 6. zostały zgłoszone do art. 2 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o czasie pracy kierowców. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 6., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1836, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm, zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 1692, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia. Przypominam, że kluby złożyły wnioski o uzupełnienie porządku dziennego: - Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy - o punkt: Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych w sprawie stanu negocjacji z Republiką Czeską dotyczących dalszego funkcjonowania Kopalni Węgla Brunatnego Turów, - Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni - o punkt: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań podjętych przez Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci osób w trakcie interwencji dolnośląskich policjantów oraz działań dyscyplinarnych podjętych wobec funkcjonariuszy przeprowadzających przedmiotowe interwencje. W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam kolejno pod głosowanie wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o te punkty. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowania te nie są poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji w sprawie stanu negocjacji z Republiką Czeską dotyczących dalszego funkcjonowania Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek o uzupełnienie porządku dziennego odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań podjętych przez Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci osób w trakcie interwencji dolnośląskich policjantów. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek o uzupełnienie porządku dziennego odrzucił. Ogłaszam 5 minut przerwy.

Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Informacja bieżąca. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie kierunków i strategii polskiej polityki względem Unii Europejskiej, wybranych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych, o której przedstawienie wnosi Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców pana przewodniczącego Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Na początku pytanie techniczne, kto reprezentuje rząd, bo był to wniosek do pana premiera. Sejm jest organem kontrolującym, nadzorującym działanie Rady Ministrów, więc ma prawo żądać odpowiedzi, ma prawo pytać, ma prawo kontrolować, przede wszystkim ma prawo wiedzieć. Dzisiaj proponujemy debatę o polityce międzynarodowej, o strategii Polski wobec naszych sąsiadów, o naszej roli w Unii Europejskiej, o relacjach Polska - Unia Europejska, wewnętrznych, z sąsiadami i ze Stanami Zjednoczonymi, z naszymi sojusznikami. Po pierwsze, dobrym zwyczajem w państwach demokratycznych jest utrzymywanie wektorów polityki międzynarodowej niezależnie od tego, jaki jest rząd. Ten zwyczaj w młodej polskiej demokracji najlepiej funkcjonował na jej początku, czyli w latach 90., kiedy zgłaszaliśmy swoją akcesję do Unii Europejskiej, przystępowaliśmy do NATO. W ostatnich latach to w ogóle nie funkcjonuje, nie ma prawdziwych, realnych dyskusji, konsultacji i uzgadniania wspólnego stanowiska w sprawach międzynarodowych.

Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie marszałku, proszę się nie dziwić, że części ministrów nie interesuje polityka zagraniczna, bo oddali ją w ręce ministra sprawiedliwości, ministra Ziobry. Nie jest to dla mnie zaskoczeniem.

Nie chcieliście wykonać wysiłku i nie chcieliście takiej uwspólnotowionej koncentracji działań w polityce międzynarodowej. Szkoda, bo to jest zawsze strata dla państwa, jeżeli nie występuje jeden głos na arenie międzynarodowej. Wspólny głos w sprawach najważniejszych powinien być wspólnym głosem rządzących i opozycji, bo to jest sprawa kluczowa i dla racji stanu, i dla przyszłych pokoleń, nie tylko dla tych, którzy dzisiaj rządzą.

Z jednej strony mówicie, że nowy rząd niemiecki to nowe otwarcie w polityce, jedna z pierwszych wizyt nowego kanclerza odbyła się w Warszawie, a z drugiej strony jest informacja medialna i taki przekaz, że Niemcy proponują IV Rzeszę. Ani ładu, ani składu to nie ma.

Minęło ponad pół roku, 18 państw w Unii Europejskiej ma wypłacone zaliczki, niektórzy już będą, jak np. Hiszpanie, sięgać po środki z samego funduszu, już nie te zaliczkowe. My mieliśmy dostać 20 mld zaliczki, nic z tego do Polski nie dotarło.

Kolejna kwestia to kary, które ponosimy w związku z nieudolnością waszej polityki międzynarodowej i nieskutecznością, wymachiwaniem szabelką i skłócaniem nas z Unią Europejską.

I znów ta schizofrenia w polityce międzynarodowej się pojawia, że nie chcecie. Prezes, premier Morawiecki mówią: tak, zlikwidujemy zaraz Izbę Dyscyplinarną. Tylko żadnej ustawy w tej sprawie nie ma. Później jest wywiad. I tu pytanie do ministra spraw zagranicznych: Czy ten wywiad pana ministra Ziobry w „Financial Times” był autoryzowany? A powiedzenie, jak słyszymy od rzecznika, że to była prywatna wypowiedź ministra sprawiedliwości, jest kompletnie kuriozalne. Minister nie wypowiada się prywatnie, udzielając wywiadu w jednym z najważniejszych dzienników na świecie. On reprezentuje wtedy rząd. Stąd teza postawiona przed chwilą, że premier Morawiecki abdykował z roli kreatora polityki międzynarodowej, do czego przypisuje go konstytucja, a minister do spraw zagranicznych i do spraw europejskich w ogóle nie istnieje dzisiaj w waszym rządzie, bo to stanowisko jest wypełniane, ale nie jest w żaden sposób piastowane i nie kreuje żadnej polityki międzynarodowej. Z jakimi wskazówkami i z czyimi wskazówkami, z czyimi rekomendacjami pojedzie na szczyt europejski pan premier Morawiecki? Ze swoimi czy z deklaracjami realnego ministra spraw zagranicznych, czyli pana posła Kowalskiego? Bo on w tej sprawie się wypowiada najczęściej, w sprawie relacji Polska - Unia Europejska. Oczekujemy kilku spraw, które natychmiast trzeba załatwić. Po pierwsze, domagamy się, aby ani rząd nie przedstawiał, ani posłowie większości rządzącej nie prezentowali i nie zgłaszali żadnych ustaw, które mogą nas skłócić z Unią Europejską i ze Stanami Zjednoczonymi. To jest po prostu działanie wbrew interesowi bezpieczeństwa państwa polskiego. W tak trudnej sytuacji geopolitycznej, w tak trudnej sytuacji na Ukrainie posiadanie sojuszników i gwarancji bezpieczeństwa Unii Europejskiej i NATO jest podstawą bezpieczeństwa państwa polskiego. Jeżeli będziecie tej zasadzie przeczyć, jeżeli tę zasadę będziecie niszczyć kolejnymi wrzutkami dotyczącymi zerwania relacji gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi czy ciągłego nierespektowania zasad, na które się umówiliśmy w Unii Europejskiej, będziecie winni narażenia Polski na niebezpieczeństwo. Będziecie winni narażenia i zdrady racji stanu. Kolejny punkt to jest współpraca z opozycją w sprawie bezpieczeństwa na granicy wschodniej Unii Europejskiej, na granicy wschodniej Rzeczypospolitej. Oczekujemy tej współpracy i my jako klub parlamentarny mamy ogromne prawo tej współpracy żądać, ponieważ zagłosowaliśmy za zaporą jako jedyny klub opozycyjny. Myślę, że zrobiliśmy dobrze: widzę też działania Unii Europejskiej, która chce na to przekazać środki.

Domagamy się współdziałania w sprawie bezpieczeństwa na wschodniej granicy. Dostaliście mandat do rządzenia, ale nie zjedliście wszystkich rozumów, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy polityki międzynarodowej. Kolejna sprawa. Wykonanie postanowień trybunałów europejskich, żebyśmy nie byli stratni - szczególnie mówię tutaj o Izbie Dyscyplinarnej - jeżeli chodzi o otrzymanie funduszy na rzecz polskich przedsiębiorców, rolników, wspólnot samorządowych. Trzeba wykonać te postanowienia i sięgnąć natychmiast po pieniądze, bo te pieniądze są potrzebne na walkę z pandemią. Dojście do porozumienia z Republiką Czeską, bardzo ważne. Nie stawianie pod ścianą, tylko życzliwa, normalna rozmowa i wniosek do Republiki Czeskiej, żeby się dogadać i żeby oni wycofali swoje wnioski do Trybunału Europejskiego. To jest załatwianie sprawy w Grupie Wyszehradzkiej, tak jak powinno być między dobrymi sąsiadami. A wy nawet z dobrymi sąsiadami, z tymi państwami, na które stawialiście od początku przejęcia rządów, nie potraficie prowadzić dialogu. Wznowienie rozmów w ramach Trójkąta Weimarskiego. To jest niezwykle ważne i do tego wzywa pan prezydent Macron. Potwierdził mi to pan premier w rozmowie, którą odbyliśmy jako wszystkie kluby opozycyjne w sprawie sytuacji na Ukrainie. Przychyla się do tego kanclerz Niemiec. To jest grupa, w której Polska powinna odbywać ważną rolę, a Trójkąt Weimarski powinien odgrywać ważną rolę w Unii Europejskiej. Zaprzestanie skłócania nas z sąsiadami, którzy są członkami Unii Europejskiej. Mowa o Niemczech, bo wypowiedzi dotyczące IV Rzeszy są po prostu kompletnie niepotrzebne i nieprzystające do rzeczywistości. Dzisiaj mamy największą wymianę gospodarczą z Niemcami, mamy dobre relacje od czasu porozumienia, które zawierał rząd Tadeusza Mazowieckiego. Skłócanie nas dzisiaj z jednym z najważniejszych państw na świecie i jednym z najważniejszych państw Unii Europejskiej jest po prostu kardynalnym błędem, jest błędem w podstawach funkcjonowania polityki zagranicznej. To są nasze rady dla polskiego rządu. Nie oburzajcie się, koledzy z opozycji, że oni próbują nas obrażać.

To są nasze wezwania do rządu, to są nasze propozycje racjonalnej polityki międzynarodowej. To jest realna polityka międzynarodowa, która jest dbaniem o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej poprzez obecność w silnych sojuszach, w silnej Unii Europejskiej. w rodzinie zjednoczonych narodów, w której Polska jest państwem stanowiącym, [[Oklaski]] a nie na marginesie, nie jest czarną owcą, tak jak wy ją sprowadziliście.

Dziękuję bardzo. Zwracam się do pana posła Tułajewa, aby nie propagował niemieckich zawołań na sali sejmowej, bo jesteśmy w polskim parlamencie.

Prosiłem pana, aby pan w polskim parlamencie nie wzywał i nie używał niemieckich zawołań, a pan tego użył i nie będzie żadnego sprostowania. Jeszcze raz pana proszę, aby pan w polskim parlamencie nie używał zawołań niemieckich. W takim razie jeżeli to nie pan, to bardzo pana przepraszam.

Bardzo proszę, panie ministrze. Panie i Panowie Posłowie! Chciałbym przedstawić informację po wystąpieniu pana przewodniczącego, pana prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza. Obiecuję państwu, że to będzie wystąpienie merytoryczne, niepolityczne, bez kwiecistych sformułowań, retorycznych, a będzie dotyczyło wyłącznie faktów z polityki zagranicznej. Od 2015 r., czyli od kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości steruje polityką zagraniczną, priorytety polityki zagranicznej są niezmienne. To silna, bezpieczna, suwerenna Rzeczpospolita, odgrywająca ważną rolę w wymiarze regionalnym, europejskim, a w określonych aspektach - również w wymiarze globalnym. Pamiętajcie państwo, że Polska jest krajem średniej wielkości w Europie, ale należy też do tych krajów, które od 2015 r. nadają ton działalności w ramach Unii Europejskiej.

My po prostu ten główny nurt polityki unijnej formułujemy.

Było tyle śmiechów, było tyle drwin z tego, że to jest niemożliwe. Okazuje się, i pokazują to szczególnie ostatnie tygodnie, że cała Unia Europejska przyjęła polski punkt widzenia przedstawiany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości od 2015 r. Drugi przykład: nam chodzi nie o to, żeby nas poklepywano po plecach i mówiono: dobrze, dobrze. tylko o to, żeby realnie walczyć o polskie interesy. żeby realnie wpływać na to, co się dzieje w Unii Europejskiej. Przypominam, że to my staliśmy się, a dokładnie pan premier Mateusz Morawiecki stał się kreatorem nowej struktury organów unijnych, nowej struktury personalnej w ramach Unii Europejskiej.

Gdyby nie skuteczność naszej dyplomacji, nie byłoby ograniczenia napływu imigrantów z krajów, z których oni pochodzą. Gdyby nie skuteczność polskiej dyplomacji i działań pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana prezydenta Andrzeja Dudy, nie byłoby szeregu wypowiedzi i działań podejmowanych przez przywódców krajów zachodnioeuropejskich, potwierdzających nasz punkt widzenia na kryzys. Nie byłoby wreszcie kolejnych pakietów sankcji nakładanych z inicjatywy Polski przez Unię Europejską na Ukrainą, na reżim.

Ogromną wagę przywiązujemy również do wymiaru regionalnego.

Znowu przywołam ostatni kryzys migracyjny, ten kryzys migracyjny na granicy z Białorusią, dlatego że Polska stała się głosem regionu w tej sprawie, nie tylko w relacjach wewnątrzunijnych, ale też w relacjach atlantyckich. I wreszcie trzeci aspekt: relacje atlantyckie.

Deklaracja o obronie wartości i budowaniu dobrobytu poprzez polsko-amerykańskie partnerstwo strategiczne, jak również deklaracja o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej oraz wspólna deklaracja na temat pogłębienia współpracy obronnej - to są te elementy, dzięki którym mamy niespotykaną w historii obecność amerykańską na terytorium Rzeczypospolitej, co teraz ma szczególne znaczenie w kontekście imperialnej polityki Rosji, imperialnej polityki Białorusi, konfrontacyjnej polityki Białorusi wobec Polski, ale także wobec Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego. To właśnie dzięki tym dobrym relacjom ze Stanami Zjednoczonymi jesteśmy w stanie wpływać również na rozmowy, które się toczą w relacjach amerykańskich z partnerami ze Wschodu, nie tylko amerykańskich, ale również europejskich.

Dziękuję bardzo panu ministrowi. Proszę teraz o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pana ministra Waldemara Budę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wszyscy państwo znają stan negocjacji, nie chciałbym go powtarzać.

Wyraziliśmy zgodę na prośbę Komisji o jednomiesięczne wydłużenie tego terminu i w związku z tym ten termin upłynął 3 sierpnia. Teraz, szanowni państwo, jest sytuacja, w której w sposób wprost jawny mamy do czynienia z konfliktem działań Komisji w stosunku do tego, co jest zapisane w rozporządzeniu. Jak sądzę, to będzie spory problem, nie tylko dla nas, ale myślę, że szczególnie dla Komisji, która musi jakoś tę sytuację wytłumaczyć, a nie ma wytłumaczenia tej sytuacji.

Jeżeli z tego miejsca mógłbym do państwa zaapelować o to, ażeby nie inicjować, nie podpisywać. nie robić inicjatyw, które idą w poprzek interesowi polskiemu, chociażby w Parlamencie Europejskim, to byłbym bardzo państwu za to wdzięczny.

Naprawdę wygląda to słabo, w większości państwa koledzy albo byli inicjatorami rezolucji, albo podpisywali się pod rezolucjami, które wprost utrudniały nam dyskusję na temat zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy. Takie są niestety fakty. Nie trzeba daleko szukać, w tym parlamencie największa partia opozycyjna była przeciwko ratyfikacji decyzji Rady o zasobach własnych, która była podstawą do złożenia Krajowego Planu Odbudowy.

Natomiast te działania na arenie międzynarodowej za każdym razem utrudniają nam porozumienie.

Ale kolejność jest jasna: zatwierdzenie negocjacji i KPO i dopiero reforma wymiaru sprawiedliwości. Dziękuję bardzo panu ministrowi.

Jeżeli ktoś będzie mówił dłużej, to oczywiście uszanujemy to. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Była mowa o suwerenności. Polacy, kiedy w 1989 r. odzyskiwali niepodległość, tę zasadę suwerenności przyjęli, na nią się umówili, bo jest to istota, podstawa demokracji, doceniona przez wszystkich, ujęta w wielu dokumentach międzynarodowych. Przytoczę jeden - Karta Narodów Zjednoczonych, mówiąc o suwerenności, określając zasady postępowania członków i samej organizacji, na pierwszym miejscu wskazała suwerenną równość, zobowiązującą członków do powstrzymania się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa bądź w jakikolwiek inny sposób. Czyli tak: suwerenność (Dzwonek) oznacza, że państwa są równe wobec prawa. Każdemu państwu przysługują prawa wynikające z pełnej suwerenności. Każde państwo musi szanować podmiotowość innych państw. Zakusy, deklaracje o federalizacji Europy, która właśnie odebrałaby Polsce suwerenność, są nie do zaakceptowania. Dziękuję bardzo. Głos teraz zabierze pan poseł Sławomir Nitras. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polska w roku 1989 odzyskała niepodległość. Stworzyliśmy system bezpieczeństwa, doprowadziliśmy do wstąpienia Polski do NATO. Wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, pamiętając o tym, że Europa będzie silna tylko wtedy, kiedy okiełznane będą interesy pojedynczych państw na rzecz interesów Wspólnoty. Stworzyliśmy format weimarski po to, żeby Polska wraz z Francją i z Niemcami odgrywała kluczową rolę w Europie. Stworzyliśmy format wyszehradzki i, szerzej, format współpracy w ramach Europy Środkowej, wiedząc, że jesteśmy buforem przeciwko zagrożeniu ze Wschodu - to zagrożenie, które w latach 90., na początku tego wieku było zagrożeniem bardziej teoretycznym niż praktycznym - wiedząc, że przyjdzie kiedyś moment, kiedy zagrożenie niedemokratyczne ze Wschodu będzie zagrożeniem realnym. To zagrożenie realne dzisiaj nadeszło: to, co dzieje się na Ukrainie. Problem polega na tym, że w tym czasie polski rząd, który obecnie nastał, nie stworzył tego systemu. Rozmontowuje system bezpieczeństwa demokratycznej Europy. Rozmontowuje Unię Europejską. Rozmontowuje nawet NATO. Pani Le Pen, która jest waszym sojusznikiem, opowiada się wprost za rozmontowaniem NATO. Jeśli nie będzie NATO i nie będzie Unii Europejskiej, zostaniecie sobie z tą zwiększoną armią na wschodniej granicy i polski żołnierz będzie musiał sam stanąć naprzeciw rosyjskiej potęgi. To jest droga ku przepaści, którą mogli stworzyć tylko ludzie zarządzający armią, którzy kierują się bożoojczyźnianą retoryką, a w głowie mają sieczkę. Proszę o zabranie głosu pana posła Tadeusza Tomaszewskiego. Wysoki Sejmie! Szanowni Panowie Ministrowie! Minister spraw zagranicznych przed chwilą mówił o tym, że Polska nadaje ton pracom w Unii Europejskiej, jest w głównym nurcie polityki europejskiej, walczy o polskie interesy w Unii Europejskiej. Z informacji medialnych wynika, że we wtorek polski ambasador próbował zablokować plan priorytetów legislacyjnych Unii Europejskiej na rok 2022. Powodem było niezaakceptowanie polskiego Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską. Dokument został przyjęty mimo sprzeciwu Polski i Węgier. Chciałem zapytać, jakie sprawy na tym posiedzeniu, jakie punkty programu legislacyjnego Unii Europejskiej były blokowane przez Polskę. Z jakich powodów? Lewica od początku stała za prawem Polek, Polaków i polskich przedsiębiorców do pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, Funduszu Odbudowy. Od początku pracy w tym parlamencie w tej kadencji staliśmy za tym funduszem i głosowaliśmy. Chciałem zapytać pana ministra Budę, czy łatwiej będzie panu walczyć o szybsze uruchomienie pieniędzy z KPO, jeśli kolejni ministrowie rządu koalicyjnego tzw. Zjednoczonej Prawicy będą nawoływać publicznie, aby Polska nie płaciła składki do Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, panie ministrze.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Tak naprawdę pan minister Buda przyznał, że politykę zagraniczną Polski w Europie i świecie kształtuje opozycja, a nie rząd. To jest rzeczywiście smutna konstatacja. Chciałem pana premiera zapytać: Dlaczego pan premier w Brukseli zgłaszał propozycję wspólnych podatków, a więc chodzi o pozatraktatową federalizację Unii Europejskiej, zgłaszał propozycję i zgodził się na to dwa razy, jeśli chodzi o wspólne kredyty i zobowiązania? A jednocześnie w Polsce wszystkim tłumaczy, że jest za Europą ojczyzn i przeciwko federalizacji. Chcę więc zapytać, kiedy rzeczywiście zostaną uruchomione środki na Krajowy Plan Odbudowy. Bo te pieniądze w Hiszpanii, 19 mld euro, już pracują. A to jest porównywalne państwo. Czas najwyższy więc, żeby pan premier jasno oświadczył, o czym informuje i na co zgadza się w Brukseli. Bo tam jest zdecydowanym federalistą i to już udowodnił wielokrotnie, podejmując tam decyzje. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana posła Pawła Zalewskiego, Polska 2050. Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Fakty mówią więcej, panie ministrze, niż słowa. Zamiast starać się o wzmocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej, stawiacie na jej osłabienie, budując front z tymi, którzy są agentami Putina. To nie są frazesy, pani poseł. To nie są frazesy. Pani Le Pen, która jest waszym sojusznikiem. na której zwycięstwo wyborcze w wyborach prezydenckich stawiacie, jest osobą, która pojechała do Krymu, akceptuje aneksję Krymu. Pan premier Orbán tak naprawdę jest wykonawcą woli Kremla i Pekinu w Europie. Otóż osłabiacie Unię Europejską.

Doprowadzacie do tego, że głos Polski nie jest słuchany na równi z głosami z Paryża, Berlina, Londynu czy Rzymu. Zamiast korzystać z szans rozwojowych, które daje Unia Europejska, zadłużacie się w Chinach.

Teraz konkluzja.

Jeżeli partia rządząca stawia swój interes ponad interes narodu, będzie potępiona przez przyszłe pokolenia Polaków. Proszę o zabranie głosu panią poseł Katarzynę Czocharę. Panie pośle Zalewski, proszę nie wychodzić, bo chciałam panu powiedzieć, że w jednej kwestii muszę się z panem zgodzić. Jakie są fakty dotyczące polityki, którą prowadziło PSL? Mówił pan, panie przewodniczący, o zamachu stanu.

Szanowni Obywatele! Dzisiaj z powodu właśnie tych decyzji, decyzji polityków opozycji, ponosicie tak wysoką cenę. Wy jesteście temu winni.

Dziękuję. Głos zabierze pan poseł Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska. W tej debacie w gruncie rzeczy chodzi tylko o jedną sprawę. Które deklaracje rządu są prawdziwe? Jedna polityka to polityka zwoływania w Warszawie proputinowskiego sabatu z Marine Le Pen.

To jest wasz wielki błąd, którego nie da się zapomnieć. Ta sama polityka to tolerowanie tego, że Putin chce zbudować nowe imperium i nowy Związek Sowiecki. Pani sobie potem powie. My chcemy Polski, która bierze udział w dyskusji na temat polityki wschodniej. My mówimy: tak dla silnych instytucji europejskich, dla sądu europejskiego, dla Komisji Europejskiej, bo wiemy, co to jest polska racja stanu. Polska racja stanu może być budowana przez wspólne instytucje europejskie, panie Macierewicz. Tak, pan kiedyś też tak uważał. Polska racja stanu to bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a nie budowanie mościków po cichu z Chinami. Pan pierwszy powinien być przeciwko. Polacy muszą usłyszeć, że wy to robicie. Musicie się wreszcie zdecydować, po której stronie jesteście. w tym strategicznym sporze o bezpieczeństwo Polski. Proszę o zabranie głosu pana posła Rafała Adamczyka. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiaj z tej mównicy chciałem zapytać o koszty promocji Polskiego Ładu.

Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Jarosława Rzepę. Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Dobra i roztropna polityka zagraniczna to skuteczna polityka zagraniczna. Co mamy ze skutecznej polityki zagranicznej? Brak środków z KPO. Zlikwidujcie Izbę Dyscyplinarną, to środki będą. Nie będziemy płacić dodatkowych kar. Druga sprawa. Pan poseł Kowalski proponuje zawieszenie handlu emisjami.

Szanowni państwo, to jest bardzo niebezpieczne.

W nowej perspektywie praktycznie nie ma nic. Kiedy wreszcie, szanowni państwo, panie ministrze, zaprzestaniecie tej antyunijnej polityki, która naprawdę doprowadzi nas do katastrofy? Jeden przykład: tunel w Świnoujściu, 770 mln ze środków spójności, 125 mln ze środków samorządu miasta Świnoujście. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Roberta Winnickiego. Wysoka Izbo! Wspólnota państw demokratycznych nie istnieje, układy multilateralne są złudą, są fikcją. To nie Polska zdradziła Ukrainę, to zrobiły Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, to zrobili gwaranci nienaruszalności granic ukraińskich, ci z początku lat 90.

Przestańcie żyć złudzeniami, przestańcie żyć mitami. Jest pięć wektorów, wokół których polska polityka zagraniczna musi się koncentrować. Pierwszym wektorem są relacje z Berlinem jako dominującym graczem w Europie, drugim są oczywiście (Dzwonek) relacje czy poziom konfliktu z Moskwą, trzecim elementem są relacje ze Stanami Zjednoczonymi, czwartym elementem są relacje z Pekinem i piątym elementem jest współpraca regionalna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. I te relacje ze stolicami mocarstw w nowym koncercie mocarstw, który rzeczywiście ma miejsce i który rzeczywiście jest dla nas niebezpieczny, to jest podstawa naszej polityki zagranicznej. Unia Europejska jest wyłącznie narzędziem, a nie wartością, i to jest narzędzie, które dzisiaj spoczywa w całości w niemieckich rękach. Nie służy ono naszym interesom, bo gdyby służyło, toby nie było dyrektywy transportowej, nie byłoby Nord Streamu, nie byłoby wielu innych rzeczy, a są. Przestańcie żyć złudzeniami. Czy jest pan poseł Mirosław Suchoń? Jeżeli nie, proszę o zabranie głosu pana posła Marcina Duszka. Też nie ma. Proszę. Panie Marszałku!

Po drugie, panowie ministrowie niezwykle mi zaimponowali, mówiąc o tym, że realnie walczymy o polskie interesy w Unii Europejskiej. A gdzie są pieniądze z KPO, panie ministrze? Jedyny ślad po pieniądzach z KPO jest na tych propagandowych billboardach, gdzie ogłaszaliście wielkie inwestycje. Zero. Zero, panie ministrze, i z tego pan się powinien rozliczyć.

A kto zapłaci blisko 200 mln zł kary, panie ministrze, za Turów? Gdzie jest ta dyplomacja? Dlaczego przez ponad rok nie było ambasadora w Czechach, który powinien zabiegać o polskie interesy? I pan teraz, rozmawiając przez telefon, kiedy ja do pana mówię, pokazuję tę ignorancję i pokazuje to, że tak naprawdę nie myślicie o tym, jak skutecznie walczyć o polskie interesy, tylko myślicie o tym, jak uprawiać tę tandetną propagandę. Na końcu przecież za to wszystko zapłacą Polacy.

Pan poseł Jan Szopiński teraz zabierze głos. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nikt z nas tu obecnych nie ma wątpliwości co do tego, że pan minister Ziobro jest człowiekiem ambitnym i, jak sądzę, widzi siebie na stanowiskach o wiele wyższych niż obecnie zajmowane. Niestety od czasu do czasu swoje ambicje przelewa na papier, co wywołuje czasami bardzo negatywne skutki dla naszego kraju. Chciałbym zapytać, czy pan minister Ziobro posiadał stosowne umocowania pana premiera do wystąpienia do przewodniczącej Komisji Europejskiej pani Ursuli von der Leyen z żądaniami wyjaśnienia sytuacji związanych z nieprawidłowościami w TSUE opisywanymi przez francuską prasę? Jeżeli nie, to chciałbym zauważyć, że pełni pan minister funkcję prokuratora generalnego, i zastanawiam się, czy w ramach pańskich kompetencji leży kierowanie wezwań do składania wyjaśnień do prezydentów czy premierów innych państw, krajów, jak i do władz Unii Europejskiej. Panie ministrze, na wyjaśnienie w pańskim resorcie czeka sprawa Funduszu Sprawiedliwości, wyborów kopertowych, sprawa (Dzwonek) dwóch wież, czeka sprawa pana Mejzy. A co do upoważnienia pana ministra do wystąpienia do pani Ursuli von der Leyen, uprzejmie poproszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Głos teraz zabierze pan poseł Dariusz Klimczak. Wysoka Izbo! Podczas dzisiejszej debaty doszło do sytuacji niebywałej w historii polskiego parlamentaryzmu. Otóż kiedy prezes ludowców mówił o wzmocnieniu polskiej polityki zagranicznej, priorytetach i strategii, jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości zaczął intonować hymn Niemiec. Niebywałe. PiS ma na swoim koncie bardzo wiele porażek: ochrona zdrowia, rolnictwo, energetyka, ale perłą w koronie waszych porażek jest polityka zagraniczna. Przykładem chociażby pieniądze na KPO - ich brak bardzo silnie oddziałuje na polską gospodarkę, na bieżące funkcjonowanie polskich przedsiębiorców, np. z Podhala. Jak nasi przedsiębiorcy mają z nimi konkurować? Do kogo przyjadą goście? Kto będzie miał lepsze warunki? To jest wasza zasługa. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Polityka Unii Europejskiej w różnych zakresach zakłada, że kierunki i zakres działań powinny być podobne w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jednocześnie oczywiste jest, że polityka ta powinna uwzględniać krajowe ograniczenia, m.in. finansowe, punkty wyjścia i inne preferencje krajowe, rządowe. Stawiam pytanie, jak pan minister ocenia traktowanie Polski w Unii Europejskiej w różnych zakresach. Czy tak samo są traktowane wszystkie kraje np. w sprawach, w których zapadły niekorzystne wyroki? Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Koledzy i Promotorzy Mejzy! Zapisać i zadeklarować można wszystko. Wy też wielokrotnie powtarzacie, że Polska odgrywa dzisiaj jakąkolwiek rolę w Unii Europejskiej, że wzmocniła swoją pozycję w ciągu ostatnich 6 lat. Każdy, kto przynajmniej potrafi przeczytać prosty artykuł w gazecie, widzi, że wszystko, co dało się zepsuć, a w zasadzie zlikwidować, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, w ciągu tych 6 lat wy dokładnie zepsuliście. Tu patrzę na pana ministra Macierewicza.

To wy zorganizowaliście w Warszawie zlot polityków (Dzwonek), którzy są wprost proputinowscy w całej Europie, i to wy zorganizowaliście spotkanie w Warszawie jedynych proputinowskich polityków. Przecież Marine Le Pen mówi wprost, że Ukraina powinna być w sferze wpływów rosyjskich, mówi wprost, że Rosja powinna być pozbawiona sankcji. A więc to wy koordynujecie proputinowską politykę wewnątrz Unii Europejskiej, wy, także pan, panie Macierewicz, i także cały rząd. Czy ta polityka jest po prostu wynikiem głupoty, czy jest zainspirowana z zewnątrz? Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Zdzisława Wolskiego. Mam pytanie do rządu, do pana premiera. Jak długo będzie jeszcze kontynuowana polityka pogarszania relacji Polski z Unią Europejską, a szczególnie z Niemcami?

Przypominam rok 1965 i słynny list biskupów polskich do biskupów niemieckich: wybaczamy i prosimy o wybaczenie. To był bardzo konkretny, wielki ruch mający na celu pojednanie między narodami po II wojnie światowej. Te starania były kontynuowane.

Nic z tego nie będzie, miejmy tę świadomość.

Miejmy tego świadomość. Kończę i powtarzam pytanie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Dobrym zwyczajem tej Izby była doroczna informacja ministra spraw zagranicznych o kierunkach polskiej polityki zagranicznej. Zniknął ten temat w ogóle z agendy polskiego Sejmu. Polski parlament nie dyskutuje o kierunkach polskiej polityki zagranicznej. Sejm jest tym miejscem, gdzie powinna być podejmowana przynajmniej próba kształtowania tej polityki i budowania pewnego konsensusu. Po drugie, dobre relacje z USA i z Unią Europejską powinny stanowić core naszej polityki zagranicznej, plus współpraca regionalna. Tego nie widzę. Widzę raczej, że tak powiem, krytykę czy jakieś przeżycie traumatyczne po prezydenturze Trumpa i jednocześnie dużą krytykę obecnej administracji Bidena. Nie mamy na to wpływu. To wyborcy amerykańscy zdecydowali, jaka ma być tam administracja.

Wysoka Izba nie była miejscem prezentacji Krajowego Planu Odbudowy. Owszem, zatwierdziliśmy fundusz. W jaki sposób mamy wesprzeć polski rząd w staraniach o to, żeby ten Krajowy Plan Odbudowy został odblokowany? Polska Izba, polski parlament, była w ogóle z tego procesu wyłączona.

Konsekwencje również mogą być dla polskiego budżetu. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana posła Grzegorza Wojciechowskiego. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wrócę do kryzysu imigracyjnego, do tego kryzysu, który trwa na polskiej granicy, i do wcześniejszych. We wcześniejszych kryzysach, które nie dotykały Polski, a dotykały innych krajów Polska miała przyjmować migrantów -13 tys., 10 tys. później 3 tys. czy 2 tys. W tej chwili Polska zablokowała, bardzo skutecznie zablokowała dopływ migrantów i otrzymała duże wsparcie zarówno ze strony Komisji Europejskiej, jak i ze strony poszczególnych państw członkowskich, co jest najważniejsze, i to państw członkowskich, które przy poprzednich kryzysach wpływały na Polskę, aby migrantów przyjęła.

Proszę o zabranie głosu panią poseł Kamilę Gasiuk-Pihowicz. Wysoka Izbo! Dzisiaj w rządzie PiS nie ma premiera, nie ma ministra spraw zagranicznych, nie ma ministra do spraw Unii Europejskiej. Wszyscy oni abdykowali i oddali władzę jednemu człowiekowi - Zbigniewowi Ziobrze, który okopał się w Ministerstwie Sprawiedliwości i stamtąd dowodzi wojnie hybrydowej z Unią Europejską. Przez niego i jego kilku posłów z partyjki, która nawet nie ma 1% poparcia społecznego, Polacy i Polki tracą miliardy z KPO. Dlaczego? Bo Ziobro, PiS chcą trzymać sądy pod batem politycznym, jakim jest de facto Izba Dyscyplinarna, i zapewnić sobie i swoim kolegom w ten sposób bezkarność. Ponieważ minister sprawiedliwości uznał, że posady dla kilkorga jego zaufanych w Izbie Dyscyplinarnej, w neo-KRSie (Dzwonek) są ważniejsze niż pieniądze na rozwój, na służbę, na energetykę, na informatyzację. To są najdroższe posady na świecie. Każda z nich kosztuje kilka miliardów euro. Co znaczy jego słowo?

Tę ustawę trzeba natychmiast uchwalić, a odrzucanie tych rozwiązań, bezczynność rządu świadczą o tym, że Ziobro, że Kaczyński po prostu nie chcą pieniędzy dla Polaków. Proszę o zabranie głosu pana posła Aleksandra Mrówczyńskiego. Bardzo słuszna uwaga. Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Odpowiem na pani pytanie: rządzi rząd Zjednoczonej Prawicy z panem premierem Mateuszem Morawieckim i proszę nie obrażać w takich wypowiedziach pana premiera i polskiego rządu. Wysoka Izbo! Dobrze, że dzisiaj jest realizowana ta informacja bieżąca, w której polscy parlamentarzyści winni się określić, określić swój stosunek dla Polski, do naszej ojczyzny. Toczy się spór w Europie, czy Europa państw narodowych, czy Europa federalna. Czy Europa wartości, w których człowiek jest najważniejszy, czy Europa antywartości? Proszę wsłuchać się w słowa. Więcej szacunku.

Polska znikająca. Przez 123 lata brakowało Polski na mapie, to wystarczająco długo. Dosyć. Opowiedzmy się w sposób jednoznaczny: Polska wartości, Polska niepodległa, Polska suwerenna, żeby Polska była polska, a Europa - Europą wartości, Europą państw narodowych. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią poseł Barbarę Nowacką. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z prawej strony słyszymy tyle o wartościach europejskich. Czy wy wiecie, że te wartości to prawa człowieka, to dostęp do wolnych mediów, to demokracja, to szacunek do prawa, to prawa kobiet, to otwartość i tolerancja? To pod tymi wartościami obywatelki i obywatele Rzeczypospolitej podpisywali się, wstępując do Unii Europejskiej. To tych wartości Unia Europejska i NATO chcą bronić. A wy co? Wy pod dyktatem Ziobry uderzacie w polskich przedsiębiorców i w polskich pracowników. A wszystko to jest polane narodowo-patriotycznym bogoojczyźnianym sosem, a tak naprawdę - pisane cyrylicą. Ustawy, które przychodzą, uderzające w kobiety, uderzające w społeczność LGBT są ustawami toczka w toczkę - to może państwo zrozumiecie - wziętymi od Putina. Jak chcecie budować wspólnotę z tą Unią?

Przez to społeczności tracą pieniądze. To wy uchwalacie przepisy, przez które Polki w Polsce zwyczajnie są torturowane, umierają. To wasze przepisy powodują, że społeczność międzynarodowa, tak jak Czesi, chce nam pomóc. A co na to polska dyplomacja? Znowu walnie w kobiety. Jeżeli tyle mówicie o wspólnocie, to spójrzcie wokół siebie.

Głos zabierze pan poseł Paweł Hreniak. Jeżeli nie ma, to pan poseł Dariusz Rosati.

Panie Marszałku! Właściwie nie ma się co dziwić w sytuacji, gdy pana ministra spraw zagranicznych w ogóle nie widać, pan premier pokazuje inną twarz tam, inną tu, a właściwie za sznurki pociąga pan Zbigniew Ziobro. Pan minister Wawrzyk mówił o sukcesach Polski, więc przypomnę, że jeśli chodzi o tak ważną sprawę jak obsada stanowisk w instytucjach unijnych, to jakoś nic wam nie wychodziło. No brawo.

Może rozejrzyjcie się wśród własnych szeregów. Gdzieś tam te przyczyny znajdziecie.

Z waszego obozu politycznego płyną głosy o okupacji brukselskiej.

Panie Pośle! Co z tego, że obsadziliście cztery komisje?

To jest prawda niepowtarzalna, niepodważalna. Tak, to niepowtarzalny przypadek.

Dlatego pragnę zapytać, panie ministrze, w jaki sposób Polska będzie w nadchodzących latach budować spójną politykę gospodarczą i fiskalną Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pani poseł Małgorzata Tracz. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Największym problemem polskiej polityki zagranicznej jest to, że stała się zakładniczką grupy radykałów ze Zjednoczonej Prawicy. De facto to politycy tacy jak Janusz Kowalski tutaj obecny wyznaczają kierunki polityki i strategię rządu względem polityki klimatycznej Unii Europejskiej i ośmieszają Polskę na arenie europejskiej. Przykładem jest podjęta ostatnio haniebna uchwała, która wzywa państwa europejskie do zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Ten system to główny sposób na osiągnięcie celów klimatycznych i realizację strategii Fit for 55, która wynika z Europejskiego Zielonego Ładu, który poparł premier Morawiecki. Środki ze sprzedaży uprawnień to przychody budżetu państwa.

One mogą być kołem zamachowym polskiej gospodarki, a wy te miliardy euro chcecie Polkom i Polakom zabrać, tak samo jak zabraliście środki z Krajowego Planu Odbudowy. I tu moje pytanie do rządu: Kiedy przestaniecie ulegać radykałom i prowadzić politykę zagraniczną pod ich dyktando?

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W ostatnich dniach media całej Europy, w tym także polskie, szeroko informują o zjawiskach obrzydliwej korupcji szerzącej się wśród polityków Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska i, panie pośle wnioskodawco, Polskie Stronnictwo Ludowe. Oczywiście oszczędny w tej kwestii jest TVN. W tym samym parlamencie regularnie toczą się dyskusje na temat praworządności Polski i Węgier, które szkodzą polskiej racji stanu, a z drugiej strony - ośmieszają politycznych przeciwników Polski. Polska jest chyba jedynym państwem, którego przedstawiciele krajowej opozycji atakują na forum Unii Europejskiej swój własny kraj. Opozycja nie wspiera Polski w sytuacjach, kiedy Komisja Europejska wstrzymuje akceptację polskiego Krajowego Planu Odbudowy i w konsekwencji wypłatę ok. 58 mld euro dla Polski. Europosłowie opozycji wielokrotnie organizowali w Unii Europejskiej nagonkę na Polskę. Kiedy kilka tygodni temu premier Morawiecki tak spokojnie, merytorycznie bronił polskich interesów na forum Parlamentu Europejskiego, europosłowie Koalicji Europejskiej wypowiadali się, jakby nie byli Polakami. Bardzo proszę, panie ministrze, o przedstawienie strategii rządu w sprawie wykazania Komisji Europejskiej zaniechania i bezpodstawnego dalszego blokowania tak ważnych dla Polski funduszy. Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Unia Europejska, wbrew temu, co zostało tutaj powiedziane, jest wartością.

Jest w Unii Europejskiej. Jeśli państwo uważają, że nie powinniśmy być w Unii Europejskiej, złóżcie taki wniosek. Zobaczymy, co odpowiedzą wam obywatele naszego kraju. Wtedy będziemy mieli jasność. Przywołujecie tutaj jakieś bzdurne debaty na temat tego, że Europa chce się stać federalistyczna. Od kilkudziesięciu. Stało się coś? Nic się nie stało. Jeżeli sami chcemy być szanowani, musimy także okazać szacunek tej instytucji, w której jesteśmy.

Wysoka Izbo! Totalna Opozycjo! Panie Pośle Zwiefka! To tak na marginesie. Szanowni Państwo! Wielokrotnie na tej sali słyszymy ze strony ław opozycji totalnej o rzekomym polexicie wywołanym niewykonywaniem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podkreślamy: jednego orzeczenia, który godzi w polską rację stanu, w polskich obywateli i polski interes gospodarczy. Traktaty jasno określają kompetencje Unii Europejskiej, kompetencje dzielone oraz te pozostające w dyspozycji państw członkowskich. Rolą każdego rządu jest dbanie o interes własnego kraju. Jest to całkowicie zrozumiałe. Niemiecki sąd konstytucyjny przyznał, że narodowe sądy muszą interweniować w rzadkich sytuacjach nadzwyczajnych, gdy dochodzi do poważnego naruszenia kompetencji. Czy o Włoszech, Grecji, Niemczech mówimy jak o zagrożonych erozją demokracji? A przecież liczba niewykonywanych wyroków TSUE jest tam zdecydowanie wyższa. Może to także wynik podwójnych standardów, które popiera Platforma Obywatelska, stosowanych przez aparat unijny niedopuszczający do dyskusji nad stanem praworządności w krajach Europy Zachodniej. Wysoka Izbo! Totalna Opozycjo! Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie: Jak polski demokratyczny rząd zamierza radzić sobie z narzuceniem formatu Europy dwóch prędkości pod względem interpretacji pojęcia „praworządność” Głos zabierze pan poseł Piotr Borys.

Wysoka Izbo! Wasz słaby rząd osłabia pozycję Polski na arenie europejskiej, na arenie światowej. Jesteście pierwszym w historii 30 lat rządem, który złamał świętą zasadę, że priorytety polskiej polityki zagranicznej są wspólnym celem całej klasy politycznej. Wybieracie sojusz z Putinem poprzez sojusze z Le Pen, Salvinim czy Orbánem. To jest po prostu niedopuszczalne. Osłabiacie w ten sposób bezpieczeństwo Polski.

Polska w Unii Europejskiej, trwały sojusz w ramach współpracy Trójkąta Weimarskiego - tego nie ma. Grupa Wyszehradzka stała się fasadą. Partnerstwo Wschodnie zostało zdewastowane. Nie jesteśmy już ambasadorem bezpieczeństwa Ukrainy i demokratyzacji Białorusi, ale tak naprawdę, nawet w tak prostych sprawach jak kwestia współpracy z Czechami... 1,5 roku nie potrafiliście wybrać ambasadora. Dzisiaj kary to ponad 200 mln zł. Moje pytanie: Kto za to zapłaci? Premier Morawiecki czy premier Sasin?

Głos zabierze pani poseł Gabriela Masłowska. Jest?

Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polityka zagraniczna to przede wszystkim skuteczność. To porównajmy skuteczność rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej i PSL-u. 2014 r. - szczyt klimatyczny, tak często tutaj podnoszony przez was, redukcja do 2030 r. CO2 o 40%. 30 mld dodatkowych, darmowych emisji dla polskiego przemysłu. Bo jakoś o tym nie mówicie. Słynna szarża pana premiera Morawieckiego na szczycie klimatycznym. I jakie efekty, szanowni państwo, po tej genialnej szarszy pana premiera Morawieckiego, panie Kowalski? I co wynegocjował dodatkowego dla polskiego przemysłu? Drożyzna, ceny energii idą w górę, bo nie potraficie załatwić nic dla polskich interesów. Dziękuję bardzo. Głos zabierze teraz pani poseł Teresa Pamuła. Szanowni Państwo! Jestem dumna z tego, co robi rząd Rzeczypospolitej Polskiej. To, że liczą się wszyscy z nami. Wszyscy się liczą z nami w Polsce. Proszę się nie śmiać. Jesteśmy osobami, które chcą narzucić pewien stan demokracji w Unii Europejskiej. Chcemy, aby w Unii Europejskiej było ważne wszystko, co jest ważne dla nas, dla rodzin, dla kobiet, dla gospodarki, dla wszystkich. My dążymy do tego, żeby opozycja. Naprawdę najgorszy jest wróg w swoim własnym domu, który donosi, mówi nieprawdę, zaprzecza wszystkiemu. Wiecie państwo o tym dobrze, że mówicie nieprawdę.

Głos zabierze pan poseł Andrzej Kryj. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na środki Krajowego Planu Odbudowy czekamy wszyscy, czekają polskie samorządy, czekają polscy przedsiębiorcy. Dotychczasowe wykorzystanie środków unijnych przez Polskę zostało bardzo dobrze ocenione zarówno przez Najwyższą Izbę Kontroli, jak i przez unijnych urzędników. Niestety nie to brane jest pod uwagę, lecz wypowiedzi i antypolskie głosowania europosłów totalnej opozycji czy choćby słowa Rafała Trzaskowskiego z 2018 r. o tym, że dzięki staraniom opozycji środki unijne nie przepadną, tylko będą zamrożone, a ich odmrożenie nastąpi wtedy, kiedy opozycja wygra wybory w Polsce. Mam pytanie: Czy panowie ministrowie zgadzają się z opinią, że blokowanie środków z KPO dla Polski nie ma merytorycznych podstaw, lecz jest motywowane politycznie i ma służyć odsunięciu PiS od władzy w myśl zasady, że ma to zrobić ulica i zagranica? I drugie pytanie, proszę państwa. Padały tutaj stwierdzenia, jakim to dobrodziejstwem było to, iż politycy Platformy odgrywali rolę w Europie Zachodniej, w Unii Europejskiej. Czy panowie ministrowie mają wiedzę, co Donald Tusk zrobił, żeby zatrzymać tak antypolską inwestycję, antyeuropejską inwestycję, jakim był Nord Stream 2? Głos zabierze pan poseł Daniel Milewski. Panowie Ministrowie! Po 2015 r. polskie ustawy budżetowe charakteryzują się możliwie niskim deficytem. Do momentu wybuchu pandemii spadało również zadłużenie państwa względem PKB. Tymczasem od 2012 r. widzimy politykę podwójnych standardów wobec budżetów państw przedstawianych z deficytem finansów publicznych powyżej 3% PKB.

Wtedy zakończyło się tylko na tłumaczeniach i dość śmiesznych unikach ówczesnych komisarzy, mówiących o jednorazowym przypadku i podkreślających silną rolę w kształtowaniu Unii Europejskiej przez Francję, cokolwiek to znaczy.

Proszę o zabranie głosu pana posła

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! W ostatnim czasie z mojego punktu widzenia wydarzeniem niebagatelnym były artykuły, seria artykułów we francuskiej gazecie „Libération”

To jest po prostu niezgodne z prawem europejskim, to jest korupcjogenne i dotyczy, tak jak mówiłem, najwyższych przedstawicieli Unii Europejskiej, chociażby komisarza do spraw budżetu. Do dzisiaj nie ma żadnej reakcji ze strony władz Unii, nie ma (Dzwonek) komentarza pani komisarz, nie ma komentarza prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I to zastanawia, bo mimo wszystko wszyscy wierzymy w demokrację unijną, prawda? Opinia publiczna i politycy, my wszyscy mamy prawo wiedzieć, co tam rzeczywiście się dzieje.

To nie jest jakaś gazeta prawicowa, która być może dla państwa byłaby niewiarygodna.

Dlatego jeszcze raz zwracam się do rządu z prośbą o to, żeby pan minister udzielił informacji, dlaczego tak naprawdę tego wyjaśnienia nie ma oraz czy my domagamy się na forach unijnych tego, żeby ta sprawa została dokładnie wszystkim obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej wyjaśniona i przedstawiona. tak żebyśmy nie mieli wątpliwości, czy chociażby sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po prostu biorą pieniądze za wyroki. Głos zabierze pan poseł Arkadiusz Mularczyk. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polskę i Niemcy łączą wielowiekowe relacje, a pamięć o naszej historii wciąż oddziałuje na współczesne relacje pomiędzy Polską i Niemcami.

Niemiec w sprawie właśnie dotyczącej zadośćuczynienia i rekompensat z tytułu II wojny światowej.

Należy podkreślić, że skutki II wojny światowej do dziś oddziałują na kondycję gospodarczą, społeczną, ekonomiczną naszego państwa.

A więc myślę, że są to sprawy, o których powinniśmy mówić jednym głosem. Dlatego też z pewnym zdumieniem przyjąłem wypowiedź kanclerza Niemiec, który stwierdził, że to środki unijne są rekompensatą czy też reparacjami dla Polski, jakie dzisiaj Unia Europejska, a tym samym Niemcy, wypłaca Polsce. Należy zapytać, czy składki unijne, które wpłacają Hiszpania, Portugalia czy też nawet Polska do budżetu Unii Europejskiej, są tymi reperacjami, które Polska otrzymuje, i czy Unia Europejska wypłaca też reperacje Hiszpanii czy Portugalii, które przecież nie były sprawcami II wojny światowej. Jestem pełen uznania dla polskiego rządu, że ten temat po raz pierwszy w sposób tak jasny i zdecydowany został podniesiony na arenie międzynarodowej właśnie w relacjach z nowym rządem Niemiec.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Pan Putin w tym wywiadzie w rocznicę wybuchu II wojny światowej stwierdził, że perspektywą dla Europy i dla Rosji jest sojusz i zastąpienie Unii Europejskiej jako struktury europejskiej sojuszem z Rosją. I to jest właśnie polityka, którą od tamtego czasu prowadzi Koalicja Obywatelska.

Przepraszam bardzo. Proszę umożliwić posłowi zabranie głosu. Nawet jeżeli pan poseł się nie zgadza, to proszę, aby pan poseł Macierewicz miał szansę zabrać głos. Nawet wówczas prowadzicie tę politykę, gdy nowy rząd niemiecki jasno deklaruje, że dąży do tego, żeby zamienić Unię Europejską w państwo niemieckie. Jest to zapisane w porozumieniu między partiami, które tworzą ten rząd. Co więcej, jest jasno powiedziane, że fundamentalnym kierunkiem polityki niemieckiej jest budowa Nord Stream 2, która jest infrastrukturą gospodarczo-polityczną łączącą na trwałe Rosję i Niemcy. To my, to formacja niepodległościowa doprowadziła do tego, że Polska weszła do NATO. Byliście temu przeciwni. Byliście temu przez cały czas przeciwni. Obaliliście rząd Jana Olszewskiego, który właśnie to realizował. Byliście przeciwni temu. Panie marszałku, jeżeli pan marszałek nie umożliwi mi tego przez wyciszenie ludzi, którzy za wszelką cenę chcą kłamać.

Ja jestem tylko skromnym posłem. Tak... ...że ci ludzie, którzy niszczą Polskę, mogą teraz także uniemożliwiać mówienie prawdy.

Wysoka Izbo! Mamy dzisiaj ze strony Platformy Obywatelskiej reklamę zdrady narodowej. Mamy dzisiaj ze strony Platformy Obywatelskiej próbę wymuszania podporządkowania się dominacji rosyjsko-niemieckiej.

Panie pośle Nitras, proszę usiąść. A panu Antoniemu Macierewiczowi bardzo serdecznie dziękuję. Głos zabiera teraz pani poseł Anna Kwiecień. Panie marszałku, proszę wybaczyć.

Pani poseł Anna Kwiecień zabiera głos. Proszę zakończyć swoją wypowiedź. A pana proszę o opuszczenie mównicy, bowiem przekroczył pan już trzykrotnie swój czas. Głos zabiera teraz pani poseł Anna Kwiecień.

Głos zabiera pani poseł Anna Kwiecień.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Opozycja bardzo często wymienia nazwisko pani Le Pen, twierdząc, że jest politykiem prorosyjskim.

To jest pierwsza sprawa.

Wysoka Izbo! Bardzo dobrze, że dyskutujemy dzisiaj na temat polityki międzynarodowej, bo ona musi przede wszystkim być prowadzona na zasadzie partnerstwa, nie poddaństwa i niewolnictwa.

Mamy 100 lat niepodległości, nasi przodkowie przelewali krew za ojczyznę, a państwo z Koalicji Obywatelskiej wybieracie ulicę i zagranicę, żeby szkodzić Polsce. Jak można?

To jest skandal. Państwo (Dzwonek) musicie wspólnie z nami dbać o interes Polski, a nie o interes krajów zachodnich. Panie marszałku, proszę mi nie przerywać wystąpienia. Nikomu pan nie przerywał, gdy tutaj obrażali moich kolegów, mojego premiera, premiera Polski, i polski rząd. A pan mi przerywa i mówi nieprawdę. Ja sobie nie życzę. I jeszcze chcę dokończyć pytanie, bo pan mi uniemożliwił zadanie pytania. Proszę wreszcie zdementować te wszystkie wypowiedzi i hipokryzję naszych kolegów i koleżanki z opozycji. Opamiętajcie się. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałam na początku odpowiedzieć. Pani poseł, bardzo proszę o chwilkę, jeśli pani pozwoli. Chciałbym prosić także posłów z tej strony i z tej o wyciszenie emocji, umożliwienie zadania pytania pani poseł. Chciałabym na początek odpowiedzieć pani poseł Nowackiej. My bronimy, jako prawica, konstytucyjnego prawa do życia. Bronimy konstytucyjnego prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a wasze samorządy tolerują tortury i przemoc wobec młodzieży - przykład: Renice. Panie prezesie Kamysz, nic z pańskich tez nie jest ani prawdziwe, ani obiektywne, przykro mi. Polska prowadzi racjonalną i optymalną politykę zagraniczną, opartą na rozwoju gospodarczym, na bezpieczeństwie wewnętrznym i zewnętrznym, na solidaryzmie pokoleń i solidarności wewnętrznej. Czy boli was rozwój Polski? Pytanie do pana ministra: Jakie są cele strategiczne obecnej polityki zagranicznej Polski? Bardzo dziękuję.

Chcieliście państwo debaty? Macie debatę. Kilka słów prawdy usłyszeliście, stąd te wasze reakcje i ten śmiech, też taki szyderczy, ale szyderstwo i pogarda zawsze były po waszej stronie. Proszę państwa, dużo mówiliście tutaj o takich inicjatywach jak Grupa Wyszehradzka. Chciałabym przypomnieć, jak się zachowała wasza pani premier Ewa Kopacz w roku 2015, kiedy oszukała całą grupę.

Zrewidowaliście te swoje decyzje, tak samo i inne kraje Europy, bo wiemy, do czego to multikulti doprowadziło. Chciałabym zapytać o jeszcze jedną inicjatywę (Dzwonek), jakże ważną dla nas, dla Europy Środkowej, a mianowicie o inicjatywę Trójmorza.

Gdyby pan zechciał powiedzieć więcej o tej inicjatywie, jak ona wygląda teraz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Po reakcjach posłów opozycji widać, że prawda boli. Opozycja w Polsce przez 6 lat, obserwując działania rządu Prawa i Sprawiedliwości na polu dyplomacji, miała okazję wiele się nauczyć, ale jak widać, z tej okazji nie skorzystała. Albo jest leniwa, albo zwyczajnie nie chce czerpać z dobrych praktyk. Jak wyglądała polityka zagraniczna w Polsce za rządów Platformy i PSL-u? Wasalizacja Polski, usłużne zgadzanie się na wszystko bez względu na konsekwencje. Zgodnie z waszą polityką dziś mielibyśmy setki tysięcy uchodźców w kraju, a chcieliście przyjąć nawet milion. Mówiliście, że jesteście gotowi na każdą liczbę uchodźców. Prosicie o nakładanie sankcji na Polskę, podpisujecie deklaracje, wywołujecie rezolucje w Parlamencie Europejskim (Dzwonek) przeciw własnemu krajowi. I w tym jesteście konsekwentni, to trzeba wam przyznać. Tylko dlatego, że nie możecie zaakceptować demokratycznego wyboru Polaków. Czy z zemsty za to, że Polacy odsunęli was od władzy, dzisiaj szkodzicie polskim interesom? Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Porozmawiajmy o rządzie Donalda Tuska, o tym co zrobił dla Władimira Putina. W lutym 2008 r. reset z Putinem, spotkanie z Putinem. Dewastacja polityki śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego na wschodzie, zdrada naszych sojuszników, zdrada Litwy, zdrada państw bałtyckich, Gruzji, Azerbejdżanu. Zatrzymanie projektu Odessa - Brody - Płock - Gdańsk. Zatrzymanie Baltic Pipe, bo chcieliście kupować rosyjski gaz i zrobiliście to. W 2010 r. zawarliście umowę, która była proputinowska.

Tak właśnie Donald Tusk i Waldemar Pawlak przysłużyli się Putinowi. I nawet w marcu 2014 r. Donald Tusk zgodził się na ten fatalny system EU ETS, [[Dzwonek]] który dzisiaj powoduje, że mamy takie wysokie ceny energii i ciepła. S Szanowni Państwo! Mieliście okazję w zeszłym tygodniu zagłosować za stanowiskiem Polski, bo jutro pan premier jedzie walczyć o to, żeby ten system, który jest zdewastowany przez waszą politykę, zawiesić po to, żeby były niskie ceny energii i ciepła. Znowu zagłosowaliście za wysokimi cenami energii, znowu zagłosowaliście za stanowiskiem Berlina i Moskwy, bo gaz dzisiaj jest polityką, którą wspiera Moskwa i wspiera Berlin. Prawda boli. Donald Tusk był najbardziej proputinowskim premierem III RP. Głos zabierze pani poseł Ewa Szymańska. Szanowny Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Brawo, panie pośle, mój kolego klubowy. Fakty mówią więcej niż słowa. My chcemy Polski, która bierze udział w dyskusji na temat polityki wschodniej. Takie hasła dziś wybrzmiały z ust posłów opozycji. Ale to na skutek naszych działań zmieniło się podejście Unii do kryzysu migracyjnego. My, będąc jeszcze w opozycji, nie godziliśmy się na przyjmowanie migrantów z Unii zaproszonych szerokimi falami przez byłą kanclerz Angelę Merkel. My działamy, nie tylko mówimy. I to są fakty, fakty mówiące o tym, że teraz to my kształtujemy unijną politykę migracyjną. To my, Polska, chronimy wschodnich granic Unii Europejskiej przed nielegalnym napływem migrantów. Zarzucacie nam proputinowskie działania (Dzwonek), a przecież to wasz człowiek, Donald Tusk, był człowiekiem Putina w Warszawie. Głos zabierze pan poseł Grzegorz Lorek. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W poniedziałek 15 listopada szefowie pięciu frakcji w Parlamencie Europejskim skierowali do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen list, w którym domagają się wstrzymania akceptacji polskiego Krajowego Planu Odbudowy, KPO, do momentu, aż zostaną spełnione wszystkie instrumenty wdrożeniowe na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności. Szanowni Państwo! To wasi przedstawiciele się pod tym podpisali. A jaka jest wasza Europa? Przez estońską filię blisko 234 mld euro funduszy. Transfery z banku rosyjskiego. To jest wasza Europa. Głos zabierze pan poseł Witold Zembaczyński. Panie Marszałku! Jak słucham tej debaty w wykonaniu tej części sali, to jestem w pełni jednak przekonany, tak już ostatecznie, że najlepsza część PiS-u zginęła w katastrofie smoleńskiej. Panie pośle, przekroczył pan pewne granice, wypowiadając się w ten sposób, i chciałbym pana w tej kwestii upomnieć. Dziękuję, panie marszałku, za to upomnienie. Dzisiaj motywuje was działanie oblężonej twierdzy, ale tym wrogiem nie są instytucje europejskie, bo wystarczy być praworządnym. Wystarczy realizować wyroki europejskich trybunałów, żeby otrzymać unijne pieniądze. Dzisiaj realizujecie politykę oblężonej twierdzy, dlatego że ten wróg jest u was w środku, wewnątrz tzw. Zjednoczonej Prawicy. To są radykałowie z Solidarnej Polski. To są ekstremiści jak Antoni Macierewicz, którzy zasłaniają się wartościami narodowymi, a de facto promują antypolskie działania. Realizując wielki, okrągły antyeuropejski stół ze zwolennikami Putina w Warszawie, ostatecznie określiliście się, że patriotyzm to tylko frazes.

Wysoka Izbo! Największą bolączką polskiej polityki zagranicznej, czego pan minister jest w pełni świadom, jest to, że stała się ona zakładnikiem polityki wewnętrznej w obozie Zjednoczonej Prawicy i nie reprezentuje niestety polskiej racji stanu w ostatnich 6 latach. Ostatnio ta polityka stała się, jak powiedział pan przewodniczący Władysław Kosiniak-Kamysz, również schizofreniczna. Z jednej strony mamy Solidarną Polskę, która mówi, żeby nie płacić składek członkowskich do Unii Europejskiej - mimo że nie jesteśmy płatnikiem netto, jesteśmy póki co beneficjentem - a również sugeruje, że może będzie należało wetować wszystkie propozycje stawiane przez 26 innych państw członkowskich, czyli wyeliminować Polskę z Unii Europejskiej, de facto zrobić taki eksplozywny polexit. Z drugiej strony, czego może nie wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości są świadomi, ale pan minister Ziobro akurat jest świadom (Dzwonek), mimo negatywnego podejścia do Unii Europejskiej w rządzie Zjednoczonej Prawicy pan premier Morawiecki podpisał się pod uwspólnotowieniem i solidarnym spłacaniem długu 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, czym zrobił największy i najdłuższy krok w stronę federalizacji Europy od czasu powstania Unii Europejskiej. Jak się ma wspólny dług, to w konsekwencji płaci się wspólne podatki. Doceniam pytanie i podpisuję się pod pytaniem pana posła Rychlika, które było bardzo zasadne. Też chciałbym usłyszeć, jakie dalsze kroki na drodze federalizacji, do wspólnej polityki monetarnej i fiskalnej Unii rząd Zjednoczonej Prawicy zamierza zrobić, bo to jest bardzo istotne pytanie dla wszystkich Polaków. Rząd tej schizofrenii nie zauważa, bo żeby zacytować: Nic was nie przekona, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Bardzo dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! To pytanie sobie zadajemy. Jedni mówią, że jej nie ma, i tej wersji będą bronić posłowie z Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest mniej bolesne. Ale to nieprawda, polityka zagraniczna jest, tyle że gdziekolwiek sięgniesz, tam porażka. Krajowy Plan Odbudowy - porażka, Pakiet Mobilności - porażka, stosunki z sojusznikami - porażka, wizerunek Polski jako państwa - ostoi demokracji - porażka, Trójkąt Weimarski - porażka, dyplomacja ekonomiczna - porażka. Jest pohukiwanie, jest wymachiwanie szabelką, ale słowem najlepiej opisującym dokonania PiS w czasie ostatnich 6 lat jest słowo, sami wiecie najlepiej jakie: porażka. I jakby tego było mało, to Prawo i Sprawiedliwość wpadło na wspaniały pomysł, żeby wraz z przyjaciółmi Putina założyć de facto ambasadę moskiewską (Dzwonek) w Parlamencie Europejskim. Naprawdę nie wiem, czy nie zdajecie sobie sprawy, że to jest kierunek na zdradę. Macie reprezentować polskie interesy i tym w Parlamencie Europejskim się zająć. Zamiast dbać o pozycję międzynarodową, o naszą gospodarkę, o pieniądze dla obywateli i firm rząd Prawa i Sprawiedliwości walczy o swoje partyjne interesy. To jest niegodne urzędu, który powierzyli wam Polacy. Mieliście działać na ich rzecz, a rzuciliście się na frukty władzy. Nic gorszego Prawo i Sprawiedliwość nie mogło zrobić. Mam tylko jedno pytanie: Czy nie jest wam po prostu wstyd? Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Tracimy dziennie już milion euro w ramach kar za Izbę Dyscyplinarną, którą i tak chcecie zlikwidować. W ten sposób Izba stała się najdroższą instytucją w Polsce. Trzeba być naprawdę nieprzyzwoitym człowiekiem, by w obronie własnych obsesji narażać kraj na takie straty i jeszcze nazywać to patriotyzmem. Za każdym razem, gdy manipulujecie, siejecie dezinformację, mijacie się z prawdą w imię osłabiania jedności europejskiej, Putin otwiera szampana. I robicie to w momencie, kiedy zagrożenia na wschodzie tylko i wyłącznie rosną. Wy jesteście po prostu szkodnikami dla Polski. Dziękuję bardzo. Na tym lista posłów zapisanych do dyskusji została zamknięta. Proszę teraz o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców pana przewodniczącego Władysława Kosiniaka-Kamysza. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Widać, jak bardzo była potrzebna ta debata. Nie prowadzicie i nie prezentujecie swoich strategii w polityce zagranicznej.

To jest docenienie. Rzadko się zdarza z waszych ust, ale rozumiem, że jeżeli rządzący nie wywiązują się ze swoich obowiązków, to rolą opozycji jest przecież zaproponowanie tematu ważnego z punktu widzenia strategii polityki Polski. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia dotyczy sprostowania, bo ono musi paść z tej mównicy, obraźliwych słów i nieprawdziwych słów dotyczących roli dzisiejszej opozycji, a kiedyś partii rządzących w przystąpieniu Polski do NATO, do Unii Europejskiej. Drodzy Państwo z PiS-u! Po tej stronie sali sejmowej zasiadają ugrupowania, które walnie przyczyniły się do wstąpienia do NATO i Unii Europejskiej. Po pierwsze, wniosek do Unii Europejskiej podpisuje premier Waldemar Pawlak. Ministrem spraw zagranicznych jest Bronisław Geremek. A do Unii Europejskiej wprowadza nas rząd, w którym jest Leszek Miller i Jarosław Kalinowski. A w tym samym czasie prezydentem Rzeczypospolitej jest Aleksander Kwaśniewski.

Kiedyś zrobiliście taką wystawę w Sejmie i tam wymazaliście te postacie. Wymazać prawdę historyczną. Źle robią np. też ci z opozycji, którzy chcą zmiany nazwy ronda. To nam się też nie podoba i to mówimy jasno. Bo to jest prawda historyczna i ona jest niezależna od tego, z jakiej formacji jesteś. Bo wy macie tylko swoją historię, napisaną tylko swoimi bohaterami. Nie widzicie zupełnie innych i nie potraficie docenić tych, którzy przyłożyli rękę, a tak naprawdę położyli kamień węgielny pod Polskę w Unii Europejskiej i w NATO. I to jest nieprawda, to jest wasz wstyd, to jest wasza hańba. A ja bardzo panią proszę, pani poseł, aby pani powstrzymała emocje, jak występuje. Zastanawiam się, panie marszałku, Wysoka Izbo, czemu ich tak boli prawda. To jest naprawdę zaskakujące.

Szanowni państwo, też była mowa tutaj. Jedna z pań poseł z PiS chyba się pomyliła, bo ja mówiłem o polskiej racji stanu i przedstawiałem jej założenia.

Tak więc jeszcze raz o polskiej racji stanu. Bo nie zdementowaliście wypowiedzi ministra Ziobry, nie zaprzeczyliście dzisiaj z tej mównicy temu, co powiedział dla jednego z najbardziej opiniotwórczych dzienników światowych. I to obniża pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Polską racją stanu jest dzisiaj posiadanie dobrych sojuszników. Polską racją stanu jest współdziałanie w tematach najważniejszych. Nie proponujecie tego jako rządzący od 6 lat. Nie macie ochoty na współdziałanie w tym zakresie. Polską racją stanu jest dzisiaj załagodzenie konfliktów z naszymi sąsiadami z Unii Europejskiej, z państwami należącymi tak jak my do Unii Europejskiej, w tym z tymi z Grupy Wyszehradzkiej. Polską racją stanu jest umacnianie relacji polsko-niemieckich i gospodarczych, i politycznych. Polską racją stanu jest utrzymywanie relacji handlowych i militarnych ze Stanami Zjednoczonymi. Daliśmy wam dzisiaj szansę, przedstawiając swoje kierunki polityki zagranicznej. Jeżeli rząd abdykował, jeżeli premierem stał się w sprawach zagranicznych minister Ziobro, a ministrem spraw zagranicznych stał się Janusz Kowalski, to opozycja musi reagować na taką zamianę ról, na takie definiowanie polityki zagranicznej.

Z tego obowiązku nikt nas nie zwolni, my się z tego obowiązku nie damy wypchnąć. I nie będziecie nam odmierzać patriotyzmu, bo patriotyzm wynika nie tylko z naszego urodzenia, z naszego przywiązania, z naszej tożsamości. Wynika przede wszystkim z najważniejszej rzeczy: z prawdziwej miłości do ojczyzny. My nikomu tej prawdziwej miłości nie odmawiamy, wam również. I nie życzymy sobie, żeby ktokolwiek odmawiał jakiejkolwiek opcji politycznej czy jakiemukolwiek obywatelowi Rzeczypospolitej prawa do miłości własnej ojczyzny i działania na jej rzecz. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pana ministra Piotra Wawrzyka. Bardzo proszę, panie ministrze.

Na wstępie chciałbym podziękować panu przewodniczącemu Kosiniakowi-Kamyszowi za zakończenie wystąpienia. Jeżeli mówi pan o tym, że trzeba działać w imię polskiej racji stanu,

Tylko dwa głosy wstrzymujące się. Dzięki temu mieliśmy najlepszy w historii wynik w wyborach do najważniejszego gremium światowego decydującego o polityce bezpieczeństwa na świecie. Drugi przykład. Bardzo proszę. Jesteśmy członkami dzięki temu, że polska dyplomacja skutecznie zabiegała o te głosy. Dzięki temu możemy teraz skutecznie walczyć o prawa człowieka na Wschodzie, przede wszystkim na Białorusi, ale też w Federacji Rosyjskiej i piętnować te wszystkie antydemokratyczne działania reżimu Łukaszenki.

I to jest miara skuteczności dyplomacji. Bo polityka zagraniczna nie sprowadza się tylko do jednego dokumentu, wbrew temu, co panu się wydaje. Miarą skuteczności dyplomacji jest wybieranie, bycie wybieranym do gremiów decyzyjnych na świecie. A nam się to udaje taśmowo, można powiedzieć. To jest miara skuteczności dyplomacji i pozycji Polski na świecie. A jak to było za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego? Likwidacja ambasad, likwidacja konsulatów, bo nie było na to pieniędzy. Jak można robić skuteczną dyplomację, skoro podpisuje się kontrakt ze wschodnim partnerem tak skandaliczny, że protestuje przeciwko temu Komisja Europejska? Tak nie można, naruszacie solidarność europejską. To podpisał przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Bardzo proszę pana posła Grzegorza Matusiaka o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie pośle, zapraszam. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, druk nr 1847.

Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2021 r. wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył powyższy projekt ustawy. Dziękuję serdecznie. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń imieniu kół. Bardzo proszę panią poseł Ewę Malik z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, druki nr 1847 i 1848, po pierwszym czytaniu w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Poselski projekt ustawy przewiduje utworzenie systemu wsparcia będącego mechanizmem wsparcia publicznego dla sektora górnictwa węgla kamiennego określonym w rządowych dokumentach strategicznych. Projekt powstał z powodu konieczności stopniowego wygaszania działalności wydobywczej węgla kamiennego. Obejmuje w szczególności dopłaty z budżetu państwa do redukcji zdolności produkcyjnych oraz pokrycie kosztów wynikających z zakończenia wydobycia węgla kamiennego i likwidacji jednostek produkcyjnych. Przy czym jest to likwidacja tych jednostek, które nie są związane z bieżącą produkcją w przemyśle górniczym. Projekt przewiduje również zawieszenie, a następnie umorzenie z mocy prawa zobowiązań pieniężnych przedsiębiorstw górniczych, które są objęte systemem wsparcia, powstałych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonych i płatnika, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne, które na mocy umów zawartych przed 31 grudnia 2001 r. i obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały rozłożone na raty, lub których termin płatności został odroczony. Wczoraj podczas pierwszego czytania w komisji posłowie poparli kilka poprawek redakcyjnych do nowelizacji ustawy. Tym samym w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość rekomenduję Wysokiemu Sejmowi przyjęcie omawianego projektu. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Krzysztofa Gadowskiego z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiaj rzeczywiście debatujemy nad bardzo ważną ustawą, jeszcze raz podkreślę, bardzo ważną ustawą. Co prawda ona idzie w kierunku realizacji umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, która została podpisana 28 maja 2021 r. między stroną społeczną, stroną rządową, samorządowcami i przede wszystkim związkami zawodowymi. Rozpoczynamy kolejny etap likwidacji kopalń, który potrwa aż do zakończenia eksploatacji węgla kamiennego, zgodnie z harmonogramem, który został zawarty w tej tzw. umowie społecznej. To ważny i poważny w skutkach proces dotyczący transformacji górnictwa węgla kamiennego i, jak wspomniałem, transformacji województwa śląskiego. Przypomnę, czego on dotyczy. Chodzi o likwidację ok. 80 tys. miejsc pracy w kopalniach i 410 tys. miejsc pracy w firmach okołogórniczych. Taki proces powinien być przygotowany i przeprowadzony przez rząd. Powinien zostać zaopiniowany w pełnej procedurze, jako ustawa rządowa. Pierwsze czytanie powinno odbyć się tu, w Sejmie, a nie w zakamarkach sekretariatu Sejmu. W tym procesie powinny uczestniczyć strony tej umowy. Szanujmy te podmioty, szanujmy górników, związkowców, szanujmy tych, którzy miesiącami pracowali nad tym projektem ustawy. A co my mamy?

Wrzucony, procedowany bardzo szybko, kolanem dopinany.

Chcemy tego wsparcia udzielić, ale chcemy w sposób partnerski do tego typu ustaw podchodzić. Nikt wczoraj w komisji nie powiedział nam, w jakim zakresie ta pomoc będzie dotyczyła jednego, drugiego, trzeciego podmiotu. Jak ten proces restrukturyzacji dzisiaj się ma? Nie było żadnego prezesa spółki węglowej, która będzie korzystać z dobrodziejstwa tego projektu ustawy.

Dotyczy to składek ZUS. Zobowiązania dotyczą przede wszystkim Polskiej Grupy Górniczej. To również dotyczy Polskiej Grupy Górniczej, spółki górniczej, którą na sztandarach niosło Prawo i Sprawiedliwość. Mówimy o kosztach.

Proces notyfikacji. Nowy system wsparcia wymaga notyfikacji i akceptacji Komisji Europejskiej.

Dziś nie wiemy, czy tych środków wystarczy, czy jest ich za mało, czy w przyszłym roku będzie potrzeba więcej. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Koalicji Obywatelskiej, zdając sobie sprawę z procesu transformacji i tej górniczej, i tej energetycznej, a także widząc, w jakiej sytuacji rząd Prawa i Sprawiedliwości pozostawia spółki węglowe, podejmie się prac nad tym projektem ustawy. Będzie popierał proces wsparcia transformacji energetycznej, a zarazem górniczej Polski. Dziękuję bardzo. Natomiast chciałbym, panie marszałku, złożyć jedną poprawkę.

Bardzo proszę, pan poseł Maciej Konieczny, klub parlamentarny Lewica. Wysoka Izbo!

Przypomnijmy, że chodzi o projekt absolutnie kluczowy dla przyszłości polskiej energetyki, przyszłości Śląska. Chodzi o kilkaset tysięcy miejsc pracy, kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy w górnictwie i kilkaset tysięcy miejsc pracy w przemysłach powiązanych. Chodzi w końcu o implementację umowy społecznej, czyli zobowiązania, które wziął na siebie rząd Prawa i Sprawiedliwości po rozmowach ze związkowcami. Ten sposób procedowania jest zwyczajnie nieodpowiedzialny, biorąc pod uwagę skalę i wagę spraw, o których rozmawiamy. Jest oczywiste, że plan wygaszania polskiego górnictwa węgla kamiennego jest czymś, za co odpowiada rząd, i to rząd powinien proponować konkretne rozwiązania w normalnym, przewidzianym dla tego trybie. No, ale dowiadujemy się, że sytuacja jest nadzwyczajna.

Wydaje się, że nie ma nic rzadszego w tym Sejmie niż normalny proces ustawodawczy. Wygląda to na kompletny chaos.

To coś wyjątkowego, coś ponadstandardowego, coś, czego faktycznie potrzebujemy w związku z opóźnieniami, jeżeli chodzi o polską transformację energetyczną, w związku ze szczególną sytuacją Polski, w której energetyka w tak dużym stopniu opiera się na węglu. Potrzebujemy wyjątkowego traktowania i potrzebujemy zgody Komisji Europejskiej. Potrzebujemy tego, żeby ta transformacja była sprawiedliwa i przeprowadzana z poszanowaniem zdania mieszkańców i mieszkanek regionów pogórniczych. To jest kluczowe.

Serio, chojrakowanie ministra Ziobry naprawdę jest dla was ważniejsze niż los polskich górników, niż los Śląska, niż los polskiej energetyki? Bo na to wygląda. Tu nie chodzi zresztą tylko o notyfikację umowy społecznej, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, a w każdym razie lewica zdaje sobie sprawę, bo z wami to nie wiadomo, z tego, że transformacja energetyczna to jest ogromny proces i wygaszanie wydobycia węgla kamiennego to jest tylko niewielka jego część. Potrzebujemy wsparcia dla firm okołogórniczych na przekwalifikowanie produkcji, potrzebujemy inwestycji w nowy, zielony przemysł, potrzebujemy sensownego planu zagospodarowania terenów pogórniczych i potrzebujemy nowych, stabilnych źródeł energii. Naprawdę jest co robić i potrzebujemy na to europejskich środków. Tymczasem co robi polski rząd? Na własne życzenie wyrzuca do kosza środki z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Lekką ręką płaci codziennie wielomilionowe kary za swoją nieudolność. W końcu poważnie ryzykuje nawet utratą podstawowych strukturalnych funduszy z Unii Europejskiej. Dlaczego? Bo pan Ziobro ma taką fantazję, żeby ręcznie sobie sterować wymiarem sprawiedliwości. To jest najpoważniejsze oskarżenie, bo mamy wyjątkową sytuację. Potrzebujemy notyfikacji Komisji Europejskiej, żeby móc w sposób planowy, kontrolowany i odpowiedzialny odejść od węgla w naszej energetyce, żeby nie było powtórki z niekontrolowanego zamykania kopalń, żeby nie było powtórki z lat 90. Do tego potrzebujemy funduszy, potrzebujemy zgody, potrzebujemy wsparcia naszych europejskich partnerów.

Tak, to jest o węglu. Dokładnie to jest o węglu. Tak, przyszłość Śląska zależy od tego, czy Komisja Europejska zgodzi się na dopłatę do wydobycia węgla. Tak, to jest o węglu. Ale dla was, jak widać, przyszłość Śląska i losy pracowników (Dzwonek) górnictwa mają mniejsze znaczenie niż wasze ideologiczne wojenki. Jako lewica zagłosujemy za tą ustawą, z pełną świadomością, że to jest wasza odpowiedzialność.

My za tym zagłosujemy, bo wiemy, że od tego zależy bezpieczeństwo miejsc pracy na Śląsku, ale to jest wasza odpowiedzialność. Mam bardzo poważne wątpliwości, czy pracując w tym chaotycznym trybie jesteście w stanie w sposób odpowiedzialny zadbać o bezpieczeństwo rodzin z regionów górniczych. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę pana posła Władysława Teofila Bartoszewskiego. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mamy węgiel, który nam starczy na 200 lat. Nie zamkniemy żadnej kopalni. Żaden górnik nie będzie bez pracy. A potem przychodzi Europejski Zielony Ład i z łapanki organizujecie komisję.

Zbiera się grupka posłów - bez żadnych konsultacji, bez porozumienia społecznego, bez rozmów z górnikami. To to nie jest mała suma. Co więcej to wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej i aprobaty, ponieważ są to środki, które będą uważane za pomoc publiczną. To jest skandaliczny sposób procedowania nad tak ważną ustawą, istotną dla setek tysięcy mieszkańców Śląska, których wyraźnie sobie lekceważycie.

Jeżeli tego artykułu nie poprawicie, to sami się wpakujecie w potworne kłopoty.

To jest rola rządu, to powinien robić rząd, a nie grupa posłów, która tego specjalnie dobrze nie przemyślała.

Dziękuję. Pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja.

Wysoka Izbo! To jest ustawa likwidująca górnictwo węgla kamiennego w Polsce i to jest radykalne i jaskrawe złamanie przyrzeczeń PiS-u sprzed wyborów, z kampanii wyborczej, z pierwszych lat rządów.

O to oskarżam związki zawodowe ze Śląska. Podpisaliście ją i to powiedział Kolorz otwarcie, publicznie, wyszedł na konferencję prasową i powiedział: tak, proszę państwa, zamykamy rozdział pt. górnictwo węgla kamiennego w Polsce. Zrobiliście to razem, PiS ze związkami zawodowymi ze Śląska to zrobił. Taka jest prawda. Kapitulacja całkowita wobec Brukseli. I teraz chcecie to osładzać, tę całą kompromitację i tę kapitulację, tą ustawą. My się nie zgadzamy. Żądamy od rządu czegoś przeciwnego, żądamy wypowiedzenia pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej natychmiast, teraz, podczas najbliższego szczytu Rady Europejskiej. To jest polska racja stanu. Krzyczycie, że Tusk podpisał zobowiązania w sprawie emisji, krzyczycie, że Tusk się zgodził - to zróbcie coś z tym wreszcie. Przestańcie kontynuować politykę Tuska, która dzisiaj owocuje nie tylko likwidacją naszego wydobycia, problemami energetyki, ale również likwidacją naszego przemysłu energochłonnego, bo do tego to prowadzi, i drożyzną, jeśli chodzi o cenę energii. Unia Europejska i kontynuacja polityki klimatycznej Unii Europejskiej dzisiaj równa się: wysokie ceny prądu, likwidacja górnictwa, likwidacja przemysłu energochłonnego. I albo powiecie temu: stop, albo jesteście takimi samymi zdrajcami sprawy polskiej jak Tusk. Dokładnie tak samo. Albo tak, albo tak. Szanowni Państwo! To dziewięć poprawek, które odsyłają tę ustawę do kosza.

Pani poseł Paulina Hennig-Kloska, Polska 2050. Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! ale to potężny proces, który wymaga również szczerej i otwartej dyskusji nad wieloma aspektami tej transformacji: nad planem wsparcia dla ludzi odchodzących z górnictwa, nad planem wsparcia dla regionów, dla których górnictwo wciąż jest ważnym elementem gospodarki i umożliwia finansowanie życia społecznego. To także dyskusja o planie i naprawie szkód środowiskowych, które pozostaną do naprawienia właśnie po działalności górniczej. Niestety dziś chcecie przyjąć ustawę w ogóle bez dyskusji, bo proces legislacyjny, który towarzyszy tej ustawie, najlepiej obrazuje wasze podejście do transformacji energetycznej. Panie pośle, pan chce rozmawiać, ale myśmy nie dostali od rządu ani planu. Ale proszę mi nie przeszkadzać. Nie dostaliśmy od rządu ani planu wsparcia dla ludzi odchodzących z górnictwa, ani planu wsparcia dla regionów, ani planu naprawy szkód środowiskowych. W tej ustawie jest tylko jedna rzecz: 28 mld zł, które chcecie wydrukować z długu pozabudżetowego poprzez obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa poza kontrolą parlamentu na transformację energetyczną. Nie wiemy kompletnie, co chcecie za te pieniądze zrobić, i nikt nam tego na posiedzeniu komisji nie potrafił powiedzieć. A proces legislacyjny jest w ogóle jakimś skandalem.

Nie da się. Oczywiście podlega jeszcze dyskusji to, że nie mamy prenotyfikacji Komisji Europejskiej, i pytanie, czy Komisja w ogóle ten styl przyjmie. Ale jest też pytanie kluczowe: Jakie są prawdziwe intencje wnioskodawców? Bo mam ogromne wątpliwości, dlaczego ta ustawa w takim trybie na koniec roku musi być przyjęta. Jeżeli my nie mamy tych podstawowych informacji, to również nie mają tej informacji osoby zatrudnione w górnictwie.

Zamykam listę zgłoszonych do pytań.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Oczywiście są wielkie spółki państwowe, które otrzymują wsparcie, i to wsparcie jest kierowane szerokim strumieniem, natomiast są też prywatne spółki górnicze, jak np. spółka w Czechowicach, która nie ogląda się na budżet państwa. I pytanie jest takie: Czy również do tych firm, które do tej pory nie korzystały z państwowego wsparcia, do górników, którzy brali sprawy w swoje ręce, rząd będzie kierował to wsparcie związane z restrukturyzacją, związane z procesem odchodzenia, związane z procesem zamykania kopalń?

Czy będzie to wsparcie dla takich spółek i pracowników?

Jeszcze jedno pytanie, o którym w zasadzie zapomniałam w trakcie swojego wystąpienia: Co z regionami, w których wydobywa się węgiel brunatny? Jeszcze o węglu kamiennym w rządzie się myśli, ale są regiony, gdzie wydobywa się węgiel brunatny, gdzie problemy są dosłownie takie same, gdzie są problemy społeczne związane z odchodzeniem od węgla.

One też tam występują. I wydaje się, że te regiony zostały całkowicie pozbawione jakiegokolwiek wsparcia ze strony rządu, m.in. wschodnia Wielkopolska, z której pochodzę. Pytanie kluczowe, panie ministrze: Kiedy porozmawiamy o węglu brunatnym? Wysoka Izbo! Pani mówi, że pani niewiele wie. Warto by było pamiętać, że od maja toczy się na ten temat dyskusja. To po pierwsze. Po drugie, dobrze by było zapoznać się z uzasadnieniem, pani poseł, tej ustawy. Ta ustawa rozpoczyna bardzo trudny proces, szczególnie dla ludzi na Śląsku, ludzi związanym z górnictwem. Ale chcę powiedzieć, że ta ustawa również dotknie region warmińsko-mazurski, ponieważ są firmy, które wykonują pewne usługi na rzecz polskiego górnictwa.

Chciałbym zapytać, na jakim etapie w tej chwili są rozmowy z Komisją Europejską odnośnie do notyfikacji. Jest to pomoc publiczna i ta notyfikacja musi być. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Polska stoi na węglu. Na węglu, którego ceny w ostatnim roku osiągnęły wręcz gigantyczny poziom. Nasz kraj przyjął proputinowską politykę polegającą na sprzedaży naszych uprawnień do emisji CO2. Za te pieniądze kupujemy węgiel z Rosji. Rosyjskim węglem opalamy nasze elektrociepłownie i elektrownie, ale że już nie posiadamy praw do emisji, bo nimi zapłaciliśmy Putinowi, polski konsument ma podnoszone ceny prądu. Jednocześnie ten sam konsument, czyli podatnik, ma dokładać miliardy złotych do wygaszania polskiego przemysłu górniczego i, jak czytamy w ustawie, do umorzeń zaległych opłat składek ubezpieczeniowych oraz innych zaległości. Taka sytuacja rzeczywiście wymaga rzetelnej i szczerej rozmowy, a tej rozmowy nie gwarantuje projekt, który jako posłowie otrzymaliśmy wczoraj. Poziom rządowego zarządzania górnictwem to rzeczywiście, tak jak było mówione na tej sali, prawie Legia Warszawa. Pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W czasie komuny Polacy kupowali na kartki, a w czasie rządów Platformy i PSL-u kupowali na zeszyt. Dzisiejsza polityka klimatyczna Unii Europejskiej chce dokładnie doprowadzić do tego samego, aby Polacy znowu kupowali na kartki i na zeszyt. Dlatego bronię, szanowni państwo, polskiego węgla, bronię naszej niezależności i suwerenności energetycznej. I dzisiaj największym dla nas wyzwaniem jest to, aby ten absolutnie spekulacyjny, niezdrowy system unijnego handlu emisjami znieść.

To są pieniądze, które powinny zostać w polskiej gospodarce. Jestem przekonany, że kampania w roku 2022 to rozstrzygnie. Pan poseł Mariusz Gosek, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Nie ma zgody na spekulacyjny system handlu emisjami CO2. Nie ma zgody na likwidację polskiego węgla, dlatego że polski węgiel to 70% rynku energetycznego Polski.

W samym górnictwie pracuje 80 tys. osób, dookoła przemysłu górniczego pracuje kolejnych 400 tys. osób. Do tego jako cała klasa polityczna powinniśmy stanąć równo przeciwko eurokratom, przeciwko tym, którzy próbują spowodować… Nie ma zgody na likwidację polskiego górnictwa (Dzwonek), przemysłu cementowego i wapienniczego. Wysoka Izbo! Pierwsze: robić to państwowo, ze związkami zawodowymi i dopłacać do tego potworne sumy. Możliwość druga: zamknąć te kopalnie na polecenie Unii Europejskiej.

Dziękuję. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! To ustawa, która właściwie reguluje sytuację spółek górniczych. Przypomnę, że Platforma rządziła 8 lat i zakończyło się to strzelaniem do górników pod Jastrzębską Spółką Węglową.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Co z nimi?

Czy będzie to uzależnione od systemu właścicielskiego?

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Odwołujemy się do umowy społecznej, która została przygotowana i w maju podpisana.

Strona społeczna przygotowała projekt ustawy.

Kiedy zostanie powołany Fundusz Transformacji Śląska?

Wysoka Izbo! Rozmawiamy o wielkich rzeczach, w tle transformacja energetyczna, wielkie opłaty emisyjne.

Jeżeli doszło do wypadku śmiertelnego, to mówiło się, że górnik poległ. Ale to historia. Dzisiaj chciałem spytać, czy rząd ma świadomość - a kontakty mam cały czas - że bardzo wielu górników czuje się oszukanych przez rząd.

Pani poseł Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Chciałam zapytać o skutki finansowe dla budżetu państwa z tytułu dopłat do redukcji zdolności produkcyjnej dla przedsiębiorstw górniczych.

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przez najbliższą dekadę wsparcie górnictwa ma nas kosztować niemal 30 mld zł. Obecnie w Polsce pracuje ok. 80 tys. górników.

Panie ministrze, pytanie brzmi: Jaka część z tych 30 mld zł ma trafić bezpośrednio do tych rodzin? Co chcecie zrobić, żeby te pieniądze realnie pomogły górnikom, a nie trafiły do kieszeni zarządów Polskiej Grupy Górniczej, Tauronu Wydobycie czy jakiejś innej spółki obsadzonej przez waszych kolesi. Odejście od węgla musi być naszym wspólnym celem, ale transformacja gospodarki będzie udana tylko wtedy, gdy będzie naprawdę sprawiedliwa społecznie, czyli nikogo nie zostawi się na lodzie. Pani poseł Ewa Malik, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo! Panie Ministrze! Ten projekt jest objęty zakresem regulacji Unii Europejskiej, dlatego chciałabym zapytać, czy tę nowelizację już pan omówił z przedstawicielami Unii Europejskiej, czy na pewno nie budzi ona z ich strony żadnych zastrzeżeń i czy w ogóle jest konieczna notyfikacja tego projektu w Komisji.

Jeżeli tak, to proszę potwierdzić te moje wątpliwości. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Panie Marszałku - Wysoki Sejmie! Sprawiedliwa transformacja górnictwa musi również obejmować górnictwo węgla brunatnego. Każdorazowo my, parlamentarzyści z okręgu nr 37, pytamy o to górnictwo węgla brunatnego w kontekście Turku, Konina, ale także innych miejscowości. 17 września w czasie debaty pan minister Soboń, odpowiadając na moje pytanie, powiedział w ten sposób: 1 września rozpoczęliśmy ze stroną społeczną rozmowy w tym zakresie. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy zostaną one zakończone wypracowaniem wspólnego porozumienia i że będziemy mogli jasno powiedzieć, że dokładnie te same rozwiązania osłonowe będą dotyczyły również górników węgla brunatnego. Dziękuję.

Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Odpowiemy pisemnie po debacie. Przede wszystkim o czym mówimy? Mówimy o procesie restrukturyzacji czy likwidacji kopalń? Wchodzimy w proces likwidacji kopalń i chciałbym, żeby to było jasno określone. Kwestia zasadnicza, jeżeli chodzi o tę ustawę, to kwestia ustanowienia płynności finansowej tych firm, o których mówimy, które są przedmiotem tej ustawy, gdyż brak płynności spowoduje koniec górnictwa w sposób nieprzewidywalny, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Jeśli chodzi o nasze działania, które mają wpływ na szybkość procedowania nad tą ustawą, to jest kwestia, nie ukrywam, moich rozmów z 2 grudnia w Komisji Europejskiej. Powiem tak - i tu, przepraszam, może tak troszeczkę od końca odpowiem pani poseł - mianowicie ustawa wpisuje się w mechanizm zarówno naszego wniosku prenotyfikacyjnego, jak i tego, który złożymy w połowie stycznia, czyli notyfikacyjnego. Pan poseł Suchoń pytał o Silesię, firmę, która jest firmą prywatną, czy będzie objęta tymi dotacjami.

Pozwolę sobie, odpowiadając pani poseł... nie widzę pani poseł.

Dobrze, pozwolę sobie kontynuować. Okej.

Ktoś z państwa o tym wspominał, z Lewicy, jeżeli się nie mylę. Odniosę się do kwestii Śląska.

Ale do tego jeszcze wrócę pod koniec swojego wystąpienia. Bardzo dziękuję za to pytanie. Dlatego że w Komisji Europejskiej pokazano mi - jeżeli dobrze pamiętam - jakąś teczkę czy segregator z artykułami z polskich mediów, czy na bazie polskich mediów, przetłumaczonymi na język angielski dla moich rozmówców - adwersarzy z drugiej strony.

Nie wiem, jak to określić, w każdym razie nie są to informacje ani ode mnie, ani z Ministerstwa Aktywów Państwowych, ani tym bardziej z Komisji Europejskiej. Natomiast przewidują one jakieś rozwiązania w przyszłości. W razie pojawienia się takich artykułów, takich informacji w jakichkolwiek mediach bardzo proszę o kontakt z Ministerstwem Aktywów Państwowych, z moją skromną osobą. Będziemy bezwzględnie i natychmiast reagowali na takie informacje, zwłaszcza bezwzględnie, dlatego że to jest naruszenie polskiej racji stanu i w podległym mi resorcie takie rzeczy nie będą tolerowane.

Albo odpowiemy pisemnie, albo zaprosimy do resortu i przedstawimy wszystkie dane. Tak że jak państwo sobie tutaj życzycie, jesteśmy do dyspozycji, transparentni i otwarci, bo w przypadku pracy nad węglem inne rozwiązanie nie wchodzi w ogóle w rachubę.

To nie jest pomysł na pomoc socjalną. To jest ustawa, która ma po prostu utrzymać, uratować miejsca pracy. Taki jest cel, takie założenie. Tempo wynika z kontekstu sytuacyjnego, a nie czyjegoś lenistwa, zaniechania czy zaniedbania. Wszyscy, którzy siedzą w węglu, to rozumieją i podzielają, jak się wydaje, moje zdanie. Pani poseł Malik już odpowiedziałem.

A po drugie, chciałem podziękować za merytoryczną debatę w tym punkcie i za to, że mogliśmy dojść do konsensusu, jak się wydaje, ponad podziałami politycznymi. Serdecznie za to dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję.

W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń. Nie widzę takich zgłoszeń. Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem za zamkniętą. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Prawdziwe Boże Narodzenie, święto, w które wspominamy narodziny naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest w Polsce szczególnym dniem. Dzisiejsze Boże Narodzenie będące ważną pamiątką wynikającą z wydarzeń katolickiego roku obrzędowego różni się nieco w szczegółach od święta, jakie obchodzili nasi przodkowie.

Kiedyś z bliskimi dzielono się chlebem, zanim rodzina usiadła do wigilijnego stołu, a dziś służy do tego opłatek. To nie ma znaczenia. Dla nas, chrześcijan, katolików ważne jest to, że czcimy dzień narodzin Boga, który w ludzkiej postaci zszedł między nas, żeby dać nam zbawienie. Od ponad tysiąca lat, od chwili, gdy przyjęliśmy chrzest w 966 r., my, Polacy jesteśmy jednoznacznie osadzeni w kulturze zachodniego chrześcijaństwa. Wiele razy niektórzy, różne siły próbowały nam udowodnić, że nie należymy do Zachodu. To typowe dla narodów z pogranicza kultur. Na Wschód od nas były ludy, które przyjęły chrzest w Bizancjum, co stawiało je w zupełnie innym kontekście historycznym i mentalnym. Tam do dziś inaczej pojmuje się sprawy zasadnicze. Jakkolwiek, będąc częścią Zachodu, mimo wyraźnego obciążenia w jego kierunku, w pewnych, no cóż, niemal eschatologicznych sprawach różnimy się od jego mieszkańców zasadniczo. Ta różnica to przede wszystkim stosunek do religii, wiary, a także do tego, co oczywiste - tradycji. Dla większości Polaków, jak wspomniałem na początku, Boże Narodzenie to święto, które uświęcamy tymi samymi od stuleci obrzędami, tymi samymi pieśniami, miłością i wspólnym spędzeniem czasu.

Tak, to oczywiste. Jednak zrozumieć to, że Europa, ściśle mówiąc Komisja Europejska, w opublikowanym na początku grudnia tego roku przewodniku komunikacji inkluzyjnej ogłosiła, iż sformułowanie „Boże Narodzenie” może być dla pewnych osób obraźliwe i nie powinno się go używać. Jak to rozumieć? Czyżby ten Zachód, a w tym państwa, w których chrześcijaństwo ma dłuższą tradycję niż w Polsce, wstydziły się świętowania Bożego Narodzenia? Czy tzw. elity nie wiedzą, co to jest cywilizacja łacińska? Być może wystarczy im Christmas, w którym biskupa Mitry Mikołaja zastępuje ubrany na czerwono pajac wymyślony przez ekspertów PR firmy od napojów? W przedświątecznym rozgardiaszu i później, przy świątecznym stole między bliskimi my, tu w Polsce nie przyjmujemy złych przykładów płynących z budynków urzędów europejskich. Świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Aleksander Mrówczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dla mnie był to czas nauki, zdobywania doświadczenia parlamentarnego, poznawania arkanów polityki. Z samorządowca zostałem posłem. To ogromna różnica, ale dzięki pani poseł Jolancie Szczypińskiej nigdy nie zapomniałem, że najważniejszy jest człowiek, że najważniejsza jest pomoc słabszym, niezaradnym, tym, którzy nie potrafią przebić się przez mury urzędniczej biurokracji i braku zrozumienia. Jolanta Szczypińska odchodziła z wielką godnością i spokojem. Cierpiała w ciszy. Choroba, z którą walczyła wiele lat, niestety ją pokonała i zdecydowanie za szybko zabrała. Mogła jeszcze bardzo wiele zrobić dla Polski, dla Pomorza, dla Słupska. Przez wiele lat zabiegała o drogę ekspresową S6, która dzisiaj jest zbudowana, która połączy Szczecin przez Słupsk z Trójmiastem. I tutaj, z tej mównicy przede wszystkim pragnę pani poseł Jolancie Szczypińskiej podziękować, wszyscy winniśmy jej podziękować za wielki wkład w to dobre dzieło.

Byliśmy tam z panią poseł. Wieczorem tego dnia pojawiła się gorączka, następnego dnia zabrakło pani poseł tutaj, na sali obrad. Mija trzecia rocznica jej śmierci. Niestety nie mogłem uczestniczyć w uroczystościach rocznicowych w Słupsku.

W moim imieniu na grobie zmarłej wieniec złożył jej przyjaciel, wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk. Spoczywaj w pokoju. Amen.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pod koniec listopada pan premier Morawiecki obiecał, że rząd wprowadzi rozwiązania, które spowodują obniżenie ceny paliwa na stacjach benzynowych. Mówił m.in., że - tu cytuję - wprowadzamy obniżkę cen paliw już od 20 grudnia na 5 miesięcy, wdrażamy obniżkę cen paliw poprzez to, na co państwo ma wpływ: wysokość akcyzy zostanie obniżona do poziomu minimalnego w Unii Europejskiej, po drugie, od stycznia 2022 r. do 31 maja, też na 5 miesięcy, paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej, a także zwolnimy z opłaty emisyjnej, również na 5 miesięcy. Dokładnie tydzień temu większość parlamentarna złożona z posłów Prawa i Sprawiedliwości odrzuciła podczas prac w komisji projekt zawieszający pobór opłaty emisyjnej, czyli tej opłaty, której zawieszenie obiecał premier Morawiecki. Projekt ten został złożony przez Polskę 2050. Jest on częścią konkretnego pakietu przeciw drożyźnie, który nazwany został w mediach piątką Hołowni. Choć trzeba wyraźnie powiedzieć, że rozwiązania proponowane przez rząd są zbyt płytkie i zbyt wąskie, to w zakresie opłaty emisyjnej zostały de facto zapożyczone z programu Szymona Hołowni. Posłowie PiS odrzucili ten projekt, pomimo że realizuje on obietnicę premiera, a do Sejmu nie wpłynął żaden inny projekt w tej sprawie. Warto też zauważyć, iż jest to przedostatnie posiedzenie Sejmu w tym roku.

W związku z powyższym oczekuję od pana premiera Morawieckiego wyjaśnień, z jakich powód projekt ustawy Polski 2050, realizujący obietnicę premiera, został odrzucony. I mam pytanie: Czy to oznacza, że pan premier Morawiecki znowu okłamał obywateli i opłata emisyjna pomimo złożonej obietnicy nie zostanie zawieszona? Teraz pani poseł Monika Falej, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: Jesteśmy dumni z tego, że ludzie przyjeżdżają do Polski i widzą: o, bardzo łatwo jest się dostać do budynku, wszystko jest dostosowane, jaka ładna architektura, a jaka przyjazna. Idąc, czują, że jakoś tak jest inaczej, bardziej otwarcie, bo nie ma schodów, bo podejście jest łagodne, jest dobrze obliczone, bo nie ma utrudnień - mówi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent nie dostrzega, jak widać, potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Według niego wszystkie problemy osób z ograniczeniami ruchowymi zostały już rozwiązane. Dlatego, korzystając z funduszu europejskich, wprowadził program „Dostępność+” Jest to krok w dobrą stronę. Dostrzeżone są w nim problemy, z jakimi na co dzień boryka się milion Polek i Polaków.

Program zakłada realizację 900 inwestycji poprawiających dostępność. Sama Iława zgłosiła zapotrzebowanie na realizację 240 takich właśnie inwestycji, a to tylko jedno z wielu miast. Takich gmin i miejscowości jest więcej.

Dziś włodarze miast z mojego regionu piszą do prezesa Rady Ministrów apele o zwiększenie nakładów w ramach programu „Dostępność+” w obszarze architektura. Problem jest naglący, dlatego dołączam dziś do tego apelu i wzywam polski rząd do natychmiastowych działań.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Jacek Kurzępa, Prawo i Sprawiedliwość.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Koleżanki i Koledzy Parlamentarzyści!

Zatem dla was i o was będę mówił, ale również i o samym sobie.

Oświadczenia często odnoszą się do spraw związanych z tematyką tożsamości lokalnej, wzmacniania patriotyzmu i dziedzictwa przodków.

Nazwiska posłów, które wymieniłem, moglibyśmy przeplatać również wokół tematu. Szeroka tematyka znajduje odzwierciedlenie również, Andrzeju Kryj, w twoich wystąpieniach. Bardzo dziękuję i serdecznie gratuluję tych wystąpień. Musimy przez 5 minut względnie sensownie i logicznie mówić w imieniu naszych społeczności lokalnych bądź za nie.

Druga kwestia. Musicie być w swoim terenie, trzymać rękę na pulsie, wiedzieć, co się dzieje, co jest ważne. To jest niebywale ważne nie tylko dla nas. To jest ważniejsze dla tych, o których mówimy. Zarówno wy, jak i ja często potem spotykamy się z życzliwością tych, o których mówiliśmy. Ostatnia rzecz. Musimy pokonać własne słabości, własne niepokoje. Mówienie w tej chwili tak jak ja to czynię, stary wyga sejmowy z nieco swobodniejszą naturą, nie przychodzi samo z siebie. To trzeba przetrenować, przećwiczyć. Pozwólcie, że zwrócę się również do pana marszałka. Panie marszałku, bardzo dziękuję za waszą, marszałków Sejmu, cierpliwość, bo przecież po wielogodzinnych obradach bardzo często ten ostatni punkt jest trudny również dla was. Wielokrotnie pan marszałek mówi: przekażcie do protokołu tekst pisany. Za tę cierpliwość, panie marszałku, za wyrozumiałość (Dzwonek) również dla nadmiaru naszej gorliwości dziękuję.

Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku!

Uroczystości, których gospodarzem oraz inicjatorem był burmistrz Marek Długozima, były zwieńczeniem ogłoszonego przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego w jego 120. rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci.

Pomnik stanął na skwerze w pobliżu Międzynarodowego Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, do której bł. kard. Stefan Wyszyński wielokrotnie modlił się przy jej grobie i zawierzał jej losy swoje oraz kraju, a w swoich kazaniach i przemówieniach wielokrotnie nawiązywał do jej życia pełnego dzieł miłosierdzia. Obok pomnika znajduje się również monument innego wybitnego Polaka, papieża i świętego Kościoła katolickiego Jana Pawła II, osobiście wielkiego przyjaciela kard. Wyszyńskiego. Losy kardynała są związane z wieloma miejscami na mapie naszej ojczyzny. Urodził się na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Uczył się w Warszawie i Łomży. We Włocławku przyjął święcenia kapłańskie. Na Jasnej Górze zaś odprawił mszę prymicyjną. W latach późniejszych studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i obronił doktorat z Prawa kanonicznego. Również Trzebnica znalazła się na szlaku jego licznych podróży. Była jednym z pierwszych miejsc odwiedzonych przez Stefana Wyszyńskiego po objęciu urzędu prymasa Polski. Trzebnica to 13-tysięczne miasto, które znajduje się w pobliżu Wrocławia i wyrasta na enklawę patriotyzmu, która kształtuje w najmłodszym pokoleniu świadomość historyczną i tożsamość narodową, o czym świadczą liczne wydarzenia oraz inicjatywy, które w ostatnich latach są realizowane i do których z pewnością należy odsłonięcie pomnika błogosławionego kardynała. Na pomniku bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w Trzebnicy burmistrz Marek Długozima umieścił cytat, który warto tutaj przytoczyć: Tutaj, na ziemi polskiej, my jesteśmy gospodarzami. Do nas należy decydować o takim czy innym kierunku naszego życia i bytowania. Od tego bowiem zależy suwerenność narodu.

Stefan Wyszyński to wielka postać, wspaniały kapłan i człowiek, przez wielu nazywany duchownym przywódcą narodu. Odegrał bardzo ważną rolę we współczesnej historii Polski, a szczególnie w czasie trwania komunizmu. We wszystkim, co robił, oddany był ojczyźnie, a jej losy zawierzał zawsze Maryi. Twierdził, że bez względu na przeszkody trzeba podejmować wysiłek tworzenia lepszej przyszłości. Podkreślał ogromną rolę naszej wspólnoty narodowej oraz miejsce wiary i Kościoła w tej wspólnocie. Jego wielkie zatroskanie o suwerenność narodu stało się zadaniem, które pozostawił nam w duchowym testamencie. Odsłonięcie pomnika w centrum miasta Trzebnica to niezwykle cenna inicjatywa, za którą bardzo dziękuję. Uwrażliwia nas na kwestie wiary, wartości, a przede wszystkim polskości, którą kard. Wyszyński rozumiał jako dążenie do utrzymania suwerenności. Wierzę, że jego duchowy testament ma godnych i wartościowych spadkobierców. Pan poseł Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

Dziś właśnie w Ćmielowie odbyły się uroczystości pogrzebowe tego wybitnego artysty. Obowiązki poselskie, trwające posiedzenie Sejmu uniemożliwiły mi osobisty w nich udział. Chciałbym właśnie w formie oświadczenia poselskiego wyrazić hołd dla tego wybitnego mieszkańca powiatu ostrowieckiego i wielkiego artysty. Ukończył liceum plastyczne w Lublinie, a następnie w roku 1977 - Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Po studiach wrócił do swej rodzinnej miejscowości, gdzie tworzył. Jak sam mówił, to właśnie w rodzinnej Woli Grójeckiej znajdował inspiracje. Wracając do swego rodzinnego środowiska, wracasz do swego podglebia kulturowego i to ci daje pewne inspiracje, siły do działania, pewne skojarzenia - powiedział. Gustaw Hadyna był autorem monumentalnych rzeźb o tematyce patriotycznej, lecz również małych form przestrzennych, pomników, popiersi, medali. Zaprojektował m.in. wspólnie z Jerzym Fronczykiem Pomnik-Mauzoleum Męczeństwa Wsi Polskiej w Michniowie oraz pomnik poświęcony „Jędrusiom” w Bogorii. Zrealizował pomnik Batalionów Chłopskich na rynku w Opatowie oraz na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, a także pomniki Janusza Korczaka w Kielcach, Zawiszy Czarnego w Garbowie, Piotra Ściegiennego w Lublinie, jak również triadę Temidy na gmachu sądu w Piotrkowie Trybunalskim. Gustaw Hadyna wykonał także cykl rzeźbionych portretów wybitnych Polaków: Tadeusza Kościuszki, Romualda Traugutta, Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa, Juliusza Słowackiego, Jana Kochanowskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Mikołaja Reja, Władysława Hasiora czy Władysława Orkana. Rzeźby Gustawa Hadyny zdobią także dziedziniec X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

W listopadzie 2019 r. w uznaniu zasług dla polskiej kultury został odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, który nadał mu minister kultury i dziedzictwa narodowego wicepremier Piotr Gliński. Był wspaniałym gawędziarzem. Będzie nam go bardzo brakować. Guciu, spoczywaj w pokoju. Pani poseł Anna Pieczarka, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pragnę serdecznie podziękować Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Aktywów Państwowych za wspieranie polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych i polskiej myśli technicznej. Przykładem tego są Zakłady Mechaniczne w Tarnowie. Nowe kontrakty i zamówienia pozwoliły w ostatnich latach zwiększyć zatrudnienie w firmie o ok. 400 osób i zbudować pozycję zakładu jako kluczowego w Polsce przedsiębiorstwa obronnego. Obecnie zatrudnionych jest blisko 1000 osób. Tarnowskie Zakłady Mechaniczne obchodzą w tym roku 70-lecie uruchomienia produkcji zbrojeniowej. Obchodzą ten jubileusz w dobrej kondycji i z dobrymi perspektywami na przyszłość, choć firma z trudem przetrwała okres transformacji gospodarczej. Odbić się od dna pozwoliły właśnie nowe kontrakty i zamówienia. Mechaniczne” są m.in. liderem technicznym dużego projektu w pełni z epoki cyfrowej, polegającego na zbudowaniu i dostarczeniu dla polskiej armii sześciu przeciwlotniczych zestawów Pilica. Kontrakt ten jest największym zamówieniem realizowanym w całej historii działalności spółki. Obecnie firma oferuje szereg nowoczesnych konstrukcji, takich jak: karabiny wyborowe i maszynowe, działa do ostrzeliwania przeciwnika czy granatnika. W Tarnowie wyprodukowano już 650 kompletów moździerzy, którymi dysponuje praktycznie każda kompania lekkiej piechoty V rodzaju naszych Sił Zbrojnych. Podążanie za rozwojem techniki wojskowej umożliwia własne centrum badawczo-rozwojowe. Tarnowscy inżynierowie i konstruktorzy opracowują innowacyjne i konkurencyjne wyroby z kilku obszarów produktowych. Aktualnie pracują m.in. nad tym, aby na pole walki można było posyłać roboty zamiast ludzi. Temu celowi ma służyć np. Perun, autonomiczny pojazd kołowy z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych. Warto podkreślić, że Wojsko Polskie nie jest jedynym odbiorcą wyrobów z Tarnowa. Zakłady mechaniczne zajmują drugie miejsce na liście liderów eksportu wśród spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wielkim atutem jest bowiem niezawodność wyrobów. Ostatnio przedsiębiorstwo zyskało kolejny zagraniczny kontrakt, w którym kluczową rolę odegrały jakość oraz poziom wykonania dostarczonych do testów egzemplarzy. Pragnę też poinformować, że „Mechaniczne” produkują elementy do wyrzutni rakiet Patriot, które wchodzić będą w skład Wisły, programu obrony powietrznej kraju. Dziś, gdy widzimy tyle zagrożeń dla bezpieczeństwa naszego kraju, warto uświadomić sobie, jak ważne było uratowanie i utrzymanie przedsiębiorstwa produkującego uzbrojenie w oparciu o własną myśl techniczną. Kończąc, dziękuję również wszystkim pracownikom sektora zbrojeniowego w Polsce za profesjonalną, ofiarną i rzetelną pracę na rzecz obronności naszego kraju.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Chciałem z tego miejsca podziękować panu oraz ministrowi Dariuszowi Piontkowskiemu za dotowanie inwestycji województwa podlaskiego i prosić o niezaprzestawanie wspierania. Dziękuję wam za wspieranie rozwoju Podlasia. Środki przekazane w ostatnich latach na inwestycje mojego regionu są rekordowe. Nigdy przedtem województwo podlaskie nie miało takich pieniędzy i to trzeba powiedzieć bardzo głośno. O to dba marszałek województwa Artur Kosicki, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Im też z tego miejsca bardzo dziękuję. Wykorzystanie wsparcia widać niemal na każdym kroku. Rozwój województwa jest widoczny. Zmienia się krajobraz, infrastruktura, zmienia się jakość życia mieszkańców. Ten region staje się atrakcyjny pod względem życiowym, inwestycyjnym, coraz więcej młodych ludzi wybiera województwo podlaskie na miejsce swojego życia. To wszystko dzięki wam, ale wciąż potrzebujemy pieniędzy, by gonić lepiej rozwinięte regiony kraju, które wcześniej otrzymały większe pieniądze na rozwój. Każde pieniądze będą wydane najlepiej, jak można wydać, na polepszenie jakości życia mieszkańców. Pani poseł Joanna Frydrych, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przed nami nowy rok budżetowy. Najwyższy czas skierować środki finansowe tam, gdzie są naprawdę potrzebne. Najwyższy czas powstrzymać finansowanie propagandy rządowej i skierować te miliardy złotych na cele prospołeczne. Jako poseł z Podkarpacia zgłosiłam szereg poprawek do budżetu na 2022 r., tak aby środki mogły trafić do naszego pięknego województwa. I tak, kolejno poprawki dotyczą: w Krośnie - modernizacji drogi wojewódzkiej nr 991 Krosno - Lutcza, rewitalizacji linii kolejowej między Jasłem a Krosnem oraz obniżenia niwelety linii kolejowej nr 108 w Krośnie na odcinku 2 km, budowy łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie, budowy łącznika drogowego ul. Sikorskiego i ul. Bieszczadzkiej w Krośnie, budowy łącznika drogowego łączącego Krosno z drogą ekspresową S19, modernizacji sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie, uzbrojenia nowej strefy inwestycyjnej w Krośnie; w Przeworsku - dofinansowania rewitalizacji zespołu pałacowo parkowego; w Przemyślu - budowy ścieżek rowerowych i przystani wodnych nad rzeką San, budowy mostu na rzece San łączącego drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 884, rozbudowy budynków Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych o Audytoryjne Centrum Koncertowe; w Jarosławiu - dofinansowania inwestycji na terenach sportowo-rekreacyjnych nad Sanem, rozpoczęcia budowy mostu na rzece San; w Jaśle - budowy północnej obwodnicy Jasła od drogi krajowej nr 73 do Warzyc, bardzo ważnej inwestycji. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Każda ze złożonych poprawek ma na celu poprawę życia mieszkańców Podkarpacia.

Kolejne poprawki ważne dla rozwoju sportu i rekreacji dotyczą budowy ścieżek rowerowych i infrastruktury sportowej nad Sanem w Przemyślu i Jarosławiu. Mieszkańcy Podkarpacia zasługują na realizację tych inwestycji, zasługują na poparcie złożonych poprawek. Apeluję szczególnie do posłów z Podkarpacia: poprzyjcie złożone poprawki do budżetu na 2022 r. Jeszcze macie szansę, w najbliższy piątek odbędą się głosowania nad nimi. To są ważne inwestycje, które mogą zostać zrealizowane dla dobra mieszkańców naszego regionu. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu posłowie mają prawo do złożenia poprawek, które następnie są rozpatrywane przez Komisję Finansów Publicznych. Składane na tym etapie poprawki dotyczą głównie problemów regionalnych, których rozwiązanie jest oczekiwane przez społeczność, a często w wyniku tych problemów powstają bariery ograniczające rozwój regionów. Te poprawki opracowywane są z dużą precyzją i sztuką respektującą wszystkie zasady klasyfikacji budżetowej, a następnie są przekazywane do Biura Analiz Sejmowych. I na tym kończy się profesjonalizm i powaga działania. Niestety Komisja Finansów Publicznych nie dokonała ich przeglądu ani analizy. Wiele z nich po analizie można było skierować do poszczególnych ministerstw, by szukać rozwiązania umożliwiającego pomoc regionom, samorządom czy organizacjom społecznym. Nie zawsze chodzi przecież o pieniądze.

Wymienię niektóre z nich. Pierwsza grupa poprawek dotyczy barier rozwojowych i braku możliwości walki ze smogiem z powodu ograniczeń w dostawie gazu ze względu na niewydolność sieci przesyłowych. To jest zadanie PGNiG, ale odkładane w czasie. Takie miejscowości turystyczne jak Szklarska Poręba, Piechowice czy Wleń nie tylko nie mogą realizować zadań w zakresie budownictwa i rozwijać się ze względu na brak źródła ciepła, ale też nie mogą skutecznie walczyć ze smogiem, co jest na tym obszarze nakazem chwili.

Droga krajowa nr 30 w kierunku Zgorzelca i granicy państwa jest coraz bardziej obciążona ciężkim transportem towarowym, TIR-ami. Tymczasem ciągle odkładana jest budowa chodnika w miejscowości Chmieleń - o czym wielokrotnie mówiłam z tej mównicy - wzdłuż drogi krajowej nr 30.

Wnioskowałam o wsparcie finansowe budowy przedszkoli we Lwówku Śląskim, w Gryfowie Śląskim czy we Wleniu, a także o pomoc przy budowie szkoły podstawowej w Kowarach. To miasto poprzemysłowe, z wieloma problemami infrastrukturalnymi, i jedna z biedniejszych gmin pod względem dochodu na mieszkańca. Potrzebne jest także wsparcie samorządów w tworzeniu nowych bibliotek w małych miejscowościach. To niezwykle ważne, że samorządy chcą rozwijać sieć bibliotek. Pomóżmy im w tym szlachetnym działaniu.

Byłam przekonana, że takie zadania jak poprawa bezpieczeństwa w górach, kiedy w ostatnich latach masowo rośnie liczba turystów wędrujących szlakami górskimi, nie będą budziły wątpliwości i rząd znajdzie kilkaset tysięcy złotych na dofinansowanie budowy stacji ratunkowej GOPR w Karpaczu. Niestety nie ma. Bardzo przykra sprawa. Jak ja to powiem ratownikom górskim, którzy pracują społecznie?

Pytam: Kiedy nastąpi poprawa komunikacji?

Inaczej nie mogę powiedzieć ludziom w terenie. Apeluję, aby podczas głosowania w piątek jednak nastąpiła refleksja i posłowie z okręgu nr 1 poparli te poprawki. Wysoka Izbo! W tym roku 13 grudnia mija dokładnie 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, a jutro - 40 lat od pacyfikacji kopalni Wujek. Tarnogród, miasto w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim, to miejsce silnie powiązane z wydarzeniami w katowickiej Kopalni Węgla Kamiennego Wujek. To tu urodził się Józef Krzysztof Giza, jedna ze śmiertelnych ofiar krwawej pacyfikacji. Co roku w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w rodzinnej miejscowości Józefa Gizy odbywają się uroczystości upamiętniające to tragiczne wydarzenie. Zostały zaplanowane na 2 dni. 18 grudnia, w najbliższą sobotę, odbędzie się rekonstrukcja wydarzeń z grudnia 1981 r. oraz odtworzenie scen z życia codziennego w stanie wojennym przygotowane przez lokalną grupę rekonstrukcyjną, natomiast w sali widowiskowej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury odbędzie się projekcja filmu „Autor nieznany”, po której będzie można spotkać się z twórcami tego dokumentu. Film swoją premierę miał wczoraj w telewizji polskiej. Opowiada historię Jerzego Kośnika, fotoreportera, którego zdjęcia dokumentują najważniejsze wydarzenia lat 80., oraz Marka Janickiego, autora dramatycznych fotografii z krwawego tłumienia przez wojsko i milicję strajku w kopalni Wujek, który przez 30 lat, od grudnia 1981 r., ukrywał zdjęcia dokumentujące te tragiczne wydarzenia. Na zakończenie przewidziano koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego pt. „Odważnym wszystkim pokłon niski. Drugi dzień obchodów to zgodnie z tradycją uroczysta msza święta z udziałem górników, pocztów sztandarowych, parlamentarzystów i władz samorządowych, po której nastąpi złożenie kwiatów na grobie Józefa Krzysztofa Gizy. Kolejnym punktem uroczystości jest program patriotyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie, a także wręczenie nagród laureatom „Konkursu wojewódzkiego na projekt logotypu patriotycznego związanego ze stanem wojennym” Dzięki udostępnieniu zbiorów z zasobów Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności została również przygotowana wystawa pt. „Kopalnia strajkuje.

Wszystkich państwa, którzy chcieliby oddać hołd ofiarom stanu wojennego oraz wziąć udział w regionalnych uroczystościach, zapraszam do Tarnogrodu. Pani poseł Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pracujemy nad jedną z najważniejszych w roku ustaw, czyli ustawą budżetową. Od 2015 r., kiedy po raz pierwszy zostałam posłem, zabiegam o najważniejsze inwestycje w województwie pomorskim, w tym o obwodnicę Gardei. Z prośbą o wsparcie budowy tej obwodnicy zwrócili się do mnie mieszkańcy i władze gminy Gardeja, dlatego jest ona jednym z moich priorytetów. Ta obwodnica w śladzie drogi krajowej nr 55 odciążyłaby z ruchu tranzytowego całą gminę Gardeja. Złożyłam więc poprawkę do budżetu przyznającą 20 mln zł na rozpoczęcie prac projektowych, dokumentację i wykup gruntów pod budowę obwodnicy. Mieszkańcy i władze gminy Gardeja zabiegali o wpisanie swojej obwodnicy do rządowego projektu budowy 100 obwodnic w całej Polsce, ale niestety pomimo uzasadnionej potrzeby budowy tej obwodnicy rząd nie wpisał jej do tego programu. Mam nadzieję, że posłowie poprą moją poprawkę i mieszkańcy będą mogli się cieszyć z tej obwodnicy, chociaż mam co do tego wątpliwości, dlatego że już odbyło się głosowanie na posiedzeniu komisji finansów i nawet posłowie PiS z Pomorza nie poparli tej poprawki, choć jeszcze niedawno zapewniali, że chcą pomagać mieszkańcom i wspierać ich potrzeby. Słowa, słowa, słowa. Apeluję więc do rządu o przeznaczenie tej kwoty na tak ważną dla mieszkańców obwodnicę. Dziękuję. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

Wielkopolska Izba Rolnicza na walnym zgromadzeniu 26 października przyjęła stanowisko adresowane do władz publicznych, w tym do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W tym stanowisku podkreśla się przede wszystkim bardzo trudną sytuację na rynkach związanych z hodowlą zwłaszcza trzody chlewnej, z której Wielkopolska słynie.

Średnio rzecz biorąc, do produkcji jednego tucznika trzeba dopłacić 150 zł. Sytuacja dotyczy również warchlaków. Takich przypadków w ubiegłym roku w Polsce mieliśmy 110, a Wielkopolsce - 8.

Dotykają one również producentów, rolników, w szczególności jeśli chodzi o cenę nawozów azotowych.

Podobnie jeśli chodzi o inne nawozy - wzrost o 138 zł, o 62%. Tak że są rekordowe ceny nawozów, za tym idzie również wszystko to, co jest związane ze wzrostem cen energii, paliwa. Mimo że uchwaliliśmy kolejną nowelizację ustawy o dopłatach do paliw rolniczych, to oczywiście ta dopłata w żadnym stopniu nie nadąża za inflacją i za wzrostem cen paliw. Także bardzo wysokie są ceny produkcji i prowadzenia rozwoju gospodarstw, np. ceny materiałów budowlanych.

Po drugie, są instrumenty związane z tzw. tarczą osłonową, związane z inflacją. One też są kierowane do gospodarstw rodzinnych, ale w znacznej mierze nie pokrywają rzeczywistych wzrostów kosztów, cen towarów i usług. Dlatego też w imieniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej wspólnie z panem posłem Wiesławem Szczepańskim skierowaliśmy interpelację do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Mam nadzieję, że również w czasie tej debaty budżetowej i głosowań w najbliższy piątek panie i panowie posłowie wesprą działania, które są przygotowane zarówno przez stronę rządową, jak i kluby opozycyjne, i które mają na celu właśnie tę pomoc w dopłatach do zakupu nawozów mineralnych. Byłaby to istotna pomoc w prowadzeniu małych i średnich gospodarstw rolnych, które są konstytucyjną istotą naszego ustroju rolnego. Bardzo na to liczę. Pani poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przyznam, że nie chciałabym, żeby po moim wystąpieniu został tylko ślad w stenogramie. Chciałabym, żeby temat, który poruszę, był przedmiotem debaty.

To był piękny dzień, a to już tyle lat - 19 lat temu.

Nie uczestniczyłam w tym wydarzeniu z oczywistych powodów - obowiązki poselskie nie pozwoliły mi pojechać do Gdyni - ale to naprawdę trudny i smutny dzień, bo właściwie trzeba uczciwie powiedzieć, że pożegnaliśmy swoje okręty podwodne.

Musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Wiem, że wczoraj kilkadziesiąt osób uczestniczyło w tym pożegnaniu, w tym ostatnim opuszczeniu bandery.

Nie ma debaty na ten temat. Naprawdę gorąco apeluję, żebyśmy to zrobili, tym bardziej że, jak mówię, słucham nie byle jakich dyskutantów, tylko słucham marynarzy, którzy całe życie służyli w Marynarce Wojennej. Musimy pamiętać, że Marynarka Wojenna jest nam potrzebna i okręty podwodne są nam potrzebne. Bo to nie jest tylko tak, że jest nam potrzebna tarcza w postaci fregaty. Nam jest również potrzebny miecz w postaci okrętu podwodnego. Broń ofensywna to też obrona. Stąd mój szczery apel o to, żeby taka debata się odbyła.

Nie chciałabym, żeby tak się zakończyła historia okrętów podwodnych w naszym kraju. Po raz kolejny powtarzam: marynarze uważają, że okręty podwodne są nam bardzo potrzebne. Apeluję, bo to jest nasz wspólny interes, nie mój, nie pojedynczych posłów, tylko naszego państwa, obywateli naszego kraju, żeby dobrze, mądrze wszystko przygotować i żeby jak najszybciej okręty podwodne wróciły do naszego kraju. Chciałabym bardzo - po raz kolejny to podkreślam - żeby ten temat był bardzo poważnie przez wszystkich potraktowany, a przede wszystkim przez rządzących, to jest oczywiste. Ale pamiętajmy o tym, że to nie są tylko takie sobie opowieści, to jest coś ważnego dla naszego bezpieczeństwa. Gorąco o to apeluję. Pan poseł Waldemar Andzel, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 22 czołgi, 44 wozy bojowe, 760 żołnierzy i 1400 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i ZOMO - przy udziale takich sił przeprowadzono masakrę katowickiej kopalni Wujek i strajkujących górników. Od godz. 8 rano pacyfikacja postępowała. Milicja otoczyła kopalnię, użyto armatek wodnych i gazu. O godz. 12.30 skierowano do kopalni specjalny pluton ZOMO, finalnie zamordowano wtedy dziewięciu górników. Zomowcy użyli pistoletów maszynowych. Strajk zakończył się tego samego dnia. Dowódca plutonu Romuald Cieślak po 27 latach został skazany na 6 lat pozbawienia wolności. Wyroki usłyszeli też jego podkomendni. Za zbrodnie nigdy nie odpowiedzieli towarzysze Kiszczak i Jaruzelski. 2 lata temu Chorwacja wydała Polsce Romana S., kolejnego milicjanta z plutonu specjalnego ZOMO poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Cześć pamięci zamordowanych górników!

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W naszej historii nie brakuje tragicznych wydarzeń, które budzą dzisiaj wiele emocji. Jednym z nich jest wprowadzenie stanu wojennego. Grudzień to miesiąc wyjątkowy, w którym pamięcią sięgamy do tragicznych i smutnych wydarzeń z 1981 r. Wprowadzony stan wojenny, którego kolejną rocznicę obchodziliśmy 13 grudnia, był przejawem bezradności i strachu komunistycznej władzy wobec rosnącej siły „Solidarności” Okupiony został on jednak tragicznie, ofiarami. Jak kiedyś powiedział św. Jan Paweł II, „Solidarność” to nigdy jeden przeciwko drugiemu, ale zawsze jeden razem z drugim. Tej zasadzie byli zawsze wierni śląscy górnicy, którzy stawili największy opór w kraju przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.

Władze, nie godząc się na żadne ustępstwa, zdecydowały się użyć siły wobec górników stanowczo odmawiających przerwania strajku. 16 grudnia doszło do największej tragedii stanu wojennego. Oddziały wojska i ZOMO przez obalony czołgami mur wtargnęły na teren kopalni. W wyniku otwarcia ognia do bezbronnych cywilów na miejscu zginęło sześć osób, a trzy kolejne zmarły później w szpitalu.

Przed pierwszą zmianą w kopalni Manifest Lipcowy członkowie Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” zorganizowali masówkę. W cechowni znajdowało się ok. 2 tys. osób.

Ok. godz. 9 dotarła wiadomość o brutalnej rozprawie z górnikami w kopalni Jastrzębie, a o godz. 11 przed kopalnię Manifest Lipcowy przyjechały oddziały milicji i wojska. W kierunku strajkujących rzucano petardy i pojemniki z gazem łzawiącym. Ok. godz. 11.45 na teren zakładu wkroczył specjalny pluton ZOMO uzbrojony w broń palną i amunicję. Gdy górnicy ruszyli do przodu, padły pierwsze strzały w stanie wojennym. Ranni zostali: Franciszek Gąsiorowski, Czesław Kłosek, Zdzisław Kraszewski, Bogusław Tomaszewski. Postrzelonych przewieziono do szpitala, na szczęście nikt nie zmarł. Przywódców strajku: Jana Bożka, Józefa Błauta, Waldemara Macieszka, Eugeniusza Zandlera aresztowano pod koniec roku lub na początku nowego. Brutalne ataki na protestujących w kopalni Manifest Lipcowy opisuje na stronach serwis Pamięć Jastrzębska. Ówczesny przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Jan Bożyk pisze: Wreszcie podjechali czołgami i wozami pancernymi pod bramę, ktoś mówił coś przez megafon, ale wycie silników zagłuszało jego głos. Ludzie śpiewali „Jeszcze Polska nie zginęła”, „Boże coś Polskę” Na plac poleciały świece dymne i gazowe. Gaz miał nieprzyjemny zapach i szczypał w oczy. Ludzie parli do przodu. Stojąc na czele, próbowałem ich powstrzymać. ZOMO-wcy wycofali się z kopalni przez bramę towarową lub przez osobową. Próbowaliśmy z Maciaszkiem, Błautem i Zandlerem zatrzymać załogę, żeby nie doszło do bezpośredniego starcia.

Tak padły pierwsze strzały stanu wojennego.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dziękujemy za to, że znaleźli się odważni ludzie, dla których wiara w ideały okazała się ważniejsza od strachu napędzonego przez komunistyczny reżim, który i tak upadł.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na moje dyżury poselskie trafia wiele osób poszkodowanych przez tzw. mafię mieszkaniową. Są to zazwyczaj osoby starsze, nieposiadające zdolności kredytowej, które w pewnym momencie swojego życia zmuszone zostały do poszukiwania pomocy finansowej chociażby ze względu na to, aby znaleźć środki na operację. Ponieważ banki nie chciały lub nie mogły tym osobom udzielić kredytu lub pożyczki, odzywały się do nich różne podmioty, które z chęcią udzielały wysokich pożyczek, ale w zamian za przekazanie własności domu, mieszkania czy gospodarstwa rolnego aż do czasu spłacenia takiej pożyczki. Brak spłaty wiązać się miał z utratą własności mieszkania i w ten sposób za pożyczenie 50 tys. zł pożyczkobiorca oddawał mafii mieszkaniowej nie tylko pieniądze, ale także swój majątek idący niejednokrotnie w setki, a nawet w miliony złotych. W procederze tym oprócz wyspecjalizowanych przestępców brali udział notariusze, którzy przygotowywali akty notarialne. Akty te albo nie były odczytywane, albo odczytywane w taki sposób, aby pożyczkobiorca nie zorientował się, że traci cały swój majątek. Domy, mieszkania czy gospodarstwa rolne przestępcy szybko starali się zbyć, tak aby utrudnić ich odzyskanie. Rozkwit tego typu działań przestępczych miał miejsce po zmianach, jakie wprowadzono za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Stowarzyszenie 304 KK, które założyli poszkodowani przez mafię mieszkaniową i które zajmuje się tropieniem tego typu przestępstw, stworzyło nawet mapę przestępców gospodarczych z całej Polski i współpracujących z nimi notariuszy. W zeszłej kadencji powstał Zespół Parlamentarny ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy. Okazało się, że tego typu przestępczą działalnością zajmują się nie tylko ludzie z parabanków czy firm finansowych nastawionych na szybki zysk, ale także sędziowie, którzy udzielali pożyczek na wysoki procent, przewyższający odsetki dopuszczone ustawą, a potem szantażowali pożyczkobiorców. Jakiś czas temu udało się zmienić przepisy w taki sposób, że notariusze nie mają możliwości tworzyć aktów notarialnych, których celem jest dokonanie pożyczki na tzw. przewłaszczenie. Wiem, że rząd, a szczególnie Ministerstwo Finansów, zamierza uszczelnić te przepisy jeszcze bardziej, dzięki czemu liczba poszkodowanych spadnie. W wielu miejscach udało się rozbić mafię mieszkaniową, czego przykładem jest sytuacja z Gdańska.

Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.